Ta konstrukcja funkcjonuje już od jakiegoś czasu. To są właśnie środki przekazane na leki 75+. Nikt nie zaniechał tego projektu. Co więcej, te nakłady sukcesywnie rosną.

To pokazuje, jak istotnie te środki rosną, praktycznie o 200 mln w 2 lata, a jak zaczynaliśmy ten program, były na poziomie ok. 600 mln zł. Pan poseł pytał również o fundusz modernizacji szpitali. Ta ustawa, o której przed chwilą wspominałem, która weszła w życie, ten fundusz określa i stanowi o obowiązkach ministra zdrowia w związku z tym funduszem. My już w najbliższym czasie przedstawimy Radzie Ministrów założenia szczegółowe odnośnie do tego funduszu i w ramach utartej ścieżki, przyjętego programu wieloletniego, mam nadzieję, że przez Radę Ministrów niedługo ten fundusz zostanie przyjęty i to wsparcie dla szpitali w Polsce zostanie skierowane. Pan poseł Szczerba sam wspominał o tym, że to niekończąca się historia - program alzheimerowski. Ja wiele razy z tej mównicy odpowiadałem, dlaczego ten program w formule programu polityki zdrowotnej nie ma sensu, dlaczego nie ma podstaw do takiego finansowania programu, o który pan poseł pytał. Pytał pan również w zapytaniach pisemnych. Natomiast, mam nadzieję, dobra informacja nie tylko dla pana posła, ale dla wielu osób chorych na choroby otępienne. My w ramach negocjacji z Komisją Europejską, w ramach przygotowywania kolejnej perspektywy unijnej dyskutujemy (Dzwonek) o możliwości wsparcia właśnie chorych na choroby otępienne w zakresie utworzenia pewnych dziennych form pomocy, dziennych domów wsparcia pamięci.

Wracam do tego. Te świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jeżeli tylko pan poseł wyrazi takie oczekiwanie, to ja chętnie na forum podkomisji, zespołu chyba akurat w tym przypadku, rzeczywiście wspólnie gotów jestem zastanowić się nad pewnymi rozwiązaniami rozszerzającymi, szczególnie że jesteśmy w przededniu tak naprawdę pokazania publicznie planu odbudowy zdrowia Polaków, o którym mówił pan minister Niedzielski. Tam jednym z bardzo ważnych filarów są badania profilaktyczne, w różnym obszarze, oczywiście istotne z punktu widzenia onkologii, ale nie tylko, bo chociażby pewien program profilaktyczny dla Polaków w wieku 40+ również zostanie zaprezentowany. Jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pani poseł Hennig-Kloska odnosiła się do podatku cukrowego. Apeluję chyba do wszystkich parlamentarzystów: nie używajmy argumentu, że dziecko w sklepie nie kupi już trzech soczków, tylko dwa. To bardzo dobrze dla zdrowia naszych dzieci i dla zdrowia młodych Polaków. Niech kupią wodę. Niech kupią wodę niesłodzoną, niech zrezygnują z zakupu dwóch soczków i niech ten podatek cukrowy wymusi właśnie takie działania. Możemy nie pić napojów słodzonych. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę teraz pana Andrzeja Bittela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, o udzielenie odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To w mojej ocenie świadczy o tym, że budżet, który został zaplanowany w tej dziedzinie, jest bardzo dobry. To zdanie podziela również Komisja Infrastruktury, a wypowiedzi koreferenta budżetowego pana ministra Grabarczyka, posła Grabarczyka, też o tym świadczą, że budżet na rok 2021 jest budżetem niezwykle interesującym, bardzo dobrym, na dodatek zrównoważonym pomiędzy sektorem drogowym a sektorem kolejowym. Starając się odpowiedzieć na tych kilka pytań, które padły, z których niektóre są pozabudżetowe.

Było pytanie o modernizację dworca Poznań Główny. PKP SA szykuje razem z miastem Poznań konkurs architektoniczny, urbanistyczny, tak aby ta inwestycja jak najlepiej odpowiadała potrzebom mieszkańców aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskiego i całej Polski, bo to ważne miejsce na mapie kolejowej.

Ta inwestycja - most - jest realizowana w ramach programu rządowego „Mosty dla regionów”

S14 znajduje się w budowie, w dwóch odcinkach, na oba zostały podpisane umowy z wykonawcami.

Tu można powiedzieć, że po wielu trudach - a te trudy opierają się, polegają na pełnym procesie odwoławczym od decyzji środowiskowej - ta decyzja już jest. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowa.

Jeśli coś pominąłem, postaram się odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę teraz pana Ryszarda Bartosika, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o zabranie głosu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie! Pytania do ministra rolnictwa dotyczyły m.in. wydatkowania środków budżetowych. Było pytanie: Dlaczego nakłady na rolnictwo spadają od 2015 r. Otóż chciałem chyba po raz kolejny Wysoką Izbę poinformować, że nakłady na rolnictwo od tego czasu znacznie wzrosły, a w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z budżetu krajowego, łącznie z wydatkami na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wynoszą 28 960 784 tys. zł i będą wyższe w porównaniu z ustawą budżetową na rok bieżący. Zwiększone zostały również wydatki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych i zwierząt gospodarskich, zostały także zwiększone wydatki na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o kwotę 120 tys. zł, na KRUS, na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na funkcjonowanie szkół rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego. Ogółem wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wzrastają w ustawie budżetowej w stosunku do roku bieżącego o 11,51%. Wysoka Izbo! Mówimy tu o wydatkach stricte na rolnictwo i sektor rolniczy, ale w tym miejscu trzeba powiedzieć o środkach, z jakich korzysta i będzie korzystała polska wieś, środkach, które też mają ogromny wpływ na komfort życia na wsi, na rozwój środowisk rolniczych. Chcę tutaj powiedzieć również o środkach, które zostają przekazane na ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, Fundusz Dróg Samorządowych. Wszystkie te działania realizowane są oczywiście poza ministerstwem rolnictwa, ale mają ogromny, znaczący wpływ na życie na wsi. W ostatnim czasie - i warto też to przy okazji ustawy budżetowej powiedzieć - ministerstwo rolnictwa wprowadziło program: komputer dla rodziny. Ten program będzie niebawem realizowany. Nabór prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Prowadzimy także wsparcie dla producentów trzody chlewnej. Ten program również jest w tej chwili w realizacji. Szanowni Państwo! Warto też wspomnieć, że takie środki jak środki z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również trafiają na wieś. Są to podwyżki emerytur, trzynasta emerytura, ale także wsparcie rodzin rolniczych w czasie pandemii. Rodzice opiekujący się małymi dziećmi otrzymują wsparcie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Oprócz działań nakierowanych stricte na rolnictwo, jak widzimy, wsparcie jest dużo, dużo szersze i ogromny strumień pieniędzy wpływa do rolników. Nie wspomniałem jeszcze o pomocy COVID-owej, która w ramach poszczególnych tarcz również trafia do rolników. Szanowni Państwo! Na resztę pytań odpowiem pisemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Kolejna osoba odpowiadająca na pytania to pan Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Bardzo proszę.

Szanowny Panie Marszałku! Postaram się zbiorczo odpowiedzieć na pytania zadawane przez państwa posłów. Dużo pytań dotyczyło funduszu inwestycji lokalnych. Chciałbym zwrócić uwagę, że państwo odnosili się tylko do części podziału ponad 4 mld, które zostały podzielone przez międzyresortowy zespół. Koledzy posłowie, możecie troszkę ciszej rozmawiać?

Padło również pytanie o kwestie związane z wydatkami niewygasającymi. Pracujemy nad rozporządzeniem Rady Ministrów i do końca tego miesiąca to rozporządzenie będzie wydane. Proszę bardzo o zaprzestanie rozmów i umożliwienie udzielenia odpowiedzi panu ministrowi.

W zakresie jednostek samorządu terytorialnego i ich dochodów zwracam uwagę na wzrost subwencji ogólnej do kwoty ponad 70 mld, czyli o ponad 5%, w tym subwencji tzw. części oświatowej o ponad 2,2 mld. Padło również pytanie o brak środków na trzynastą emeryturę. Te środki będą zapewnione i wypłata trzynastej emerytury nie jest zadłużona. Jeżeli chodzi o kwestię podatków i opłat, to zwracam uwagę, że estoński CIT jest rozwiązaniem systemowym proinwestycyjnym. Szacujemy z tego tytułu nawet ubytki w podatku w sektorze finansów publicznych.

Część tej opłaty będzie trafiać do Narodowego Funduszu Zdrowia, a część do jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie państwowego długu publicznego już dziś mogę powiedzieć, że nasze ostatnie szacunki pokazują, że dług w ujęciu general government, czyli unijnym, nie przekroczy w tym roku 60% PKB.

Mówię o roku bieżącym, czyli roku 2020.

Nie myślimy o całkowitej likwidacji janosikowego, ale myślimy o takim rozwiązaniu, które umożliwiłoby jego spłaszczenie, tzn. żeby wpłata janosikowego była na poziomie stabilnym i antycyklicznym.

Pan nie zrozumiał tego, o czym mówiłam. To nie jest tak - i pan dobrze o tym wie - że dochody z VAT wyższe, niż założyliście w nowelizacji, przekładają się na zmniejszenie luki VAT-owskiej. Odnoszę się do luki VAT-owskiej.

Chwalił się pan tutaj, że Komisja Europejska szacuje, że w tym roku nasz dług nie przekroczy 60% według ich metodologii, ale nie odpowiedział pan na moje pytanie o to, co z inflacją.

Bo jeśli manipulujecie inflacją po to, żeby obniżyć sobie dług publiczny w relacji do PKB, to płacą za to najbiedniejsi Polacy, o czym pan dobrze wie. Nie powiedział pan też nic o stopach procentowych i wysokiej inflacji. Powiedziałam: stopy procentowe europejskie, inflacja polska, nie odniósł się pan do tego w ogóle. Być może będzie na to szansa w wypowiedzi pana posła Henryka Kowalczyka, sprawozdawcy komisji, którego bardzo serdecznie zapraszam.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nie będę tego powtarzał.

To za waszych rządów wasz kolega, prof. Balcerowicz, zainstalował licznik długu publicznego w centrum Warszawy i to wtedy właśnie był ten kryzys.

Natomiast akurat w tym roku będzie zwiększenie długu, bo jest ogromny kryzys, bo trzeba ratować przedsiębiorców - zresztą bardzo skutecznie, bo bezrobocie praktycznie nie wzrosło.

Kilkaset poprawek naprawdę nie zakrzyczy tego budżetu, natomiast pozbawia szansy. Rzeczywiście, gdyby poprawki były merytoryczne, było ich kilkanaście czy kilkadziesiąt, można by się było nad nimi zastanawiać. Natomiast brak tej odpowiedzialności zarówno w czasie prac komisji nad ilością poprawek, jak i niestety dzisiaj, w trakcie drugiego czytania. Ale są niestety kluby, które takich poprawek złożyły kilkaset.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy wniosek o odrzucenie i poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rezerwach strategicznych (druk nr 829)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy o rezerwach strategicznych. Obowiązująca aktualnie ustawa o rezerwach strategicznych nie zawiera dostatecznego poziomu regulacji dających możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze rezerw strategicznych w kontekście dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami. Pandemia COVID-19 wskazała na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych. Zmiany te, od procesu tworzenia rezerw strategicznych zarówno w ramach Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, jak i poza nim, przez zadania agencji i ich finansowanie, aż po kwestie związane z dystrybucją rezerw, determinowane są pilną potrzebą lepszego i sprawniejszego reagowania na zagrożenia, zwłaszcza te, które trudno przewidzieć i w krótkiej, i w długiej perspektywie czasu. Obecnie tworzenie rezerw, jak również ich udostępnianie następuje wyłącznie w oparciu o decyzje centralnych organów administracji rządowej. Powoduje to m.in. wydłużenie procesów, których szybkie przeprowadzenie, nawet z godziny na godzinę, może być wymagane w niektórych sytuacjach kryzysowych. Agencja Rezerw Materiałowych nie uczestniczy w tworzeniu Rządowego Programu Rezerw Strategicznych. Brak też w tym procesie innych jednostek niższego szczebla działających w obszarze zarządzania kryzysowego, tj. Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i innych organów administracji rządowej oraz służb, inspekcji i innych jednostek realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego, w tym sprawujących na mocy ustaw nadzoru nad realizacją tych zadań wykonywanych przez przedsiębiorców. Brak głosu ww. jednostek w procesie planowania i programowania prowadzi do niedostatecznego sprecyzowania potrzeb co do zakresu i ilości utrzymywanych rezerw strategicznych. Kolejnym istotnym problemem na gruncie obecnych przepisów jest brak w obecnym stanie prawnym właściwych narzędzi dających możliwości szerokiej dystrybucji rezerw przez agencję, tak aby przy użyciu pozostających w jej dyspozycji zasobów logistycznych docierać z nimi szybko i sprawnie do odbiorców końcowych. Proces udostępniania rezerw strategicznych odbiorcy końcowemu jest skomplikowany i wielowymiarowy. Zgodnie z przepisami odbiorcy muszą we własnym zakresie organizować transport, co znacząco utrudnia efektywne wykorzystanie udostępnionych rezerw. W obecnym stanie prawnym ograniczona pozostaje również możliwość efektywnego wykorzystywania zasobów stanowiących rezerwy strategiczne, które mogą podlegać zwrotowi, tak aby ograniczać koszty ich utrzymywania oraz realizować zadania istotne społeczne w czasie, kiedy nie występuje żadna sytuacja kryzysowa. Wysoka Izbo! Na mocy nowej ustawy o rezerwach strategicznych system rezerw strategicznych zostanie znacząco przebudowany. Celem tej zmiany będzie bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie niektórych towarów i dóbr na rynku, a tym samym - negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli. Biorąc pod uwagę konieczność uproszczenia procedur, a co za tym idzie - zwiększenia skuteczności i podniesienia efektywności działań Agencji Rezerw Materiałowych, wprowadzone zostaną nowe instytucje prawne zapewniające realizację tych celów, inne zaś zostaną znacząco zmodyfikowane. Prezes Rady Ministrów stanie się organem bezpośrednio nadzorującym system rezerw strategicznych, co pozwoli na najbardziej skuteczne zarządzanie nimi. Jest to uzasadnione, gdyż nawet w dotychczasowym układzie w systemie rezerw znajdują się towary z obszaru właściwości różnych działów administracji rządowej. W konsekwencji tego z uwagi na rolę i funkcję agencji w systemie zarządzania kryzysowego będzie ona nadzorowana przez prezesa Rady Ministrów. Zostanie ulepszony proces tworzenia rezerw strategicznych w ramach Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, a także ich przechowywania, tak aby lepiej odpowiadały potrzebom bezpieczeństwa RP. W tym celu rozszerzono zakres zadań, dla których wsparcia tworzone są rezerwy strategiczne. Stworzono nowe instytucje prawne, które dotyczą, po pierwsze, udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu technicznego odpłatnie lub nieodpłatnie, co będzie mieć na celu zwiększenie efektywności wykorzystania asortymentu rezerw, w szczególności optymalizację kosztów związanych z utrzymywaniem rezerw oraz odpowiednio wsparcia realizacji celu ochrony zdrowia lub celów społecznych, a po drugie, możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów o tzw. pozostawaniu w gotowości zawieranych przez agencję z określonymi podmiotami w przedmiocie utrzymywania zdolności produkcyjnych lub umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia określonych usług na potrzeby rezerw strategicznych, zapewniając tym samym większą dostępność rezerw i ograniczając problemy z zakłóceniami w łańcuchach dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Asortyment i ilość rezerw będzie określał, tak jak dotychczas, „Rządowy program rezerw strategicznych”, który będzie opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z agencją na okres 5 lat. W projekcie ustawy rozszerza się zakres zadań dla wsparcia realizacji których tworzone są rezerwy strategiczne. Dodano zadania z zakresu realizacji interesów narodowych RP oraz z zakresu udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. Poszerzenie celu tworzenia rezerw w zakresie międzynarodowym o podmioty prawa międzynarodowego publicznego umożliwi udzielanie wsparcia nie tylko państwom, ale także organizacjom międzynarodowym. W ten sposób zostanie osiągnięty efekt uelastycznienia w zakresie udzielania przez Polskę pomocy międzynarodowej. Utrzymane zostaną dotychczasowe zadania agencji z jednoczesnym znacznym poszerzeniem ich katalogu. Po pierwsze, wprowadzone zostaną nowe zadania dla agencji w zakresie organizowania usług, w tym usług transportowo-logistycznych na własną rzecz oraz na rzecz innych organów lub podmiotów realizujących działania wspierające zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, wypełnienia zobowiązań międzynarodowych i realizacji interesów narodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia innym państwom i organizacjom międzynarodowym. Celem wprowadzenia nowej kompetencji agencji jest potrzeba większego jej zaangażowania w proces udostępniania rezerw strategicznych i większego wykorzystania zasobów, w tym zasobów ludzkich, a także podniesienie efektywności procesu udostępniania asortymentów, w tym w szczególności skrócenie czasu jego dostarczania do odbiorcy końcowego. Kolejnym nowym zadaniem ma być zadanie w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność lub pozostającymi w posiadaniu agencji lub świadczenia innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Celem tej kompetencji jest optymalizacja wykorzystania nieruchomości będących własnością agencji, możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań agencji oraz na jej funkcjonowanie w wyniku efektywnego wykorzystywania tych nieruchomości. W przypadkach, w których agencja nie wykorzystuje magazynów rezerw strategicznych do przechowywania w nich rezerw, powstaje możliwość wykorzystania ich na cele komercyjne poprzez umowy najmu czy dzierżawy. Projekt usprawnia i optymalizuje likwidację rezerw, tzn. poszerza sposoby likwidacji rezerw oraz poszerza katalog podmiotów, którym agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwidowanych rezerw. Będą nimi podmioty, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu. Takie rozwiązanie będzie dawało możliwość wsparcia podmiotów realizujących ważne społecznie cele uzasadniające nieodpłatne przekazanie. Wraz z nową ustawą wprowadzona będzie zmiana nazwy agencji. Dotychczasową nazwę „Agencja Rezerw Materiałowych” zastąpi nazwa „Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych” Zmiana nazwy jest nie tylko zabiegiem semantycznym, ale ma na celu odzwierciedlenie rzeczywistego zakresu zadań i kompetencji agencji. Jednym z założeń ustawy jest wprowadzenie zmiany w przepisach regulujących zasady zatrudniania w agencji. W projekcie ustawy podniesiono poziom wymagań w zakresie dotychczasowego doświadczenia zawodowego dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku prezesa oraz zastępcy prezesa agencji. Zgodnie z projektowanymi regulacjami osoba taka niezależnie od innych wymagań musi posiadać co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma pozostać agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wysoka Izbo! Projekt ustawy o rezerwach strategicznych przedłożony Wysokiemu Sejmowi przez Radę Ministrów wpisuje się w całościową politykę państwa, która wyciąga wnioski z sytuacji kryzysowych, w tym przede wszystkim z obecnie trwającej naszej wspólnej walki z epidemią koronawirusa. Wyrażam nadzieję, że zawarte w projekcie zmiany i nowe rozwiązania będą stanowiły znaczące wsparcie i ułatwienie w funkcjonowaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a przez to wpiszą się w proces zmian w systemie zarządzania kryzysowego państwa polskiego. Uprzejmie proszę panie i panów posłów o przyjęcie zaproponowanego projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Proszę pana posła Rafała Bochenka, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Nie widzę. Zatem zapraszam pana posła Sławomira Neumanna, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jakie wnioski wyciągnęliście, składając tę ustawę, z walki z koronawirusem? Składacie ustawę, która ma poprawić chaos i bałagan, który dzisiaj jest w Agencji Rezerw Materiałowych, ale tą ustawą wprowadzacie jeszcze większy chaos. Na początek tylko jedno pytanie związane z koronawirusem: Ile do dzisiaj Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła lodówek, które mogłyby przechowywać te szczepionki Pfizera? Mam pytanie: Czy agencja, która powinna być odpowiedzialna za przygotowanie tej całej infrastruktury, zakupiła choć jedną taką lodówkę, żeby przekazać ją do małej przychodni na wsi, żeby można było tam szczepić ludzi, Polaków? Czy zamiast tego zajmujecie się wyłącznie przygotowaniem ustawy, która ma znowu zmienić nazwę agencji, która nie dała sobie rady w trudnej sytuacji? Po co tak szybko? Po co w tej chwili? Po co w momencie, kiedy toczy się walka z koronawirusem, kiedy wiadomo było, że nie dajecie sobie rady? Agencja nie dała sobie rady w lutym czy w marcu przygotować się na koronawirusa, mimo że świat już o tym wiedział. Mimo że zakupy w wielu krajach były robione, w Polsce tego nie robiliśmy. Potem przyszły czasy miesięcy wakacyjnych. Premier ogłaszał zwycięstwo z epidemią. Znowu nic nie kupowaliśmy. Znowu się okazało, że agencja jest niepotrzebna, bo premier zlecił zakup maseczek, respiratorów czy innego sprzętu spółkom Skarbu Państwa. Po co taka agencja? Potem jeszcze premier witał wielki samolot, który przyleciał ze sprzętem do niczego się nienadającym. Dzisiaj chcecie tę agencję zmienić w agencję podległą premierowi, jakby do tej pory premier nie podejmował decyzji, jakby do tej pory premier nie pojawiał się w magazynach agencji, na tle przenoszonych pudeł i kartonów, pokazując, jak ta agencja świetnie działa.

Czy remedium na takie działanie jest nowa ustawa, która wprowadzi jeszcze większy bałagan? Czy nie wynika z tego, że tam pracują po prostu niekompetentni ludzie, którzy nie są w stanie dokonać racjonalnych zakupów, nie są w stanie podejmować decyzji? Czy nie lepiej od środka to poprawiać, niż zmieniać nazwę czy zmieniać podporządkowanie?

A przypomnę, że z waszego własnego uzasadnienia widać, że z agencją współpracuje 15 tys. aktywnych kontrahentów, 84 tys. przedsiębiorców zaangażowanych jest w utrzymanie rezerw strategicznych, ok. 1 tys. jednostek Policji, Straży Granicznej czy straży pożarnej, plus samorządy: województwa, powiaty, gminy. Nikt ich nie pytał o zdanie, a oni z wami współpracują. Dlaczego tak szybko i dlaczego w takim momencie, kiedy jest kryzys i kiedy należy raczej uspokajać i sobie z tym radzić w sposób bardziej zorganizowany, jeszcze wprowadzacie zmianę?

Nie macie w pamięci tego, co zrobiliście z BOR-em? Zmieniliście ustawę o Biurze Ochrony Rządu, żeby zmienić je na Służbę Ochrony Państwa, bo były dzwony na ulicach. Nie, bo to nie chodzi o nazwę, tylko chodzi o ludzi tam pracujących i ich kompetencje. Argument za tą centralizacją, tym podciągnięciem tego wszystkiego pod premiera. Przecież w lutym, zamiast dostarczyć do szpitali środki ochrony osobistej dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu, nie mogliście tego zrobić, bo agencja była zawalona węglem, który na wniosek z rządu i premiera agencja musiała kupić, nie po to żeby tworzyć rezerwę strategiczną, tylko po to żeby pomóc kopalniom. Wy nie rozumiecie w ogóle, po co taka agencja jest, i żeby przykryć ten swój własny bałagan, tworzycie nową ustawę. Ta ustawa nic nowego nie wnosi poza kolejnym bałaganem w agencji, która już sobie nie daje rady. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o te konsultacje, których zabrakło, ten pośpiech, który był w rządzie, da się to naprawić w Sejmie i przynajmniej w Sejmie będziemy mogli chwilę nad tym popracować i popytać wszystkich interesariuszy tej ustawy o ich zdanie, bo tego wyście nie zrobili. Dziękuję bardzo. W imieniu klubu parlamentarnego Lewica stanowisko przedstawi pan poseł Wiesław Szczepański. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko odnośnie do projektu ustawy o rezerwach strategicznych, zawartego w druku nr 829. Projekt wpłynął do Sejmu 9 grudnia br., ale do projektu nie załączono żadnych opinii ani ekspertyz, a z uzasadnienia wynika, że nie przewiduje się poddania projektu konsultacjom publicznym z uwagi na konieczność pilnego procedowania nad nim w związku z COVID-em oraz pilną potrzebą jego uchwalenia. Działania rządu, tak jak zawsze, przypominają mi bajkę o pomysłowym Dobromirze, któremu kuleczka lata nad głową, coś pomyślał, a więc wpadł na pomysł, a rząd to przygotował i Sejm musi to błyskawicznie uchwalić. Według projektu zmieni się nie tylko nazwa Agencji Rezerw Materiałowych, ale również zasady jej działania. Wprowadza się możliwość odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego. Powstała w wyniku przekształcenia Agencji Rezerw Materiałowych Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podlegać będzie teraz bezpośrednio premierowi, a nie, jak poprzednio, ministrowi właściwemu do spraw klimatu. Projektowana ustawa reguluje zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych, a także zasady ich finansowania. Rozbudowany zostanie również zakres zadań realizowanych przez agencję rezerw strategicznych. Rząd chce poprawić proces tworzenia i przechowywania rezerw strategicznych, tak aby lepiej odpowiadały potrzebom państwa. Zmiana też zaproponowana została w wyniku doświadczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanymi nią niedoborami asortymentu medycznego. Jako przykład należałoby podać brak maseczek ochronnych, rękawiczek, respiratorów, kiedy wiadomo było już, że w Chinach grasuje COVID.

Nie mówię już o kilkuset milionach złotych, które utopiono w węglu dzisiaj leżącym na hałdach. W projekcie ustawy zawarto nowe rozwiązania prawne przewidujące możliwość udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu technicznego odpłatnie lub nieodpłatnie. Myślę, że może to dotyczyć również tych respiratorów zakupionych od handlarza bronią, które dzisiaj leżą i nie są wydawane. Pojawia się nowa definicja dotycząca specjalistycznego asortymentu medycznego rezerw strategicznych. Asortyment ten obejmuje maszyny, urządzenia i inne przedmioty wykorzystywane do celów związanych z ochroną zdrowia. Zgodnie z ustawą premier będzie upoważniony do odpłatnego udostępniania państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego. Czy można prosić o umożliwienie spokojnego wystąpienia panu posłowi? sprzętu specjalistycznego, medycznego stanowiącego część rezerw strategicznych w warunkach innych niż sytuacja kryzysowa na zadania związane z ochroną zdrowia. Ma to zoptymalizować koszty utrzymania tych rezerw i ich wykorzystania. Ustawa przewiduje również utrzymanie rezerw strategicznych na podstawie umów zawieranych przez agencje o pozostawaniu w gotowości do utrzymania zdolności produkcyjnych lub świadczenia określonych usług na potrzeby rezerw strategicznych.

Mój klub opowiada się za skierowaniem tego projektu do dalszych prac we właściwych komisji, tak abyśmy mogli nad nim procedować, dlatego że od momentu wpływu tego projektu do Sejmu minęło 5 dni. Natomiast dziś po prostu wiemy, że również z tej ustawy wynika, że na okres 10 lat nastąpi wzrost kosztów w agencji o 350 mln zł.

Mam nadzieję, że te wszystkie kwestie wyjaśnimy sobie w komisji i dopiero po pracach w komisji podejmiemy decyzję, jak będzie głosował klub Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Teraz w trybie zdalnym głos zabierze pan poseł Mieczysław Kasprzak, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Następnie poprosimy o zabranie głosu pana posła Rafała Bochenka. I później, także w trybie zdalnym, pan poseł Janusz Korwin-Mikke przedstawi stanowisko Koła Poselskiego Konfederacja. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt wypowiadać się w imieniu klubu Koalicja Polska w zakresie przedstawionej ustawy o Agencji Rezerw Materiałowych, zwanej rządową, w nowej wersji Agencji Rezerw Strategicznych. Zmiana nazwy i zmiana wielu zapisów w tej obowiązującej dotychczas ustawie budzi nasz wielki niepokój, dlatego że mamy jak do tej pory przykre doświadczenia z wiosny ubiegłego roku, kiedy to agencja nie mogła sobie poradzić z zakupem, a w tle były te wszystkie zdarzenia związane z zakupem maseczek czy respiratorów, i do dzisiaj z tym są problemy, z rozliczeniem tego wszystkiego. Obawiam się, że zmiana, tak szybka zmiana, bo w trybie ekspresowym, tej jakże ważnej ustawy, może mieć na celu ukrycie gdzieś tego i spowodowanie, że nikt nie będzie dochodził już tych nieprawidłowości, które miały miejsce. Ja przypominam, że zakupiono respiratory bez instrukcji, bez możliwości funkcjonowania, które gdzieś leżą. Zastanawia mnie również, po co dokonywać zmiany w tak trudnym okresie.

Myślę, że zdjęcie obowiązku i danie wielkiej swobody, bo w tej ustawie daje się dość dużą swobodę agencji, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, o przestrzeganie wszystkich zasad związanych z zakupem, jak również ze zbywaniem zgromadzonych materiałów, zawieraniem umów z podmiotami na przechowywanie tych rezerw, budzi też w nas niepokój. Do tej pory mieliśmy przykłady, że pojawiały się gdzieś w tle korupcyjne działania.

Kolejna rzecz, która pozbawia nas też w pewnym sensie kontroli, to fakt, że wiele zakupów jest objętych tajemnicą. My nie możemy w Sejmie dowiedzieć się, np. ile węgla zakupiono - to, co mój poprzednik powiedział - na zapasy Agencji Rezerw Materiałowych. Ja kilkakrotnie w Sejmie pytałem, ile tego węgla jest, po co ten węgiel kupowano, bo przecież węgla było pod dostatkiem, i do dzisiaj chyba nikt w Polsce w trybie jawnym nie może się dowiedzieć, ile tego węgla zakupiono.

Bo nie widzę tutaj żadnego sensu i żadnej potrzeby, aby pędzić i jeszcze na tym posiedzeniu, bo takie są, jak słyszę, zakusy, uchwalać tę ustawę. Z takimi zjawiskami spotykamy się na co dzień.

To nie jest tak, jak dawniej było. Doświadczenie i życie pokazało nam, że agencja musi mieć bardzo elastyczne podejście i mieć dobre rozeznanie. Swoboda z tego tytułu jest więc bardzo duża.

Dziękuję, panie marszałku, i dziękuję, Wysoka Izbo, za wysłuchanie. Dziękujemy bardzo panu posłowi. Prosimy teraz pana posła Rafała Bochenka, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Obowiązująca ustawa o rezerwach strategicznych nie zawiera dostatecznego poziomu regulacji dających możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze rezerw strategicznych wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Przykład pandemii COVID-19 i wywołanych w związku z nią niedoborów asortymentu medycznego jest jedną z przyczyn wskazujących na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych w obszarze organizacji, zadań i obowiązujących procedur tworzenia rezerw Agencji Rezerw Materiałowych oraz ich dystrybucji. Celem wprowadzonych zmian jest bardziej efektywne zabezpieczenie Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli na wypadek zagrożeń mogących wywołać zakłócenia w podaży i popycie na niektóre towary i dobra na rynku, a tym samym negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, w tym dla życia i zdrowia obywateli. Celem tej ustawy jest uproszczenie lub w niektórych sytuacjach uelastycznienie procedur, w oparciu o które działa Agencja Rezerw Materiałowych. Projektowana ustawa reguluje przede wszystkim zagadnienia z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych, a także zasady ich finansowania. Rozbudowany zostaje także zakres zadań realizowanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, która na mocy tej ustawy zmienia swoją nazwę na: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. W przedmiotowym akcie prawnym poszerzono zakres zadań, dla realizacji których tworzone są rezerwy strategiczne, poszerzono także katalog asortymentu niezbędnego do osiągania celów określonych w art. 3 przedmiotowej ustawy, co pozwoli lepiej reagować na szybko zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarczo-polityczne. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy organu nadzorującego, którym z mocy niniejszej ustawy zostaje prezes Rady Ministrów, co wydaje się uzasadnione z uwagi na to, iż to właśnie premier jest koordynatorem zarządzania kryzysowego na szczeblu centralnym, będąc jednocześnie przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. To również premier będzie organem właściwym do wydawania decyzji dotyczących udostępniania rezerw. Prezes Rady Ministrów uzyska także kompetencje kreacyjne wobec agencji, tj. powoływanie jej kierownictwa, prezesów, zastępców oraz nadawanie statutu. Ustawa w procesie planowania i programowania zasobów przewiduje uwzględnienie nowych przesłanek, takich jak ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz interesy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Szereg przepisów zawartych w projekcie umożliwia szybsze i sprawniejsze działania agencji, m.in. poprzez odformalizowanie procedur zakupowych czy zasad tworzenia rezerw lub zawierania umów związanych z przechowywaniem rezerw, jednak zawsze z zastosowaniem przejrzystych, niedyskryminacyjnych i konkurencyjnych warunków wyłaniania kontrahentów. Takie rozwiązanie będzie sprawdzać się szczególnie w sytuacjach nagłych i kryzysowych. Nową ustawową instytucją jest również możliwość utrzymywania rezerw przez agencję w formie umów o pozostawaniu w gotowości świadczenia usług. Rozbudowane możliwości likwidacji zgromadzonych rezerw Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych daje rozdział 5 przedmiotowej ustawy, wprowadzając inne formy od znanych dotychczas sprzedaży zlikwidowanych rezerw w drodze aukcji lub na giełdzie towarowej, a także np. nieodpłatne przekazanie na rzecz organizacji pozarządowych. Ustawa poszerza zadania agencji o nowe obszary, w szczególności o usługi transportowo-logistyczne, a także zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami, w których właścicielem jest agencja lub które znajdują się w jej posiadaniu, co przyczyni się do większej operacyjności i efektywności jej działań. Projekt reguluje także katalog osób objętych obowiązkami w zakresie ograniczenia prowadzenia działalności, co ma szczególne znaczenie w kontekście argumentów tutaj podnoszonych przez mojego przedmówcę, jeśli chodzi o pewien nadzór, przejrzystość i transparentność agencji. Ci pracownicy, poszerzony ich krąg w stosunku do dotychczas zakreślonego kręgu, będą zobligowani do składania okresowych oświadczeń o stanie majątkowym, co zapewni większą przejrzystość działania. Zabezpieczy to również interes Skarbu Państwa. Źródłem finansowania agencji pozostanie dotacja z budżetu państwa, a także przychody z tytułu świadczonych przez agencję usług na zasadach rynkowych. Przyjęcie przedmiotowej ustawy jest jak najbardziej zasadne, zwłaszcza w obliczu zjawisk epidemicznych, z jakimi dotychczas się mierzymy, i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Bardzo dziękuję panu posłowi.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli są różne działania rządów, to my uważamy, że rząd się niepotrzebnie wtrąca do gospodarki. Rezerwy to jest jedyna w zasadzie działalność rządu, która należy do rządu, i państwo powinno nią dysponować. Dlatego z wielką uwagą podchodzimy do tej ustawy. Nie chcemy krytykować zbyt dużo drobiazgów.

Skoro część zadań agencji przejmuje prezes Rady Ministrów, to dlaczego zwiększamy budżet agencji? Przy okazji zwracam uwagę na to, że nie mamy żadnego rządu w Polsce, tylko mamy Radę Ministrów, czyli trzecią izbę parlamentu wybieraną w wyborach pośrednich.

To jest całkowicie sprzeczne.

Dziękuję bardzo panu posłowi.

Wysoka Izbo!

Oczywiście utrzymanie tego idzie w miliardy, ale tego akurat nie neguję.

Zamiast oszczędzać i zamiast iść w stronę, o której zawsze propagandowo w kampaniach wyborczych się mówi. Oczywiście nie negujemy też tego, że będą jakieś koszty zmiany szyldu.

Troszkę szkoda.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz panią poseł Hannę Gill-Piątek, posłankę niezrzeszoną, o przedstawienie stanowiska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Najistotniejsze w tej ustawie jest to, co państwo nawyprawiali z Prawem zamówień publicznych, a właściwie z wyłączeniem spod Prawa zamówień publicznych.

Przepraszam bardzo, i dyrektywy unijne, i nasze Prawo zamówień publicznych stanowią bardzo wyraźnie, że katalog wyłączeń spod prawa zamówień publicznych musi być bardzo jasno sprecyzowany. Państwo tą ustawą naruszacie dobro publiczne właśnie w ten sposób i bardzo proszę o to, żebyście powzięli namysł, czy to rzeczywiście ma tak wyglądać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Na tym zakończyliśmy wystąpienia klubów, koła oraz pani poseł, która reprezentowała swoje stanowisko. Jeżeli nie ma więcej chętnych, to zamykam listę. Ustalam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Nie ma. W takim razie pani poseł Paulina Hennig-Kloska. Nie ma. Pan poseł Krzysztof Gadowski. Proszę bardzo. Panie Ministrze! Trzeba jasno powiedzieć, że ta ustawa to kolejne wotum nieufności wobec wicepremiera Sasina, który nadzoruje Agencję Rezerw Materiałowych i nie umie sobie dzisiaj poradzić w takiej sytuacji, a przecież mieliśmy w ostatnich czasach wiele przykładów tego, że nie daje rady. Mam do pana takie pytanie: Rządowy Program Rezerw Strategicznych jest ustalany co 5 lat.

Kolejne pytanie: Ile będzie kosztowało wejście w życie tej ustawy?

W krajach Unii Europejskiej funkcjonują podobne agencje, które zajmują się [[Dzwonek]] sprawami, które są zapisane w strategii. Chciałem się zapytać: W ilu krajach Unii Europejskiej szef rządu nadzoruje bezpośrednio podobne agencje? Proszę pana posła Dariusza Wieczorka o zadanie pytania. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oczywiście macie państwo prawo do tego, żeby tego typu zmiany wprowadzać, ale moje pytanie jest takie: Czy ta zmiana, ten projekt ustawy wprowadzany w takim tempie będzie miał swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na rok 2021?

Czy ta agencja będzie miała swoje działy, czy też wojewoda będzie odpowiadał za funkcjonowanie tych jednostek w poszczególnych województwach? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Pan poseł Tomasz Piotr Nowak. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo! W wypadku kryzysu, jak słyszymy, agencja może działać w sposób odformalizowany, z pominięciem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów zobowiązujących do stosowania przejrzystych, transparentnych, niedyskryminacyjnych i konkurencyjnych warunków wyłaniania sprzedawców. Proszę powiedzieć, kto stwierdza, że jest kryzys. W przypadku ustaw COVID-owych musimy stworzyć ustawy związane z kryzysem COVID-owym, chyba że jest stan zagrożenia, te trzy stany określone w konstytucji.

Dziękuję. Teraz prosimy panią poseł Zofię Czernow. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Proszę państwa, to jest bardzo ważny projekt ustawy i tu potrzebna jest rozwaga, trzeba przeanalizować, dlaczego agencja w tak trudnym okresie pandemii nie spełniła swoich zadań, nie spełniła swojego celu.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo!

Do tego służyła agencja. Kiedy był kupowany sprzęt, to tak jak z respiratorami: trzeba było technika z firmy, która sprzedała te respiratory, i dodatkowych części, o których nikt nie wiedział.

Mam bardzo konkretne pytanie: W jaki sposób ministerstwo, rząd tym projektem zamierza zagwarantować to, że ten sprzęt, który będzie przechowywany w dyspozycji agencji, będzie sprawny i możliwy do uruchomienia niezwłocznie? Nie tak jak teraz państwo z agencji robią, że [[Dzwonek]] trzeba technika, trzeba dodatkowej złączki, tylko w jaki sposób państwo zagwarantują to, że nie będzie konieczności czekania tydzień na uruchomienie jakiejś rezerwy?

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Mieszacie nazwami, mieszacie różnymi ustawami, ale tak naprawdę od tego mieszania nic w tych agencjach nie przybywa. Poza tym, że przybywa faktur na produkty, które albo się nie nadają do użytku, patrz: maseczki, albo ich nie ma, patrz: respiratory. Chciałbym zadać państwu konkretne pytanie: W jaki sposób procedowana przez państwa ustawa wpłynie na to, że faktycznie do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przybędą certyfikowane maseczki? Chciałbym państwa poinformować, że radomskie pogotowie otrzymało, uwaga, kilkanaście sztuk maseczek, które mają stosowne certyfikaty. A więc pytam: W jaki sposób chcecie państwo zagwarantować, że ta ustawa, w tym zmiana nazwy tej agencji, spowoduje, że popłynie strumień produktów niezbędnych do walki z koronawirusem? Bo to jest dziś najważniejsze. A w przyszłości: W jaki sposób ta ustawa ma zagwarantować, [[Dzwonek]] że będziemy gotowi na inne zagrożenia, które na nasz kraj mogą czyhać? Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Sławomir Neumann, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dwa pytania na koniec: Dlaczego tak szybko? Dlaczego procedujecie w takim terminie? Chodzi o to, że właściwie dzisiaj mamy pierwsze czytanie, jutro komisja, drugie czytanie, i chcemy tę ustawę przyjmować jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Przejęcie wszystkiego przez premiera, właściwie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w połączeniu z wyłączeniem działania ustawy o zamówieniach publicznych, każe zadać pytanie:

Jaki jest tego powód, jakie jest tego cel? Bo na pewno nie jest to jakiekolwiek rozjaśnianie sytuacji, [[Dzwonek]] jakakolwiek transparentność. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę państwa, to jest następna ustawa, której nie powinno być na tej sali teraz i w tym czasie. To jest następna ustawa, którą wrzucacie w poniedziałek, we wtorek chcecie iść z nią do komisji, w środę będzie drugie czytanie, a w czwartek albo w środę wieczorem odbędzie się głosowanie. To jest, panowie i panie, ewidentne psucie prawa. To jest, proszę państwa, psucie państwa. Tak nie wolno robić. Od tego jest Sejm, żeby ustawy tego typu były procedowane zgodnie ze wszystkimi szykanami. Od tego są komisje, które powinny - wszystkie - przyjrzeć się tej ustawie. Powinniście zdjąć tę ustawę i nie procedować nad nią w taki sposób.

Szpitala Narodowego, które pewnie wyjdą? Wydajecie pieniądze bez żadnego nadzoru i bez żadnego sensu. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Panie Marszałku! Oczywiście, każda państwowa instytucja ma prawo zmieniać swoją organizacyjną formę działania, zmieniać nazwy, ale dobrym zwyczajem jest to, żeby pozamykać sprawy, które budzą wątpliwości, a które były związane z działalnością tej instytucji. Korzystając z okazji, chciałbym zapytać i prosić o odpowiedź na piśmie na następujące pytania: Ile zostało wszczętych postępowań wobec agencji w ostatnim czasie?

Dziękuje bardzo. Proszę pana posła Marka Rutkę, Lewica, o zadanie pytania. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Procedowany projekt ustawy powstał bez konsultacji społecznych, to jednak nic nadzwyczajnego, to częsta praktyka rządu Zjednoczonej Prawicy. Projekt ustawy dotyka jednak bardzo ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa problemu, jakim jest zabezpieczenie materiałowe, i to nie tylko w przypadku pandemii, ale także w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak chociażby powodzie czy wichury. Niezaproszenie do prac nad ustawą doświadczonych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa państwa, którzy gotowi są do współpracy w wielu organizacjach pozarządowych, nie da się wytłumaczyć szybkim tempem pracy. Nie chcę jednak całkowicie krytykować przedmiotowego projektu i z uznaniem przyjmuję podporządkowanie agencji bezpośrednio premierowi. Niejako przy okazji zmianie ulegnie nazwa, z Agencji Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Mam pytanie o koszt tej operacji, wymiany szyldów w 13 regionalnych składnicach na terenie kraju, setek pieczątek, druków itd. Dziękuję bardzo. Na tym lista posłów zapisanych do zadania pytania została wyczerpana.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Postaram się odnieść do kwestii poruszonych przez państwa w trakcie zadawania pytań i poukładać je może w kilka kluczowych zagadnień. Jeżeli chodzi o samą ustawę, to chciałem podkreślić, że rząd przygotował nową ustawę, która właśnie całościowo i systemowo ma regulować kwestię funkcjonowania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Te rozwiązania bazują przede wszystkim na wnioskach, jakie rząd wyciąga z dotychczasowych doświadczeń w walce z epidemią koronawirusa. Jeżeli chodzi o procedowanie nad ustawą, oczywiście zależy nam na możliwie szybkim wejściu jej w życie, ponieważ niewykluczone, że będziemy musieli się zmierzyć z trzecią falą epidemii, a te dobre naszym zdaniem rozwiązania ułatwią walkę z epidemią. Jeżeli chodzi o przekazanie nadzoru nad agencją prezesowi Rady Ministrów, to chciałbym tutaj informacyjnie przekazać panu posłowi, że obecnie nadzór na agencją sprawuje minister właściwy do spraw energii, czyli pan minister Kurtyka. Jeżeli chodzi o samo przejście agencji pod nadzór prezesa Rady Ministrów, to wynika to z tego, że obszar ten wymaga szczególnej koordynacji. Wiąże się to choćby z tym, że w ramach agencji funkcjonują różne rezerwy, tzw. rezerwy techniczne, rezerwy medyczne czy rezerwy żywnościowe. Poza tym prezes Rady Ministrów jako konstytucyjny organ nadzoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, i to są te argumenty, które przemawiają na rzecz właśnie przekazania agencji pod nadzór szefa rządu. Wydaje się to w pełni uzasadnione. Padło pytanie o wzrost zatrudnienia w agencji. Rzeczywiście, taki wzrost jest przewidywany. On się będzie wiązał przede wszystkim z nowymi zadaniami przypisanymi agencji w zakresie logistyki i usług transportowych.

Jeżeli chodzi o kwestie przekazywania zasobów rezerwy do organizacji międzynarodowych, to tutaj chciałem wyjaśnić, jaka jest intencja. Są sytuacje, kiedy w zasobach agencji znajdują się np. sprzęty, którym kończy się resurs i których z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będziemy w stanie wykorzystać na potrzeby naszego kraju. Wtedy wydaje się w pełni uzasadnione, żeby istniała podstawa prawna do przekazania takich zasobów organizacjom międzynarodowym zapewniającym pomoc humanitarną w regionach czy w krajach dotkniętych jakimiś kataklizmami. Jeżeli chodzi o kwestie niejawności, to chciałbym nadmienić, że rzeczywiście Rządowy Program Rezerw Strategicznych ma charakter niejawny, ale takie rozwiązania funkcjonowały też do tej pory i wynikały z dotychczas obowiązujących przepisów. To się przede wszystkim wiąże z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa w kluczowych segmentach funkcjonowania państwa. Jeżeli chodzi o działania agencji, co się już nie wiąże bezpośrednio z ustawą, od wiosny, od wybuchu pandemii to oczywiście Agencja Rezerw Materiałowych zakupuje materiały na potrzeby walki z pandemią: środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące, sprzęt medyczny.

Jeżeli chodzi o kwestie instalowania sprzętu, który dostarcza agencja, to tutaj trzeba mieć na uwadze, że agencja nie dysponuje, nie mogłaby dysponować, uprawnieniami, które pozwolą modyfikować wymogi instalowania sprzętu, które narzuca ich producent. Jeżeli producent ma na względzie bezpieczeństwo działania danego sprzętu i w sposób jasny i precyzyjny określa wymogi, które muszą być spełnione przy jego instalacji, to trudno wymagać, żeby agencja mogła je modyfikować. Jeżeli chodzi o kwestie przepisów o zamówieniach publicznych, to tutaj warto zwrócić uwagę, że art. 13 projektowanej ustawy mówi o sytuacji (Dzwonek), kiedy już wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa czy obronności państwa, porządku, zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, więc nie mówimy tu o hipotetycznym zdarzeniu, tylko o zdarzeniu, które już miało miejsce. Jeżeli chodzi o to, jak to będzie stwierdzane, to prezes Rady Ministrów będzie posiadał kompetencje do wydawania decyzji o utworzeniu rezerw poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych i tam będzie wskazywane, że wystąpiło zagrożenie, o którym mowa w art. 13 projektowanej ustawy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Jeszcze pan poseł Mirosław Suchoń, który uznał, że został źle zrozumiany. Panie ministrze, powstaje pytanie, czy to pan nie zrozumiał czy państwo nic nie zrozumieli z tego kryzysu, który ma miejsce.

Już pomijam handlarza bronią, ale te respiratory, które były na stanie, dostarczyliście i one stały, bo nie było kompetencji technicznych do ich uruchomienia. A kiedy jest kryzys, to te kompetencje są niezbędne.

Bo chyba nic. Ta odpowiedź pokazuje, że państwo kompletnie nic nie zrozumieli. W jaki sposób państwo zapewnią kompetencje techniczne do uruchomienia tych urządzeń, którymi państwo dysponują? Proszę o kompetentną, konkretną odpowiedź na piśmie. Powstaje pytanie, czy ma zależeć czy dalej będziecie siedzieć na ministerialnych stołkach i udawać, że nic się nie stało. Dziękuję.

Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o rezerwach strategicznych, zawarty w druku nr 829, do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej (druki nr 801 i 819) Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, druki nr 801 i 819.

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania i po szczegółowym rozpatrzeniu projektu ustawy wnosi, aby Wysoka Izba raczyła uchwalić załączony projekt ustawy.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zapraszam pana posła Krzysztofa Lipca, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chcę przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, którego tytuł został rozszerzony po pierwszym czytaniu przeprowadzonym w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pan poseł przewodniczący komisji powiedział dokładnie, czego ta ustawa dotyczy, oraz że ważnym aspektem procesu legislacyjnego jest również fakt, że przepisy tej ustawy zostały rozszerzone i dotyczą również sytuacji Służby Więziennej, a tak naprawdę szpitali więziennych.

Poprawka przede wszystkim ma na celu uporządkowanie sformułowań zwartych w propozycji, która wyszła po pierwszym czytaniu tego projektu ustawy.

W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę poinformować Wysoką Izbę, że będziemy tę ustawę popierać wraz z poprawką, która zostanie rozpatrzona w trzecim czytaniu i po uprzednich pracach w komisji sejmowej. Bardzo dziękuję. Na ręce pana marszałka składam tę poprawkę. A stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pan poseł Michał Szczerba. Panie Ministrze!

Natomiast, Wysoka Izbo, stanowczo protestujemy wobec traktowania projektów rządowych jako miejsca wrzutek, poprawek poselskich, które wykraczają poza przedłożenie rządowe.

Panie ministrze, jak to się stało, że państwo nie przygotowaliście nowelizacji dwóch projektów, dwóch ustaw, mianowicie ustawy o chorobach zakaźnych, ustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-owi, tylko pozwoliliście na to, żeby komisja w sprawozdaniu zawarła poprawkę, która wykracza poza przedłożenie rządowe? Stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii trwa w Polsce od marca tego roku. To były kwestie, które należało w sposób systematyczny doprecyzować. Chodzi o kwestie związane z organizacją, zadaniami podmiotu leczniczego. Chodzi również o kwestię badania osadzonego przed przetransportowaniem do innej jednostki penitencjarnej. Chodzi o kwestię porad lekarskich w sposób bez kontaktu z pacjentem, o kwestię podawania leków. One nie budzą jakichś naszych bezpośrednich zastrzeżeń. Natomiast absolutnie sprzeciwiamy się tej formie procedowania, ponieważ Biuro Legislacyjne na posiedzeniu komisji stwierdziło, że tego typu wrzutka może zostać uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny, który będzie te przepisy analizował, kiedy one zostaną po prostu zaskarżone. Dlatego też opowiadamy się za tym, żeby wykreślić art. 2 i art. 3. Nie może być tak, że robimy taki śmietnik legislacyjny. Natomiast chcemy również rozmawiać o sytuacji więziennej służby zdrowia, bo to jest kwestia bardzo ważna. Państwo pamiętacie sprawę, którą analizowała Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w 2018 r. Ta kwestia dotyczyła śmierci pani Agnieszki Pysz w areszcie śledczym na warszawskim Grochowie. Później za nią przepraszał pan Patryk Jaki matkę osoby zatrzymanej, osadzonej. Mianowicie lekarze więzienni utrzymywali, że osadzona symuluje. Efektem tej symulacji była śmierć. Po prostu nie udzielono jej odpowiedniej pomocy medycznej.

Chcemy zapytać, panie ministrze, korzystając z okazji, jak wygląda przygotowanie jednostek penitencjarnych w stanie epidemii. Ilu więźniów zostało przebadanych w czasie trwającej od września, przepraszam, od marca w naszym kraju stanu epidemii? Wreszcie mam przed sobą, Wysoka Izbo, cztery wystąpienia rzecznika praw obywatelskich z ostatnich kilku miesięcy. Chciałbym, ponieważ nie na wszystkie udzielane są informacje. Co ciekawe, Wysoka Izbo, państwo również w odpowiedzi na część tych wystąpień rzecznika informujecie, że są to informacje zastrzeżone. Jaki jest powód, w przypadku którego państwo, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Służba Więzienna, używacie tej klauzuli zastrzeżenia, żeby nie udzielać konkretnych informacji? I to nie są informacje dotyczące kwestii zabezpieczenia w czasie pandemii, które mogą zostać po prostu gdzieś schowane przed organem, w szczególności organem, jakim jest rzecznik praw obywatelskich, organ konstytucyjny, który stoi na straży praw człowieka i obywatela.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Pani posłanka Anna Maria Żukowska przedstawi stanowisko klubu parlamentarnego Lewica. Wysoka Izbo! Zastanawiam się, dlaczego zawsze jest tak, że kiedy jest prosty projekt ustawy, dobry projekt ustawy, który opozycja chce poprzeć, bo są konkretne zmiany, które powinny zostać wprowadzone, to Prawo i Sprawiedliwość musi zrobić tak, żeby człowiek nie miał ochoty tego robić, bo robi to tylnymi drzwiami, przy braku przygotowania i w sposób niezgodny z regulaminem Sejmu.

Proponowane na posiedzeniu komisji poprawki, które zostały nam dostarczone jako członkom i członkiniom komisji 15 minut po rozpoczęciu komisji - nikt się do nich na początku nie chciał przyznać, nie było wiadomo, czyje to poprawki - wykraczają po prostu poza zakres przedłożenia. Tak nie powinno być. Powinno być albo zwołane posiedzenie połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia albo w ogóle tak naprawdę te poprawki nie powinny znaleźć się tutaj. Czy będzie tak, że argumentem na wszystko będzie COVID? Czy będzie tak, że do wszystkiego będziecie jako Prawo i Sprawiedliwość dopychać rozwiązania, które powinny być w normalnej ustawie, którą obywatel rozpozna po tytule i nie będzie musiał szukać regulacji w innych ustawach, na które po prostu nie przyjdzie mu do głowy nawet zerknąć? Czy będziecie zmieniać ustawę o nasiennictwie i dorzucać tam rzeczy związane ze służbą zdrowia? Niestety nadal się do tego nie przyzwyczaiłam, Lewica się do tego nie przyzwyczai i będziemy to kontestowali.

To są nasze uwagi. Co do meritum, to popieramy zarówno podwyższenie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na ryczałt na dojazdy dla funkcjonariuszy, którzy dojeżdżają do swojego miejsca pracy spoza miejsca zamieszkania. To jest rozwiązanie, które musimy po prostu przyjąć. Natomiast wszystkie inne rozwiązania po prostu powinny się znaleźć w ustawie COVID-owej, a nie w ustawie zmieniającej ustawę o Służbie Więziennej, i nie powinny być ze sobą łączone. Powinniście to państwo jako Prawo i Sprawiedliwość przewidzieć wcześniej i nowelizację ustawy COVID-owej przeprowadzać na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Dziękuję pani posłance. Teraz stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawi pan poseł Krzysztof Paszyk. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Koalicja Polska również jest za tym, aby znowelizować ustawę o więziennictwie w tym zakresie, w którym jest to niezbędne, i w tym zakresie, o którym mówi projekt rządowy.

Chciałbym dowiedzieć się przy okazji, panie ministrze, czy te poprawki zarówno na posiedzeniu komisji, jak i dzisiaj, zostały złożone w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy to jest jakaś kolejna odsłona wojenki, która się rozgrywa między tą większością Prawa i Sprawiedliwości a środowiskiem, które pan reprezentuje. Bo trochę to dziwnie wygląda, a myślę, że warto by to było wyjaśnić.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze dwóch panów posłów. W pierwszej kolejności pan poseł Krzysztof Tuduj, następnie pan poseł Dobromir Sośnierz. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początek i na zachętę kilka pochwał. Dobrze, że ustawodawca dba o funkcjonariuszy Służby Więziennej dojeżdżających do miejsca pracy. O wszystkich funkcjonariuszy trzeba dbać, aby rósł etos służby dla niepodległej Rzeczypospolitej.

To daje poczucie, że ktoś coś planuje, tak że to są jakieś plusy. Oczywiście trudno przewidzieć wartość tych pieniędzy za parę lat przy obecnych nieustannych podwyżkach podatków, dodrukowywaniu pieniędzy. To jest taka pułapka jak PiS-owski sztandarowy projekt 500+, którym udało się przekonać wyborców, że państwo stało się przyjazne, a jednocześnie wzrost danin publicznych, podatków powoduje, że te pieniądze realnie straciły swoją wartość, pewnie już są warte połowę tego, co były warte, jak je wprowadzano. Tak że dalej rozwijacie ten zagmatwany system, tak zagmatwany, że nawet wykładowcy uniwersyteccy nie chcą używać frazy „system podatkowy”, bo to, co ma miejsce w Polsce, to już nie jest system, bo system to jest coś kompletnego.

Pilnujcie tylko, żeby nie była to okazja do ucieczki więźniów i, co było wytykane, do przekrętów finansowych urzędników, którzy źle pojęli zachętę do przedsiębiorczości. Ale jeśli już zaglądamy do więzienia przez dziurkę od klucza, to możemy zobaczyć coś ważnego. Więzienia przypominają nam o sprawiedliwości, przypominają o tym, kto tam powinien siedzieć, a nie siedzi, i kto nie powinien siedzieć, a siedzi. Kto nie powinien siedzieć? Nie powinna siedzieć sprawiedliwość, a siedzi tam i cichym głosem pyta: Dlaczego nie siedzą ci, co powinni? Nie ma w więzieniach zdrajców Polski z ostatnich dekad. Zdrada stanu w Polsce praktycznie jest niekarana, co woła o pomstę do nieba. Nierozliczona prywatyzacja z lat 90., wszystkie kanty okrągłego stołu trwające do dziś, ale też 8 lat rządów PO-PSL, ogromna liczba afer. Przecież na tym wygraliście wybory, szanowni państwo. I chciałbym przypomnieć, że był taki minister skarbu PiS Dawid Jackiewicz, który nawet to wyliczył, prezentując z mównicy sejmowej rok po objęciu rządów przez PiS „Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL” Cytat z ministra Jackiewicza: Jest to dokument cząstkowy, fragmentaryczny, ponieważ nasze badania i analizy wciąż trwają i przychodzą nowe informacje. Z takimi właśnie działaniami mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat, jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym, który nie należy przecież do polityków, nie należy do urzędników, należy do nas, do wszystkich Polaków. Te słowa to pazerność, niegospodarność, rozrzutność, łamanie procedur, wykorzystywanie spółek do celów politycznych oraz działania na szkodę interesu państwa - koniec cytatu. Aferzyści nierozliczeni, ministra nie ma w rządzie ani w polityce. Naruszył układ i się od niego odbił. Ręka rękę myje. My waszych nie ruszamy, wy naszych nie ruszacie. Okrągły stół trzyma się mocno, ale tak nie będzie w Polsce w nieskończoność. Czekamy, czekamy i zrobimy go za was, bo wy nie chcecie, nie potraficie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Dobromir Sośnierz jest obecny na sali lub w trybie zdalnym? Przystępujemy do zadawania pytań, do których zgłosiło się siedmioro państwa posłów. Jeżeli nie ma więcej osób chętnych, zamykam listę. Ustalam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Pierwszy pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.

Rok temu NIK skierowała do prokuratury aż 16 zawiadomień dotyczących nieprawidłowości w programie „Praca dla więźniów” Najwyższa Izba Kontroli opublikowała teraz wyniki szczegółowej kontroli, w której skupiła się na omijaniu przetargów przez jednostki podległe ministerstwu. NIK zarzuca Służbie Więziennej nierzetelny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi podległymi i nadzorowanymi przez ministra, który sprzyjał powstawaniu mechanizmu wehikułu inwestycyjnego polegającego na dopuszczeniu możliwości zlecania przez zakłady podmiotom zewnętrznym podwykonawstwa w dowolnym zakresie. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że od stycznia 2017 r. do połowy 2019 r. do prywatnych przedsiębiorców trafiło w ten sposób ponad 560 mln zł. Jak się resort sprawiedliwości odnosi do wyników ustaleń niezależnych kontrolerów NIK? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania panią poseł Katarzynę Kretkowską, Lewica.

Czy mógłby pan powiedzieć, ilu tych funkcjonariuszy mamy w tej chwili, tj. na koniec listopada br. Ile mamy wolnych wakatów? Ilu z nich korzysta? Panie pośle, jest pan wieloletnim posłem, prawnikiem. Czy to jest niezgodne z konstytucją? Dlaczego państwo nie zaproponowaliście tej poprawki do ustawy COVID-owej, która jest w tej chwili w Sejmie?

Dziękuję bardzo. Proszę pana posła Aleksandra Miszalskiego, Koalicja Obywatelska, o zadanie pytania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Generalnie ustawa o ustanowieniu tych nowych limitów wydatków na ryczałty ma sens. Po pierwsze, wskazujecie, że dotyczy to ponad 26 tys. osób. To jest jednak liczba wszystkich funkcjonariuszy. Pytanie, ilu z nich faktycznie będzie przysługiwał ten ryczałt. Pewnie wielu, skoro przenosicie ich na drugi koniec Polski, np. za to, że ujawnili nadużycia w Służbie Więziennej.

Czy dlatego właśnie zwiększacie te wydatki na te ryczałty, że tak dużo funkcjonariuszy przenosicie za karę w inne miejsca Polski i będziecie je musieli podnieść? Proszę o informację na piśmie, ilu funkcjonariuszy otrzymywało ten ryczałt w ostatnich latach, jak te liczby się zmieniają. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Trudno nie mieć takiego wrażenia, że w tej ustawie - pomimo tego, że dotyczy tylko kwestii finansowych - widzimy jak w pigułce, jak niszczycielskie dla państwa, dla jego służb są rządy Zjednoczonej Prawicy. Panie Ministrze! Wszyscy słyszeliśmy o tych absolutnie niedopuszczalnych przypadkach, w których de facto państwa rząd przykłada ręce do ukarania funkcjonariuszy działających dla służby, dla poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, karząc ich za to, że próbują ze swojego środowiska, ze Służby Więziennej eliminować patologie, które wy umacniacie. Umacniacie patologie w tej służbie. Mam więc pytanie: Kiedy rzeczywiście przeprowadzą państwo obiektywną, racjonalną, pożądaną reformę i zmianę warunków pełnienia służby w taki sposób, żeby warunki tej służby odpowiadały odpowiedzialności, którą ponoszą codziennie funkcjonariusze? Kiedy ze środowiska zaczniecie eliminować te patologie, które wam dzisiaj służą? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę pana posła Konrada Frysztaka, zatem uznaję, że lista posłów zapisanych do zadania pytania została wyczerpana. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy. Dziękuję za te głosy na temat pierwszej części przedłożonej przez rząd, a mianowicie na temat limitów finansowych na ryczałt za dojazdy, za delegowanie. W tym zakresie jest ogólne poparcie, tak że za to dziękuję. Natomiast dziękuję także Klubowi Parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwość za zgłoszenie poprawek, bardzo sensownych poprawek, usprawniających funkcjonowanie Służby Więziennej w dobie pandemii. Te poprawki rząd popiera i zmierzają one w kierunku dalszej, skutecznej walki z szerzącą się epidemią, także za kratami. Chociaż trzeba powiedzieć, że do cel koronawirus nie zagląda. Za chwilę o tych szczegółowych danych będę mówił. Poprawki wprowadzają możliwość delegowania funkcjonariuszy Służby Więziennej do wsparcia także cywilnej służby zdrowia czy wolnościowej służby zdrowia, gdyby była taka potrzeba.

Szanowni państwo, dzisiaj z mównicy sejmowej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z dumą mogę podziękować tysiącom funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy bardzo dobrze radzą sobie z pandemią koronawirusa. Drodzy państwo, niech o tym świadczą dane, konkretne dane.

Czyli we wszystkich tych krajach niestety radzą sobie gorzej niż u nas. Dzisiaj wypada podziękować Służbie Więziennej za tę ciężką, codzienną, profesjonalną pracę, która spowodowała, że rzeczywiście z koronawirusem Służba Więzienna radzi sobie bardzo dobrze.

Co do pytań i odpowiedzi w ramach klauzuli zastrzeżonej, to pan poseł doskonale zdaje sobie sprawę, że część spraw jest na tyle wrażliwych, związanych z bezpieczeństwem państwa, że wymagają nadania takiej klauzuli i także co do tego trybu nie miał dotychczas zastrzeżeń i nie zgłaszał ich rzecznik praw obywatelskich, na którego pan poseł się powołał w tym zakresie. Co do pytań o raport Najwyższej Izby Kontroli.

Zostały one uznane przez te instytucje za właśnie absurdalne. Przecież to jest coś normalnego, że są preferencje w ramach przetargów dla tych, którzy zatrudniają skazanych, po to, żeby ich resocjalizować. Takie preferencje są nie tylko w Polsce, ale są także na całym świecie, bo przecież system penitencjarny nie służy tylko wymierzeniu kary - to jest oczywiście pierwsza, podstawowa jego powinność - ale także resocjalizacji skazanych, readaptacji społecznej. To jest wykonywane.

Pan marszałek wybaczy, ale jeśli chodzi o pozostałe pytania o rzekome przenoszenia karne - zupełnie absurdalne pytania - czy o umacnianie patologii - znowu lanie słów bez konkretów - nie za bardzo jest na co odpowiadać, bo Służba Więzienna jest bardzo dobrą formacją, sprawną formacją, trzecią pod względem wielkości uzbrojoną formacją w Polsce, która doskonale radzi sobie nie tylko z pandemią, ale też chroni polskie bezpieczeństwo, i która w ostatnich latach, w ostatnich 5 latach została doinwestowana na taką skalę (Dzwonek), o jakiej w czasie poprzednich rządów mogli tylko pomarzyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Jeszcze w tej kwestii w trybie, powiedzmy, sprostowania głos zabierze pan poseł Michał Szczerba. Jakby ewentualnie pan minister później uznał, że chce odpowiedzieć, to też proszę bardzo. My oczywiście nie mamy żadnych wątpliwości, że praca dla więźniów powinna służyć więźniom. Problem jest taki, że Najwyższa Izba Kontroli w swoich wnioskach pokontrolnych przedstawia tę informację całkiem inaczej.

Komercyjnych podwykonawców, którzy, panie ministrze, nie mieli nałożonego obowiązku zatrudniania więźniów.

Proszę do tej sprawy albo się odnieść, albo przedstawić na piśmie konkretne wyjaśnienia, ponieważ raport NIK-u w tej sprawie jest jednoznaczny i nasze stanowisko jest takie, że powinniśmy po prostu przyjąć te wyjaśnienia. A jeżeli pan twierdzi, że jakieś organy się tą sprawą zajmowały - tak, zajmowały się organy śledcze, takie jak chociażby prokuratura. Prokuratura, która jest podporządkowana temu samemu ministrowi, który sprawuje nadzór nad Służbą Więzienną. Pan minister udzieli odpowiedzi, panie pośle. Nie wiem, czy w trybie sprostowania, ale jeszcze raz.

Po to są wprowadzone preferencje ustawowe, żeby więźniowie pracowali przy takich pracach, do których się nadają, gdzie mogą dobrze, sprawnie wykonać swoją pracę, bo przez pracę się resocjalizują. I jest oczywiste dla każdego, że jeżeli budujemy halę produkcyjną, jakieś inne wysokotechnologiczne, skomplikowane miejsce, to przy takim zatrudnieniu w sposób oczywisty są podwykonawcy. Ale też jest oczywiste, że w tych umowach zastrzega się także - w większości przypadków - to, że to więźniowie przy tym pracują, panie pośle, i serdecznie polecam szczegółowo doczytać, przyjrzeć się tej sprawie, żeby popierać dobre programy, które służą readaptacji społecznej tych, którzy są wykluczeni. Jako ostatni głos zabierze pan poseł Marek Ast, który jest sprawozdawcą komisji. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim członkom komisji za uwagi zgłoszone w trakcie pierwszego czytania projektu i procedowania nad nim w komisji, za poparcie tego podstawowego projektu, ale również za uwagi zgłoszone do poprawek. Pan poseł Wiesław Szczepański pyta o zgodność z konstytucją takiego procedowania.

Działamy w nadzwyczajnej sytuacji, a te poprawki zmierzają wprost do ochrony zdrowia i życia osadzonych i funkcjonariuszy, więc też z tego względu. Tym bardziej że co do merytorycznej zawartości tych poprawek właściwie żaden z klubów nie zgłosił zastrzeżeń. Zwracam się też i w imieniu komisji o poparcie tych poprawek i całego projektu. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druki nr 766 i 812) Proszę pana posła Mariusza Trepkę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. To jest druk nr 766. Marszałek Sejmu, zgodnie z regulaminem, skierowała w dniu 20 listopada 2020 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania. Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2020 r. wnoszą: Wysoki Sejm przyjąć raczy załączony projekt ustawy. Panie Marszałku! Procedowana ustawa podczas wspólnych posiedzeń Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury była, powiedziałbym, przyjęta bardzo zgodnie przez wszystkich parlamentarzystów uczestniczących w pracach tych komisji. Za tym projektem ustawy głosowało 51 posłów, nikt nie był przeciw, 3 się wstrzymało. Projekt ustawy będzie stanowił podstawę prawną realizacji programu: lokal za grunt, pierwszego z instrumentów tzw. części rynkowej pakietu mieszkaniowego. Program ten jest jednym z narzędzi mających niwelować negatywne skutki pandemii COVID-19 w sferze budownictwa. Ma na celu szersze wykorzystanie nieruchomości publicznych pod zabudowę, w tym zabudowę mieszkaniową. Program: lokal za grunt opiera się na formule częściowego rozliczenia ceny nabywanej przez inwestora nieruchomości publicznej, tj. z gminnego zasobu nieruchomości lub pochodzącego z Krajowego Zasobu Nieruchomości, lokalami mieszkalnymi lub użytkownymi, które inwestor przekaże gminie. Podstawowy model zakłada wykorzystanie nabytej nieruchomości na cele mieszkaniowe. W tym modelu gmina w przetargu nieograniczonym dokona sprzedaży inwestorowi nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. Część rozliczenia ceny nieruchomości zostanie dokonana w postaci pieniężnej, natomiast reszta będzie podlegała uiszczeniu w terminie późniejszym, po wybudowaniu mieszkań. Następnie inwestor wybuduje budynek mieszkalny i przekaże część mieszkań gminie. Gmina będzie mogła te mieszkania wykorzystać jako mieszkania komunalne albo wnieść je przykładowo do spółki gminnej. Wniesione do spółki gminnej mieszkania będą mogły być przeznaczone do wynajmu, np. z dojściem do własności. Najemcy tych mieszkań będą mogli dodatkowo ubiegać się o dopłaty z czynszu w ramach programu „Mieszkanie na start”

Dodatkowe zachęty dla gmin do angażowania się w działania służące realizacji polityki mieszkaniowej państwa przewidują preferencje przy łączeniu działalności promieszkaniowej z innymi formami działania gmin na rzecz lokalnej wspólnoty prowadzonymi z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych lub Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo panu posłowi.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poprawa dostępności mieszkań przez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych jest jednym z priorytetów polityki mieszkaniowej państwa określonej w „Narodowym programie mieszkaniowym” przyjętym w 2016 r.

Nowy model inwestycyjny zainicjowany w roku 2016 to budownictwo na wynajem z opcją stopniowego dojścia do własności realizowany przez PFR Nieruchomości SA, który powinien uzupełnić budownictwo komunalne i budownictwo społeczne. Ogromnie istotną rolę mają inwestycje zwiększające zasoby mieszkań o stosunkowo niskich czynszach prowadzone z zaangażowaniem gmin. Tu czynnikiem stymulującym powinien być rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa zasilony kwotą 1,5 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz bardzo wysokie wsparcie finansowe dla gmin, które aktywnie angażują się w inwestycje mieszkaniowe.

Wysoka Izbo! Wobec negatywnych skutków dla gospodarki pandemii COVID-19 konieczne jest wprowadzanie działań stymulujących budownictwo mieszkaniowe i likwidujących bariery w jego rozwoju. Jedną z takich barier ograniczających rozwój budownictwa, zwłaszcza rynkowego, jest dostępność gruntów pod zabudowę. Problemem jest także brak uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną i niski dostęp do infrastruktury społecznej. Rozwiązania przewidziane w omawianym projekcie ustawy z druku nr 766 określają - w art. 1 - zasady zbywania nieruchomości przez gminy z rozliczeniem w cenie nieruchomości z gminnego zasobu ceny lokali lub budynków przekazywanych w zamian za grunt przez inwestora, czyli nabywcę nieruchomości, czyli tzw. rozliczenie „lokal za grunt”, a także zasady kwalifikowania, zbywania i rozliczania. Dodajmy, że status tej działki musi być ustalony - albo musi być zapis planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzja o warunkach zabudowy, a nie kot w worku dla kontrahenta, jeśli chodzi o ten teren. Warto zauważyć, że cena gruntu to jest między 5% a 20% wartości zabudowanej nieruchomości, zatem taka może być skala pozyskiwanych przez gminy mieszkań do zasobu komunalnego. W projekcie ustawy określa się również sposób postępowania z tak pozyskanymi lokalami w razie podjęcia decyzji o wniesieniu ich do spółki - spółki gminnej albo spółki Skarbu Państwa. Projekt po jego uchwaleniu umożliwi gminom uzyskanie wsparcia na budowę infrastruktury technicznej bądź też infrastruktury społecznej dla przedsięwzięć z zakresu mieszkalnictwa. Stanowi o tym chociażby art. 15, który zawiera zmiany do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych itd. Projekt pozwoli także na udzielenie preferencji gminom w dostępie do środków z Funduszu Dróg Samorządowych, o czym mówi art. 18, który zawiera zmiany do ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, a także ułatwi dostęp do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - mówimy o art. 19. Wszystko to dla lepszego skomunikowania i obsługi powstającego zasobu mieszkaniowego. Najemcy tak pozyskanych mieszkań będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu z programu „Mieszkanie na start” Tu z kolei są zmiany zawarte w art. 17, zmiany do ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Żeby polskie rodziny mogły normalnie żyć, wychowywać nowe pokolenia Polaków, potrzebują nie tylko pracy, stabilnego zatrudnienia za godziwą zapłatę czy wsparcia w wychowaniu dzieci, lecz także własnego lub wynajętego na możliwych do udźwignięcia warunkach mieszkania. Poprawa dostępności mieszkań to najważniejszy problem do rozwiązania.

Oba te projekty ustanawiają nowe instrumenty realizacji programu mieszkaniowego rządu Zjednoczonej Prawicy. Dotrzymujemy słowa. Wiarygodność i realizacja publicznie składanych obietnic to wyróżnik odpowiedzialnej i rzetelnie prowadzonej polityki. Dlatego mój klub Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za projektem ustawy z druku nr 766. Panie Marszałku! Pozwolę sobie w imieniu mojego klubu złożyć trzy poprawki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł, za przedstawienie stanowiska klubu parlamentarnego i złożenie poprawek. Teraz pan poseł Michał Krawczyk przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Czytając uzasadnienie do przedmiotowego projektu ustawy, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ten projekt ustawy, o którym dziś rozmawiamy, zwany potocznie lokal za grunt, został stworzony po to, aby dzięki samorządom rząd Prawa i Sprawiedliwości uratował „Narodowy program mieszkaniowy”, tak hucznie zapowiadany wraz ze sztandarowym programem „Mieszkanie+”, podczas inauguracji którego ówczesna premier Beata Szydło, dokładnie 4 lata temu, bo 12 października 2016 r., mówiła: „Mieszkanie+” staje się faktem. Rozpoczynamy wielki program mieszkaniowy dla polskich rodzin i Polaków, dla tych wszystkich, którzy marzą o własnych mieszkaniach. Zostawiliście państwo polskie rodziny z tymi marzeniami, no bo na pewno nie z nowymi mieszkaniami. Przez 4 lata funkcjonowania programu „Mieszkanie+” w ramach jego części rynkowej powstało 1017 mieszkań - 250 mieszkań rocznie. W „Narodowym programie mieszkaniowym”, na który powołujecie się państwo w uzasadnieniu projektu ustawy, założyliście, że do 2030 r. w Polsce liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców będzie zrównana średnio ze średnią unijną. W Polsce wynosi ona obecnie 380, w Unii Europejskiej - 435.

W ciągu państwa kilkuletnich rządów średnia liczba wybudowanych mieszkań.

Choć sam pomysł i zamiar rozliczania ceny wybudowanego lokalu czy budynku w cenie nabywanego gruntu nie jest zły, to musicie sobie państwo zdać sprawę z tego, że tylko takim pomysłem i tylko przerzucaniem odpowiedzialności na samorządy nie uratujecie państwo „Narodowego programu mieszkaniowego” i „Mieszkania+”

Z punktu widzenia ładu przestrzennego zdecydowanie lepiej jest, jeśli inwestycja lokalizowana jest - i mówię to także jako były samorządowiec - na gruntach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Natomiast projekt ustawy niewątpliwie jest krokiem w dobrym kierunku, choć, tak jak powiedziałem, dopiero po pewnym czasie okaże się, czy te wątpliwości, które ja tu dzisiaj zgłaszam, uniemożliwią jej funkcjonowanie w praktyce, a jest takie bardzo poważne zagrożenie. Stanowisko klubu Lewica przedstawi Wysokiej Izbie pani poseł Monika Falej. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z problemem niedoboru mieszkań i wysokimi cenami już istniejących mamy problem od wielu lat. Nie wspomnę już o tym, co jest tego pochodną - wiele Polek i wielu Polaków nie stać na wynajem mieszkania. Zatem cieszy każda próba regulacji na rynku mieszkaniowym. Każda, która jest na plus, każda, która nie jest iluzoryczna, bo jak wiemy, wielki projekt „Mieszkanie+” okazał się wielką klapą. O zaletach przedstawionego projektu, rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, nie będę mówiła, bo wielokrotnie takie słowa padały z ust ustawodawców i partii rządzącej.

Wskażę jednak na kilka mankamentów budzących wątpliwości związane z tym projektem.

Ustawa nie precyzuje, jaki procent powierzchni mieszkaniowej powinien być zagwarantowany gminom. Możliwa jest sytuacja, że gmina na inwestycje 500 mieszkań otrzyma tylko jedno. Od razu nasuwają się wątpliwości, czy to nie będzie prowadzić do nadużyć. I kolejna rzecz, która nie została doprecyzowana, to kwestia, czy mieszkania pozyskane w ten sposób pozostaną w zasobie stałym gmin. Wiemy również, że wybudowanie przez gminę mieszkań może być tańsze. Nie ma więc idealnej sytuacji. Ustawa też przychodzi za późno w sytuacjach tych gmin, które mają braki w gruntach, a były zmuszone je wyprzedać wcześniej. Dopracować należy m.in. zapisy o dofinansowaniu przez gminę czynszów w lokalach przekazywanych przez inwestorów, a zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. To wspólnoty będą ustalały wysokość czynszu, a nie gminy. Koszt utrzymania takiego mieszkania może przekroczyć możliwości gminy, a nie jest to do uregulowania na etapie ustaleń z inwestorem. Ustawa daje możliwości, z ograniczeniami, bez gwarancji sukcesu, jednak Lewica popiera każde rozwiązanie, które może przynieść pozytywne efekty, jednak w przypadku doprecyzowania wyżej wymienionych wątpliwości. Składam poprawki w imieniu klubu Lewicy. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska pan poseł Jacek Tomczak. Bardzo proszę, panie pośle.

Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska w sprawie sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Projekt ustawy wprowadza możliwość nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości, w cenie lokali lub budynków mieszkalnych lub użytkowych przekazanych gminie przez nabywcę nieruchomości. Lokale lub budynki, których cena będzie zaliczana na poczet części cen nieruchomości, będą mogły być wykorzystywane przez gminę do realizacji jej zadań. Możliwe będzie również pozyskiwanie przez gminę w tym trybie powierzchni pod obiekty kulturalne, edukacyjne czy opieki zdrowotnej.

Celem projektu jest ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnych, wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań. Drugim istotnym celem rozwiązania zawartego w projekcie ustawy jest umożliwienie samorządom ubiegania się o grant na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu.

Pamiętajmy, że uwarunkowanie każdej inwestycji jest kompletnie inne, więc regulowanie tych cen nieruchomości i parametrów, w oparciu o jakie będą dokonywane te transakcje przez rady gminy, może być rzeczą, która po prostu zablokuje te procesy. Natomiast warto pamiętać, że dzisiaj w polityce mieszkaniowej, którą chcielibyśmy rozwijać, jednym z głównych problemów jest przede wszystkim dostęp do kredytu.

Jeżeli nie zmienimy akurat tego aspektu i nie będzie sensownego programu wsparcia dla Polaków w uzyskaniu kredytów właśnie na pozyskanie mieszkania, to wówczas nie będzie szansy na to, ażeby ta polityka mieszkaniowa ruszyła, i żaden z projektów tak naprawdę tego nie zmieni. A więc warto spojrzeć na efekty programu MdM, „Mieszkanie dla młodych” Ze wszystkich wskaźników, jakie możemy analizować z perspektywy lat, porównując go do „Mieszkania+” i innych programów mieszkaniowych, wynika, że był to najskuteczniejszy program, który wsparł najwięcej polskich rodzin w uzyskaniu dostępu do mieszkania. Warto nad tym się pochylić i pomyśleć o innych, nowych instrumentach, które mogłyby wspierać polskie mieszkalnictwo i umożliwić polskim rodzinom dostęp do mieszkań. Pewnie praktyka spowoduje, że będziemy ją nowelizować, natomiast niewątpliwie jest to krok w dobrą stronę. Klub Parlamentarny Koalicja Polska będzie wspierał przedłożony projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Stanowisko koła Konfederacja przedstawi pan poseł Krystian Kamiński.

Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości dotyczy określenia zasad zbywania w przetargach nieograniczonych nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości z możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań. Czyli chodzi o to, że rząd chce zwiększyć dostępność gruntów pod inwestycje mieszkaniowe poprzez ograniczenie jednej z podstawowych barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w Polsce, jaką jest zbyt mała oferta rynkowa nieruchomości odpowiednich pod zabudowę. Samorządy gminne mają otrzymać dodatkowe wsparcie w realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej, mogą liczyć m.in. na zwiększenie liczby lokali na swoim terenie oraz finansową pomoc państwa w realizacji infrastruktury technicznej i społecznej. Jak to ma wyglądać w praktyce? W podstawowym modelu inwestor, czyli nabywca nieruchomości od gminy, budowałby budynek, ewentualnie remontował, przebudowywał i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować w swoim zasobie lub wnieść je do spółek gminnych, TBS-ów. Dlaczego to jest dobry program? Dlatego że pierwszy raz - pierwszy raz, w przypisie, to zawsze jest coś nowego - nie wszystko państwo ma robić czy nie wszystko gmina ma robić, tylko pozwalamy prywatnym inwestorom współpracować. Pozwalamy na to, żeby prywatny inwestor mógł współpracować z kimś, mógł razem z gminą coś stworzyć.

To zwykle gminy mają problem z budowaniem mieszkań komunalnych, ponieważ z jednej strony brakuje funduszy, a jak już są te fundusze, to potem trzeba je jakoś rozliczyć, potem ewentualnie jest przekazywanie tych mieszkań, sprzedaż, zgoda rady miasta na sprzedaż mieszkań, bonifikaty itd. To są zawsze utrudnienia. W związku z tym jest to krok w dobrym kierunku. Uważam, że im więcej prywatnych pieniędzy, im więcej prywatnych inwestorów, im mniej gminy, im mniej państwa przy budowie mieszkań - tym lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Przed chwileczką go gdzieś widziałam, ale dobrze. Bardzo proszę, pani poseł.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Kiedy czytamy uzasadnienie tego projektu ustawy, to zastanawiamy się, dlaczego to uzasadnienie nie jest oparte o fakty. Projektodawcy piszą, że zapaść czy może nie zapaść, ale trudna sytuacja w gospodarce mieszkaniowej wynika z zaniedbań procesów inwestycyjnych w poprzednich latach, dopiero ostatnio jest poprawa. Kolejna sprawa - niska skłonność gmin do angażowania się w bezpośrednie procesy inwestycyjne. A kto do tego doprowadził? Dlaczego samorządom zabiera się pieniądze, a w okresie pandemii w ogóle się je pozbawia jakichkolwiek środków, żeby mogły inwestować?

To jaki to jest projekt ustawy, kiedy sami podkopujemy swoje możliwości realizacji? Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, klub Lewica, zdalnie. Czy mamy połączenie? W takim razie może pani poseł Magdalena Biejat, klub Lewica. A na połączenie poczekamy. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To, w jakiej sytuacji jest obecnie rynek mieszkaniowy w Polsce, stanowi źródło wielu problemów, zwłaszcza dla młodych ludzi. Od dawna rozmawiamy o tym, że brakuje tanich mieszkań na wynajem, brakuje mieszkań, które można będzie wynająć w ramach organizowanych w jakiś sposób przez instytucje publiczne, po to żeby były wyjęte spod tej zupełnie bezlitosnej logiki wolnego rynku, która każe obecnie zadłużać się na całe życie, żeby móc mieć swój dach nad głową. W tej sytuacji tworzenie wszelkich narzędzi służących do tego, żeby zwiększyć zasób komunalny, zwiększyć zasób lokalowy w zasobie gminnym, jest słusznym kierunkiem. Pytanie tylko brzmi, dlaczego państwo w żaden sposób nie zabezpieczacie możliwości zachowania tych lokali w zasobie gminnym, ponieważ nic w obecnie procedowanej ustawie nie stoi na przeszkodzie, żeby następnie gminy mogły te lokale wyprzedawać.

Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Doceniam bardzo tę troskę o gminne zasoby mieszkaniowe. Doceniam tym bardziej, że od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia z zapaścią budownictwa komunalnego. Poprzednie rządy zrzuciły problemy mieszkaniowe milionów Polek i Polaków na deweloperów. Kolejki oczekujących na mieszkanie rosną. A co robią młodzi ludzie?

Nie może być tak - a wy na to pozwalacie - by deweloper, korzystając z waszej ustawy, mógł na preferencyjnych warunkach wybudować 1000 mieszkań, a jedną kawalerkę oddać do gminnego zasobu mieszkaniowego. Dlatego zgłosimy poprawkę, która to ureguluje. Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Składową częścią „Narodowego programu mieszkaniowego” jest program „Mieszkanie+”, który funkcjonuje od 2016 r. Jest to rządowy program Prawa i Sprawiedliwości. Jest kompletnie niewydolny i nie spełnia swojego zadania, ponieważ został źle skonstruowany. Do błędnych rozwiązań legislacyjnych programu „Mieszkanie+” dochodzi jeszcze koniunktura gospodarcza.

Zapraszam, pani poseł. Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W Polsce wciąż zmagamy się z deficytem mieszkaniowym, mimo iż rok 2019, jeżeli chodzi o liczbę oddanych mieszkań, był najlepszy po 1989 r. Przyjęty do realizacji „Narodowy program mieszkaniowy” określa główne cele i środki realizacji polityki mieszkaniowej państwa w perspektywie do roku 2030.

Szansą zwiększającą dostęp do nieruchomości jest wykorzystanie możliwości inwestycyjnych tworzonych przez zasoby nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. Moje pytanie brzmi: Czy proponowana ustawa zwiększy udział samorządów i firm deweloperskich w budowaniu takich mieszkań? Kolejne pytanie zada pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Pani poseł Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska. Nie ma. Ale, szanowni państwo, to po co się zgłaszać do pytań? Bardzo proszę, panie pośle.

Wysoka Izbo!

Po drugie, w gminach wielkomiejskich takich jak na przykład Kraków - skąd jestem - duża część mieszkańców sprzeciwia się w ogóle przekazywaniu kolejnych terenów deweloperom pod budowę nowych mieszkań i woli je zagospodarowywać na tereny zielone. To też może być proces, który uniemożliwi tego typu działanie w dużych miastach. Obawiam się osobiście, że państwo po prostu robicie tę ustawę w celach propagandowych, po to żeby, po pierwsze, nie musieć tłumaczyć się z tego, dlaczego „Mieszkanie+” jest jedną wielką klapą i fiaskiem, po drugie, zrzucić odpowiedzialność na samorządy i później mówić, że to samorządy sobie nie poradziły i mimo dobrej ustawy tego nie zrobiły. Dziękuję bardzo. Pan poseł Cezary Grabarczyk. Nie ma. Pan poseł Marek Rząsa, Koalicja Obywatelska. Nie ma.

Nie zadaje pan pytania? Pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska.

Zaraz będziemy to wyjaśniać. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście wszyscy wiemy, że program mieszkaniowy rządu to jest klapa, absolutna klapa i kompromitująca klapa.

Te przepisy tworzą wyłam w decyzjach gmin, w zasadzie bez możliwości konsultacji czy w ogóle bez konsultacji z mieszkańcami. To ma oczywiście taki skutek, że zabudowa rozlewa się na tereny, które do tej pory nie były w jakiś sposób uzbrojone. To powoduje, że rosną koszty związane z dostosowaniem nowych terenów do budownictwa, a co za tym idzie, cała polityka mieszkaniowa jest po prostu nieekonomiczna. W związku z tym mam jedno pytanie: Czy rząd w ogóle rozważa w trakcie prac nad projektami ustaw kwestie kosztów infrastruktury, kosztów dostosowania nowych terenów i tego, jakie one będą w przyszłości, w jaki sposób będą obciążały budżety gmin i budżet państwa? Dziękuję bardzo. Tak, akurat pan poseł tak, ale lista osób została zgłoszona do pkt 5, tak że właściwie zostało tu przekazane, błąd był gdzieś u państwa w klubie. Pani poseł Karolina Pawliczak, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związku z regulacjami zawartymi w niniejszej ustawie, wprowadzającymi możliwość nabywania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na szeroko rozumiane cele inwestycyjne z rozliczeniem w cenie tych nieruchomości właśnie o tę cenę chciałam zapytać.

Bardzo proszę o informację. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Chciałbym zapytać.

I kwartał 2017 r. Str. 75: Pakiet Mieszkanie+: Wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe, indywidualne konto mieszkaniowe - projekt ustawy: Chciałbym zapytać: Na jakim etapie są te projekty ustaw?

Widać bowiem, że na dzień dzisiejszy jedyną rzeczą, którą robi krajowy zasób mieszkaniowy, jest odpowiadanie, że nie kupuje gruntów. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Mam informację, że już mamy połączenie. Dziękuję. Mogę mówić? Tak. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed zadaniem pytania mam taką uwagę, że jeżeli głównym problemem są kredyty, to nie znaczy, że państwo ma coś robić, tylko znaczy, że banki mają za dużo pieniędzy, a ludzie za mało. Przechodząc do pytania. Mam pytanie, wy tego nie zrozumiecie, ja mówię do posłów, ale ja mówię do ludzi. Skąd państwo wiecie, że mieszkań jest za mało?

To jest czysto subiektywne i nie ma obiektywnej miary tego, ile potrzeba mieszkań. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Chciałem zapytać, czy w najbliższej przyszłości rząd przewiduje jakiekolwiek instrumenty, które będą wspierały Polaków i ułatwiały uzyskanie kredytu.

Tych mieszkań by nie było, gdyby nie ich praca.

Dziękuję bardzo. Mamy połączenie? Tak. Dziękuję. Chciałam zapytać, jaka jest relacja proponowanej ustawy do niedawno uchwalonej przez nas ustawy o popieraniu niektórych form mieszkalnictwa, która przewiduje fundusz dopłat dla gmin: w przypadku zakupu lokali - 50%, w przypadku wybudowania lokali - 80%. Czy taka dopłata będzie obowiązywała w świetle tej ustawy, kiedy nastąpi zamiana gruntu za lokal?

Czy to będzie lex specialis wobec ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy nie? Podsumowując, wydaje się, że zapisy tej ustawy są korzystne wyłącznie dla deweloperów, a nie są korzystne dla gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Chciałem tylko dopowiedzieć, bo nie zdążyłem, że poproszę od ministerstwa o odpowiedź na piśmie na zadane przeze mnie pytanie dotyczące konsekwencji kosztowych w długiej perspektywie czasowej w związku z rozlewaniem się zabudowy. Dziękuję bardzo. Na pytania postawione przez panie i panów posłów odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pani minister Anna Kornecka. Bardzo proszę, pani minister. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Zaczynając od początku, program „Mieszkanie+” zawsze zakładał współpracę z samorządami i zawsze obejmował nie tylko filar rynkowy, ale także filar społeczny.

Jeśli zastanowimy się nad tym, czy jest to, tak jak państwo użyliście takiego sformułowania, przerzucenie odpowiedzialności na gminy, to trzeba jasno powiedzieć: my tej odpowiedzialności nie przerzucamy na gminę. Program „Mieszkanie+” od początku zakładał w sobie współpracę gmin. Nie da się wykonywać jakichkolwiek inwestycji mieszkaniowych, inwestycji w nieruchomości bez współpracy pomiędzy państwem a samorządami. Mało tego, w przygotowywanych przez nas regulacjach jest niezliczona liczba instrumentów wspierających gminy w prowadzeniu inwestycji. Mamy pakiet mieszkaniowy społeczny, czyli właśnie tę ustawę, która już w tym momencie poszła do podpisu prezydenta. Proszę państwa, wsparcie w wysokości 80% kosztów inwestycji - w zasadzie nie można wyobrazić sobie silniejszego instrumentu, który pozwoli gminie podjąć decyzję o rozpoczęciu danej inwestycji. Mało tego, odchodzimy od zasady refinansowania. Te pieniądze są dostępne już od samego początku tej inwestycji, w związku z czym nie trzeba angażować ogromnych środków związanych właśnie z realizacją inwestycji na początku, co stanowi główną barierę dla gmin w realizowaniu inwestycji. Naszym celem jest współpraca w programie „Mieszkanie+” zarówno strony rządowej, jak i przede wszystkim samorządowej. Projekt: lokal za grunt jest elementem całego programu. Nie da się go rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście osobnego projektu ustawy. Bardzo państwu wszystkim też dziękuję za docenienie jakości samego projektu i przedstawionych w nim rozwiązań, pomimo tych wszystkich wątpliwości, które zaraz postaram się rozwiać.

W naszym kraju w ubiegłym roku oddano do użytkowania 207 tys. mieszkań.

Ten poziom na pewno zostanie osiągnięty ze względu na to, że wiemy, że w 2020 r. ten wskaźnik będzie jeszcze wyższy niż te dotychczasowe 207 tys. Adresujemy je nie tylko do tej części rynkowej, ale przede wszystkim wspieramy - i program: lokal za grunt również wspiera - budownictwo komunalne, budownictwo czynszowe i budownictwo społeczne. Nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na aspekcie rynkowym. Program: lokal za grunt powoduje takie odblokowanie nieruchomości, możliwości, które do tej pory nie były przez gminy wykorzystywane ze względu właśnie na te bariery, o których powiedziałam wcześniej, czyli bardzo duże koszty inwestycyjne. Pojawiło się takie pytanie o to, czy nie obawiamy się tego, że będą mogły skorzystać z tego tylko mniejsze miasta. Nie, nie obawiamy się tego. To jest właśnie program realizowany z myślą też o mniejszych ośrodkach miejskich.

Nie chodzi o to, by gminy kupowały go po cenie rynkowej, natomiast w przypadku tego typu inwestycji, inwestycji w nieruchomości, zawsze mamy do czynienia z ryzykiem, że ktoś na tym zarobi bądź straci. W związku z tym nie da się ryzyka inwestycyjnego całkowicie wyeliminować i w tym zakresie żadne przepisy ustawowe nie będą niczego zabezpieczały. Pojawiło się pytanie o to, dlaczego gmina nie ma żadnych przepisów, które by powodowały, że to mienie pozostaje przy gminie. Co do zasady w programie: lokal za grunt uczestniczymy jakby w montażu, który zakłada, że to gmina daje swój grunt. Nie jesteśmy w stanie w takim razie nakładać na gminę jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli ten grunt jest jej własnością i tak to zostało pomyślane, że to jest w zasadzie inwestycja ze strony gminy. W związku z tym można by było powiedzieć, że nakładanie takich obowiązków na gminę w tym zakresie byłoby jakimś nowym ograniczeniem w stosunku do gminy, więc jeżeli grunt jest gminny, czyli nieruchomość jest gminną własnością, to nie widzieliśmy uzasadnienia dla tego, żeby tutaj wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia. Pojawiło się pytanie o grunty objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo decyzjami o warunkach zabudowy. Te decyzje o warunkach zabudowy muszą być wydane na wniosek gminy, w związku z czym już są inwestycjami, o których przeznaczeniu w innym trybie, ale również uprzednio, zadecydowano. Dlaczego nie promujemy tylko i wyłącznie tych nieruchomości, które są położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Dlatego że adresujemy ten program też do gmin wiejskich, a w większości gmin wiejskich mamy do czynienia z taką sytuacją, że tych planów nie ma. Zaznaczam, że nie chodzi o grunty, które nie posiadają w ogóle żadnego przeznaczenia. One posiadają wydaną przez gminę i na rzecz gminy, zgodnie jakby z jej preferencjami co do zakresu inwestycji, decyzję o warunkach zabudowy.

W związku z tym, jeżeli gmina wprowadzi np. kwestie dotyczące standardów mieszkania albo właśnie kryteriów dla najemców bądź wysokości czynszu, to wówczas również będziemy mieli to tylko i wyłącznie w uchwale rady gminy. Jeśli chodzi o Krajowy Zasób Nieruchomości, to trzeba też powiedzieć, że Krajowy Zasób Nieruchomości dysponuje 900 ha własnych gruntów. Z tego, co wiem, na dzień dzisiejszy zawarte jest ok. 70 porozumień, a w planach jest jeszcze kolejne 30, czyli ok. 100 porozumień z gminami. Mamy ogromne zainteresowanie gmin, zarówno tą społeczną częścią pakietu mieszkaniowego, jak i inwestycją „lokal za grunt” Samorządy są tym bardzo zainteresowane, natomiast są zainteresowane zarówno te mniejsze, jak i duże miasta.

Dziękuję, pani minister. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Rafała Webera o przedstawienie dokumentu. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Przedstawiam sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w roku 2019. Dokument zawiera wnikliwą analizę wszystkich elementów, które wpływają na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokument obrazuje w ten sposób również największe zagrożenia dla życia ludzkiego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Są tutaj zgromadzone dane statystyczne, którymi dysponuje Policja, ale także inne instytucje, które są członkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tak że to, co robi wrażenie, to właśnie jego szczegółowość, jego zawartość. Ze zgromadzonych danych wynika, że miniony rok był kolejnym, w którym zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. W roku 2019 odnotowano: 30 288 wypadków - jest to spadek o 4,4% w stosunku do roku 2018, 35 477 osób rannych - jest to spadek o 5% w stosunku do roku 2018. 10 633 osoby ciężko ranne i jest to spadek o 3% w stosunku do roku 2018. I trzeba podkreślić, że to są najniższe w historii prowadzenia danych statystycznych wartości. Rok 2019, na podstawie tych trzech parametrów, był najbezpieczniejszym rokiem, jeżeli chodzi o ruch drogowy w Polsce. W poprzednim roku aż 2909 osób straciło życie na drogach i jest to wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2018. Struktura udziału wypadków, które miały miejsce w roku 2019, jest podobna do tej z lat poprzednich. Największy odsetek stanowiły wypadki z udziałem pieszych - 23,1%, następnie spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu - ponad 20%, spowodowane przez młodych kierowców - 17%, z udziałem rowerzystów - ponad 14%, z udziałem nietrzeźwych - 9%, z udziałem motocyklistów - ponad 8%, i w wyniku najechania na drzewo - blisko 5%. Dotychczasowe działania prewencyjne skoncentrowane wokół „Narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013-2020” przyniosły wiele pozytywnych zmian dzięki zaangażowaniu członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także wielu kluczowych partnerów.

Ale - no właśnie jest to: ale z dużym wykrzyknikiem - stan bezpieczeństwa ruchu drogowego jest cały czas niezadowalający i takie stanowisko będzie przez rząd, przez Ministerstwo Infrastruktury podtrzymywane, dopóki choć jedna osoba będzie ginąć na skutek wypadku drogowego w Polsce. W roku 2019 zapłaciliśmy jako społeczeństwo najwyższą cenę za zdarzenia drogowe w postaci ofiar - przypominam tę liczbę - 2909. To oczywiście dramat ludzi i ich bliskich, z którym przychodzi mierzyć się przez kolejne lata. I aby skutecznie przeciwdziałać tym dramatom, konieczne jest dalsze prowadzenie systematycznych działań na wielu płaszczyznach, poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, w szczególności, po pierwsze, poprzez inwestycje w bezpieczne drogi, po drugie, poprzez zmiany w przepisach prawa, które pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, i po trzecie, poprzez edukację i wzmocnienie świadomości wszystkich tych, którzy korzystają z polskich dróg, nie tylko kierowców, ale również pieszych, rowerzystów, wszystkich tych, którzy na (Dzwonek) co dzień korzystają z infrastruktury drogowej. Szanowni państwo, jestem otwarty na pytania, jestem otwarty na państwa ocenę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku poprzednim. Jeżeli będzie do tego okazja, to w drugiej części swojej wypowiedzi nie tylko na te pytanie odpowiem, ale powiem szerzej o tych działaniach, które w poprzednim roku były realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, ale także opowiem o naszych planach na tą bliższą przyszłość i planach na taką perspektywę 4-, a także 10-letnią. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam. Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Infrastruktury w sprawie rządowego dokumentu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.”, druk nr 585. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierowała w dniu 4 września 2020 r. powyższy dokument do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia. Komisja Infrastruktury, po rozpatrzeniu tego dokumentu na posiedzeniu 7 października 2020 r. oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, bardzo merytorycznej, konstruktywnej i konkretnej, wraz z odpowiedziami pana ministra Rafała Webera, wnosi, by Wysoki Sejm raczył przyjąć dokument z druku nr 585. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Piotr Król. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do druków nr 585 i 667, czyli do przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r. Dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.” zwiera szereg danych dotyczących m.in. rodzaju wypadków, liczby ofiar śmiertelnych, ciężko rannych, rodzaju pojazdów, płci ofiar, zachowań kierowców, pieszych, rowerzystów, wraz z wnioskami i rekomendacjami co do podejmowania kolejnych działań naprawczych. Szczegółowo opisuje również działania realizowane przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz instytucje współpracujące z Krajową Radą BRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedstawione analizy zostały opracowane na podstawie danych pochodzących Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji prowadzonego przez Komendę Główną Policji. Dokładne analizy danych statystycznych, wyników badań i analizy dotyczące zachowań uczestników ruchu drogowego oraz oceny ryzyka bycia ofiarą wypadku drogowego prezentowane w dokumencie pozwalają na określenie głównych profili sprawców, ofiar oraz przyczyn zdarzeń drogowych. Dane dotyczące wypadkowości w 2019 r. zostały porównane z zeszłorocznymi danymi, a także ujęte w trendzie obserwowanym na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dodatkowo w dokumencie zawarto mapy obrazujące zestaw wskaźników zagrożeń dla różnych kategorii wypadków drogowych we wszystkich województwach w 2019 r. W raporcie zasygnalizowane zostały zagrożenia i wyzwania, jakie pojawiają się w trendach demograficzno-statystycznych BRD, a mianowicie narastanie problemu zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w grupie 60+. Raport wyraźnie pokazuje, że Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podejmowała w 2019 r. kolejne konkretne kroki w celu spajania działań i wysiłków różnych podmiotów, jak również - przez sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - realizowała konkretne projekty i działania mające na celu zwiększenie siły i efektywność oddziaływania na poprawę BRD. Przykładem mogą być ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg i Policji czy również wdrożenie w 94 powiatach o najwyższych wskaźnikach zagrożenia ogólnopolskich warsztatów dla seniorów 60+ we wsparciu samorządów lokalnych, Policji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Istotnym elementem wymienianym w raporcie są informacje o poczynionych w 2019 r. badaniach naukowych i publikacjach z zakresu BRD. Dzięki wiedzy naukowej oraz dostępnych danych statystycznych zawartych w dokumencie możliwe jest określenie najważniejszych czynników zagrożenia, jak również programowanie działań na kolejne lata.

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Maciej Lasek. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wnioski z analizy ostatniego raportu na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego są niepokojące. 4 lata to też wystarczająco długi czas, żeby ocenić podjęte działania mające poprawić stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Przyjrzyjmy się więc, jaki jest ten stan.

To dobrze. To samo można powiedzieć o liczbie osób rannych w wypadkach drogowych. Liczba osób ciężko rannych w wypadkach również stopniowo maleje w prawie stałym tempie od 2011 r.

Niestety nie ma szans na osiągnięcie celu wyznaczonego w „Narodowym programie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2013-2020”

Zmniejszyła się też liczba wypadków będących wynikiem najechania na pieszego. To jest koniec dobrych wiadomości. Liczba ofiar śmiertelnych jest od 5 lat na tym samym poziomie, przy czym przez ostatnie 2 lata rośnie.

Gdyby ten trend był zachowany, to osiągnięto by zakładany cel. Niestety w 2016 r. ten trend się zatrzymał. Nie ma tutaj żadnej poprawy. Dlaczego? Liczba kolizji istotnie rośnie.

To jest 30-procentowy wzrost od roku 2014. Nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie w raporcie. Niepokojące są też statystyki dotyczące osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych z udziałem pieszych. Po pierwsze - jest to najczęstszy rodzaj wypadku, w którym dochodzi do śmierci niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Po drugie - tendencja jest rosnąca dla obu tych statystyk i to już od roku 2010. Dużo wypadków śmiertelnych z udziałem pieszych jest spowodowanych zbyt dużą prędkością kierującego - aż 48%. Są to wypadki, których liczbę zdecydowanie można byłoby zmniejszyć. 770 osób zginęło w 2019 r., ponieważ kierujący jechał zbyt szybko. Jeśli chodzi o wypadki motocyklistów, to dzieje się coś bardzo niedobrego. Liczba motocyklistów, którzy zginęli w 2019 r., jest najwyższa od 10 lat, a od 2015 r. zwiększyła się o prawie 50%. Co jest tego przyczyną? Podobna sytuacja dotyczy ofiar śmiertelnych w wypadkach spowodowanych przez kierujących samochodami ciężarowymi.

Może nie wszystkich - część spada.

Oczywiście nie da się stwierdzić, jaki byłby skutek zaprzestania tych działań, ale ogólna poprawa jest niewielka. Co jest tego powodem? Myślę, że najwyższy czas, panie ministrze, na krytyczną analizę przyjętych w 2016 r. rozwiązań i zaproponowanie nowych kierunków działań profilaktycznych. Na koniec - prędkość. Z raportu instytutu transportu drogowego z 2016 r. wynika, że po zlikwidowaniu gminnych fotoradarów aż o 46% wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w tych miejscach. Naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego do dzisiaj [[Dzwonek]] nie uregulowaliśmy dziury w systemie automatycznego nadzoru nad przekraczaniem prędkości. Przepisy ruchu drogowego są jednoznaczne, definiują dopuszczalną prędkość na drogach. Bezpieczeństwo to również stosowanie się do obowiązujących przepisów, nawet jeżeli niektórym kierowcom należy o tym przypominać. Bo na końcu chodzi o czyjeś życie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedstawiony raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r. znów pokazują, że Polska pod względem bezpieczeństwa na drogach jest daleko w tyle na tle krajów Unii Europejskiej. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak organizacji, która sprawnie działałaby na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z pewnością taką instytucją nie jest. Korzystanie z polskich dróg, mimo tylu lat wdrażania różnych rozwiązań, to nadal walka o przetrwanie. Obok bułgarskich i rumuńskich polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Według niniejszego raportu rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, o 4,4% w stosunku do 2018 r., ale nie spadła liczba ofiar śmiertelnych, wzrosła o 1,6% w stosunku do poprzedniego roku. I to są prawdziwe tragiczne dane. Najważniejszym bowiem miernikiem skuteczności polskiego rządu w tym zakresie jest liczba ofiar śmiertelnych, a ta z roku na rok wzrasta. Według najnowszego raportu Komisji Unii Europejskiej w 2019 r. w Polsce na 1 mln mieszkańców w wypadkach zginęło 77 osób, dla porównania w Czechach - 58, w Estonii - 39, a w Szwecji - 22 osoby. Skąd taki wynik? Oczywiście częścią winy za taki stan rzeczy należy obarczyć niewystarczającą sieć dróg ekspresowych, infrastrukturę, autostrady, obwodnice. Miasto Kalisz czeka na swoją obwodnicę już kilka dekad. Jest jednak coś jeszcze. Już w 2015 r. Bank Światowy analizował kwestię wypadków na polskich drogach. Rekomendował Polsce stworzenie silnej organizacji odpowiedzialnej za poprawę bezpieczeństwa na drogach. Można zapytać: Dlaczego? Zdaniem Banku Światowego instytucja, która mogłaby zmienić rzeczywistość na polskich drogach, powinna być ponadpartyjna, stabilna i na tyle władna, by rozliczać z działań poszczególne ministerstwa oraz instytucje. Ponadpartyjność to kluczowa wartość, bo działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa muszą być zaplanowane na lata i nie powinno się ich paraliżować żadną zmianą władzy. Postulatu tego nie spełnia Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organ ten, założony, tak jak wspomniałam, w 2002 r., działa przy ministrze do spraw transportu. Przy takiej koncepcji trudno się spodziewać, że krajowa rada będzie krytycznie analizowała działania Ministerstwa Infrastruktury czy rozliczała inicjatywy Policji działającej pod kontrolą ministra spraw wewnętrznych. W efekcie rada ta jest instytucją fasadową. Niestety Polska od lat pozostaje negatywnym przykładem na unijnej mapie bezpieczeństwa drogowego. Nie poprawi się to, póki nie zostanie właśnie powołana prężna organizacja, która będzie niezależna od politycznych nacisków i sprawnie będzie organizować nie tylko kampanie społeczne o ograniczonym zasięgu. Należy się nad tym bardzo poważnie zastanowić, bo te raporty, informacje, które nam państwo przedstawiają, niewiele zmieniają, a na drogach nadal będą ginąć ludzie i nadal będziemy pod tym kątem na końcu krajów Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Stefan Krajewski w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska dotyczące przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów dokumentu: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r.” wraz ze stanowiskiem komisji, druk nr 585 i druk nr 667. Z raportu tego wynika, że 2019 r. zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. Jak zaznaczał pan minister i na posiedzeniach komisji, i dzisiaj, trzy z czterech podstawowych danych mówiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego są bardzo pozytywne. Ale też pan minister mówił, że te dane są najniższe wśród wartości mierzonych w historii monitorowania wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Te wszystkie inwestycje, w dużej mierze z dofinansowaniem ze środków unijnych, miały służyć z jednej strony przyspieszeniu i poprawieniu płynności ruchu, a z drugiej strony zwiększeniu bezpieczeństwa zarówno kierowców, pasażerów, jak i pieszych. Chyba wszyscy widzą drogi, przy tych drogach ścieżki rowerowe, drogi, które mają służyć do obsługi, tzw. drogi techniczne. Tego jest coraz więcej. Natomiast chciałoby się powiedzieć, że może być zawsze lepiej, i do tego powinniśmy wszyscy dążyć, bo chodzi nie tylko o inwestycje, ale też działania Policji.

Bo wczoraj, jadąc tutaj, mijałem się z 15 dużymi samochodami Policji, które wracały z Warszawy z akcji, zamiast być tam, na miejscu. Z drugiej strony drogówka. Zamiast łapać piratów drogowych, wręczać mandaty tym, którzy faktycznie dopuszczają się dużych wykroczeń czy wręcz przestępstw na drogach, najłatwiej ścigać krnąbrnych rolników, którzy wyjechali traktorami na drogi. Tych łatwo zatrzymać, bo wolno jadą. Tych też bezpiecznie zatrzymywać, bo nie będą strzelać, nie będą stawać do bójki, tylko pokornie przyjmują mandaty, kładą uszy po sobie. Dziękują panu policjantowi za to, że ich zatrzymał, i jadą dalej. Wracają do domu trochę biedniejsi o ten mandat, który dostali przed chwilą. Ale naprawdę to nie są żarty, bo Policja powinna być wykorzystywana do zupełnie innych celów niż stanie na Żoliborzu.

To wszystko dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Nie może być tak, że się dba o bezpieczeństwo jednego największego Polaka, a wszyscy mają do czynienia z niebezpieczeństwem na drogach. Panie pośle, do rzeczy. Już o tych morderstwach za dużo słyszeliśmy na tej sali, pani poseł. Rozmawiamy o bezpieczeństwie wszystkich Polaków i trzeba to bezpieczeństwo podnosić, inwestycje powinny być. W tym raporcie nie znalazłem takich rzeczy, które przekonałyby mnie, przekonały też nasz klub do przyjęcia tego raportu.

Nie? Okej, rozumiem. Bardzo proszę. Ten raport po raz kolejny potwierdza długookresowy trend spadkowy liczby wypadków na drogach przy stałym wzroście liczby samochodów i użytkowników i dróg. Trzeba sobie uzmysłowić skalę tego sukcesu.

Rząd może się do tego przyczyniać, budując lepsze drogi. Z tym jest różnie, ale jednak pewien postęp jest i to też w tych statystykach w pewnym stopniu widać.

W tym segmencie funkcjonują różne nieprzemyślane akcje społeczne, które de facto sprowadzają się do zapraszania pieszych pod koła samochodów, testowania hamulców i do niebezpiecznych zachowań.

Nie analizujemy systemowo, co potem z tymi danymi się dzieje w wyniku weryfikacji sądowej. Takich danych w tym raporcie nie ma. Dane końcowe, różne wnioski, słupki są tylko tak dobre, jak dane wyjściowe, jeśli na początku mamy arbitralną decyzję, często niczym nieumotywowaną, to na końcu otrzymujemy mało przydatny wykres. Te dane są podatne na liczne nadinterpretacje, a nawet im sprzyjają, bo tam mamy właśnie to stale powtarzane od 10 lat porównanie z założonym arbitralnie, z sufitu wziętym spadkiem, który chcielibyśmy osiągnąć, co oczywiście nie może się udać, ponieważ zakłada się, że liczba wypadków będzie spadała równomiernie, nawet szybciej niż wcześniej. Wiemy, że im bardziej zbliżamy się do zera, tym wypadków będzie ubywało wolniej.

Po raz kolejny, drugi rok z rzędu, jak słucham tej dyskusji, pojawia się ta sama absurdalna sugestia, że mamy jakiś problem związany z tym, że rośnie liczba wypadków w grupie 60+. To jest absolutnie logiczne i nieuniknione, że jeśli dana grupa staje się liczniejsza w społeczeństwie, to liczba wypadków z jej udziałem będzie proporcjonalnie rosła.

Nie będzie to niczym dziwnym, tylko będzie skutkiem zmiany w demografii. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta. Zamykam listę osób chcących zadać pytanie. Jako pierwszy pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Finiszują prace związane z pierwszeństwem pieszych. Bardzo dobrze, że jeśli chodzi o trzy projekty, nad którymi pracujemy, to prawdopodobnie jutro zostaną sformułowane sprawozdania Komisji Infrastruktury. To czas najwyższy, ponieważ, Wysoka Izbo, w 2019 r. zginęło 2909 osób, ale w tym 793 pieszych. Chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że na przejściu dla pieszych zginęło 250 osób, a 3646 osób zostało rannych. To jest wielkie wyzwanie. Odsetek osób starszych w społeczeństwie co roku rośnie. I także dla nich powinniśmy zagwarantować jasne, dobre przepisy, które będą ich chroniły w tym miejscu, które jest przygotowane dla nich wszystkich.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym w tym punkcie ponowić pytanie, które zadałem rok wcześniej i niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Czy przygotowując ten dokument, analizując przyczyny wypadków drogowych, wzięli państwo również pod uwagę, czy jakikolwiek wpływ na przyczynę powstawania wypadków drogowych może mieć używanie przez kierującego pojazdem jadącym z naprzeciwka świateł do jazdy dziennej zamiast powszechnie stosowanych przez większość kierowców świateł mijania? Przepisy w naszym kraju oczywiście zezwalają na używanie świateł do jazdy dziennej w ciągu dnia przy dobrej widoczności, ale bywa z tym różnie. Wielu polskich kierowców nadal się skarży, że samochody jadące na światłach dziennych są w momencie wymijania słabiej widoczne niż pojazdy z włączonymi światłami mijania. Stąd moje pytanie: Czy używanie świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania ma wpływ na zwiększoną liczbę wypadków? Czy państwo przeprowadziliście taką analizę? Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Maciej Lasek, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jak ważne jest bezpieczeństwo w okolicach przejść dla pieszych, nikomu dzisiaj nie trzeba tłumaczyć. Niestety wiele przejść dla pieszych poza terenem zabudowanym i w ciągu dróg krajowych jest słabo doświetlona, słabo lub źle oznakowana. Bardzo często spotykamy się z brakiem ograniczenia prędkości w okolicach takich przejść poza terenem zabudowanym. Sam znam kilka takich miejsc, gdzie notorycznie dochodzi do wypadków. W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z pytaniem: Czy został przeprowadzony audyt stanu oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych, a jeżeli tak, to z jaką liczbą takich miejsc mamy do czynienia i jak wygląda harmonogram usuwania tych nieprawidłowości? Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska, kolejne pytanie. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Przykład - chodnik w miejscowości Chmieleń przy drodze krajowej nr 3 w kierunku Zgorzelca. Ruch rośnie bardzo szybko. Ciężki transport towarowy. Tymczasem mieszkańcy proszą, apelują, protestują, ja piszę ciągłe interpelacje i zapytania - i nic. Nie ma zgody na budowę chodnika za kilkaset tysięcy złotych. W tak wrażliwym miejscu. Odpowiedź jest ta sama: priorytety, autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice. Czy państwa naszego nie stać na kilkaset tysięcy złotych, żeby dać szansę i zapewnić bezpieczeństwo Polakom? Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, klub Lewica. Czy mamy połączenie? Mamy? Nie mamy. W takim razie pan poseł Marek Rząsa, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle, do zadania pytania. Panie Ministrze! Tymczasem z danych Komendy Głównej Policji wynika, że ich liczba wzrasta, podobnie jak liczba zabitych i ciężko rannych w wyniku takich wypadków. Niestety obowiązujące przepisy prawne związane z tego rodzaju wypadkami rozmywają kompletnie odpowiedzialność, począwszy od tzw. odpowiedzialności Skarbu Państwa, poprzez samorządy, zarządców dróg, a kończąc na kołach łowieckich. Zdarzenie drogowe z udziałem dzikiego zwierzęcia praktycznie uniemożliwia uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania za szkody zdrowotne i materialne wywołane wskutek tego wypadku lub wymaga bardzo długiej i kosztownej drogi sądowej. Każdy z kierowców, którzy przeżyli takie zdarzenie, wie, że nawet przy bardzo zachowawczej jeździe uniknięcie zdarzenia jest niemożliwe, a powstałe szkody są znaczne. W związku z tym pytam pana ministra: Czy ministerstwo posiada aktualne pełne dane na temat liczby zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt? Ilu kierowców w skali roku ubiega się o odszkodowania od ww. podmiotów z tytułu szkód poniesionych w wyniku niezawinionej kolizji ze zwierzęciem na drodze? Jaki procent wniosków jest odrzucany i jakie są główne przyczyny ich odrzucania? Mamy połączenie zdalne z panią poseł Katarzyną Kretkowską. Dziękuję bardzo. Chciałam zadać pytanie dotyczące sytuacji w województwie wielkopolskim.

Liczba wypadków wzrosła o 20%, a śmiertelnych o 7%, jest duży udział rowerzystów w tych wypadkach. Chciałam zapytać, czy rząd skieruje środki do województwa wielkopolskiego na jakąś kampanię społeczną uczulającą zarówno pieszych, jak i rowerzystów, w kwestii oznakowania, jeżdżenia z oznakowaniem i uważania na drogach. A z drugiej strony Wielkopolska czeka na osiem obwodnic. Dziękuję. Pan poseł Franciszek Sterczewski, klub Koalicja Obywatelska. Zapraszam do zadania pytania. Dziękuję. Wysoka Izbo! Zaproponowane przez rząd zmiany dotyczące ruchu drogowego są oczywiście krokiem w dobrą stronę, ale sytuacja wymaga nie kroku, ale zdecydowanego skoku i odważnych działań. W 2019 r. na drogach zginęło niespełna 3 tys. osób, a ponad 10 tys. zostało ciężko rannych. Każdy wypadek powoduje koszty społeczne, obciążenie systemu ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych, tymczasem kwoty mandatów nie zmieniły się od ponad 20 lat, choć przez ten czas znacznie wzrosły wynagrodzenia. Kilka lat temu w Finlandii były dyrektor Nokii za przekroczenie prędkości otrzymał mandat w wysokości 116 tys. euro, bo tam wysokość mandatów uzależniona jest od dochodów. W Polsce za takie narażenie innych na niebezpieczeństwo zapłaciłby 100 lub 200 zł. Każdy dzień trwania tej patologii powoduje, że na drogach kolejne osoby tracą życie i zdrowie. Kiedy rząd przedstawi propozycję zmian [[Dzwonek]] kwot mandatów karnych? Polskiego społeczeństwa nie stać na utrzymywanie raju dla piratów drogowych. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Proszę o zadanie pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Muszę powiedzieć, że systematycznie podczas tej debaty pytam o to, czy będą zmiany w kierunku zapewnienia bezpiecznych przejść dla pieszych. Nie chodzi tutaj o rozwiązania prawne, tylko raczej o rozwiązania techniczne: po pierwsze, o odpowiedni program, po drugie, o odpowiednie zmiany w przepisach. Muszę powiedzieć, że po tych kilku latach mówienia pierwszy raz usłyszałem od pana ministra kilka dni temu na posiedzeniu komisji, że będzie program dotyczący polepszenia warunków bezpieczeństwa dla pieszych na przejściach. To chcę powiedzieć. Natomiast mam pytania o dalsze kroki, czyli kwestię wymagań technicznych na budowanych czy przebudowywanych drogach, zwłaszcza w obszarach zabudowanych. Natomiast (Dzwonek) przejścia dla pieszych są zlokalizowane często na drogach, gdzie są dwa pasy. Te, powiedzmy, warunki techniczne powinny być trochę zaostrzone. Czy ministerstwo prowadzi w tym kierunku prace? miał być program fotoradarów, które łapią przejeżdżających na czerwonym świetle. Czy ministerstwo zamierza zaostrzyć w końcu warunki dla tych pojazdów? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie. Co więcej, niestety ten stan w ogóle się nie zmienia. W 2015 r. na drogach zginęło 2938 osób, w 2016 r. - 3026, w 2017 r. - 2831, w 2018 r. - 2862 i w 2019 r. - ponowny wzrost - 2909 zgonów. W ciągu tych 5 lat w sumie na polskich drogach zginęło 15 tys. osób.

Eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego mówią jasno: z jednej strony prewencja, z drugiej strony inwestycje drogowe. My zgłosiliśmy poprawki do budżetu na kolejny rok: obwodnice Mszany Dolnej, Gorlic, Grybowa i Limanowej, węzeł w Krzyszkowicach. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska, z kolejnym pytaniem. Panie Ministrze! Ten raport ma luki, które warto czy też trzeba uzupełnić. Pierwsze dotyczy dzieci i młodzieży, osób nieletnich, które giną na drodze. Nie znalazłam żadnej informacji na ten temat, a to przecież informacja niezmiernie ważna. Znalazłam informację, w jakich programach ta grup wiekowa uczestniczy, ale to jest mniej ważne.

To jest grupa przestępców niezmiernie groźnych. Niezmiernie groźnych właśnie dla młodzieży, dla dzieci, którzy szczególnie w małych miejscowościach podróżują i muszą podróżować do szkoły. W tej chwili nie, ale wróci ten czas, kiedy będą, mamy nadzieję. Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Andrzej Grzyb, Koalicja Polska. Zapraszam, panie pośle. Proszę o zadanie pytania. Panie Ministrze! Nie mogę się zgodzić z takimi opiniami, które tu słyszałem, że nie zmienia się stan polskich dróg. Być może to nie jest uprawnione stwierdzenie, bo jednak tych inwestycji było sporo. W tej materii jest potrzebny istotny postęp. W szczególności dotyczy to oczywiście rozdzielenia ruchu pieszego i ruchu pojazdów.

To jest oczywiście bardzo pożądany kierunek. Natomiast myślę, że to wszystko musi być połączone z prewencją. Nie da się tego zrobić bez prewencji. W szczególności wydaje mi się, że zaniechany został program kształcenia dzieci z zakresie ruchu.

Dziękuję, panie pośle. Kolejne pytanie zada pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Podobnie jak pan poseł Grzyb, panie ministrze, nie mogę się zgodzić z tym, że mamy jakąś stagnację. Wszyscy eksperci mówią, że bezpieczeństwo poprawia się wraz z ilością nowo budowanych dróg, pod warunkiem że są kryteria budowy, które uwzględniają poprawę bezpieczeństwa i natężenie ruchu. I dam, panie ministrze, przykład drogi krajowej nr 11 z Poznania na północ. Jest to odcinek między Poznaniem a Obornikami. Nie ruszyliście w ostatnich latach nic.

Proszę o refleksję w tym zakresie. Budować drogi trzeba w oparciu o mądre kryteria. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Od kilku lat liczba ofiar wypadków śmiertelnych w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie. To tak jakby co roku znikała w Polsce jedna mała miejscowość. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, ale od końca. Liczba ofiar śmiertelnych w Polsce na 1 mln mieszkańców to 77 osób, a średnia unijna wynosi 51. Od krajów, które są w czołówce, dzieli nas przepaść, dwukrotna przepaść. Mam więc pytanie, proszę o bardzo konkretną odpowiedź: Jakie konkretne rozwiązania zaproponuje polski rząd, aby ograniczyć liczba wypadków śmiertelnych na polskich drogach? Przypomnę, że pan premier Mateusz Morawiecki podczas swojego exposé deklarował, że przygotuje projekt ustawy wzmacniający bezpieczeństwo pieszych. Zajęło mu to rok czasu. Także ustawa przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej leżała w zamrażarce. Proszę, aby rozwiązania, o których, mam nadzieję, [[Dzwonek]] za moment usłyszymy, były szybciej niż za rok. Dziękuję, panie pośle. Chciałbym się w swoim pytaniu odnieść do słów pana ministra Webera, który stwierdził, że najważniejsze jest to, aby nikt na naszych polskich drogach nie ginął w wypadkach samochodowych. Panie ministrze, jak to się ma do faktów? Otóż raport NIK z 2020 r. dotyczy „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych”, pan na pewno go zna, realizowanego przez generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. NIK zarzuca, że przygotowanie programu jest nierzetelne. Modernizowano niewłaściwe drogi, realizacja jest nieskuteczna, a afekty mizerne. Właściwie od 2015 r. liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach się nie zmieniła. To jest ok. 2900 osób co roku. I stąd moje pytanie: W jaki sposób rząd chce zmienić, zmodyfikować powyższy program, aby jego skuteczność była wyższa? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Kolejne pytanie zada pan poseł Marek Rutka, klub Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Nawet najlepsza zmiana przepisów nie zwiększy umiejętności kierowców, a trzeba jasno podkreślić, że to one są przyczyną wypadków w największym stopniu. Sama poprawa jakości dróg nie wyeliminuje wypadków, bo polscy kierowcy są po prostu źle szkoleni. Trzeba jasno powiedzieć, że poruszanie się po autostradach, które z założenia miały być bezpieczniejsze niż drogi o niższych kategoriach, w istocie takie nie jest. W systemie szkolenia w czasie kursów na prawo jazdy brakuje szkoleń z jazdy po autostradzie. Polscy kierowcy zarówno na rodzimych autostradach, jak i poza granicami kraju nie umieją właściwie włączać się do ruchu, płynnie zmieniać pasów ruchu czy właściwie oznaczyć pojazdu, który uległ awarii. Stąd moje pytanie: Kiedy program kursu na prawo jazdy zostanie poszerzony o praktyczną umiejętność jazdy po autostradach? Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z analizy porównawczej stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwach w 2019 r. wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim, podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymał się najwyższy odsetek wypadków spowodowanych nadmierną prędkością oraz najechaniem na drzewo. W strukturze wypadków dominują wypadki z udziałem pieszych. To pokazuje, jak bardzo ważny jest to problem i jak bardzo brakuje rozwiązań w tym obszarze. Dlatego też mam pytanie: Jakie konkretne działania oraz inwestycje zamierza podjąć pan minister infrastruktury, by zmienić te niechlubne statystyki na Warmii i Mazurach i Powiślu? Brakuje również moim zdaniem w tej analizie wniosków, czyli tak naprawdę konkretnych rozwiązań, by zmienić te statystyki. Dziękuję. Kolejne pytanie, koło Konfederacja, pan poseł Artur Dziambor. Bardzo proszę. Słucham niektórych posłów i mam takie wrażenie, że niektórym przyświeca coś, co nazwałem kiedyś antysamochodzizmem. Tu u niektórych również słyszę takie jakby marzenia o tym, że jakiekolwiek ministerstwo czy jakikolwiek rząd jest w stanie sprawić, że ludzie przestaną ginąć na ulicach. To nie jest do końca możliwe. To tak jak mamy statystykę, że co roku ginie ileś osób, które zostały stratowane przez hipopotamy, tak? Tak już po prostu niestety jest. Natomiast chciałem bardzo konkretną rzecz poruszyć, może niezwiązaną z tematem, ale jednak, blokady na koła samochodowe zakładane przez straż miejską. Rozumiem, że samochód potrafi stanąć czasem tak, że blokuje ruch, potrafi stanąć tak, że blokuje chodnik i trzeba potem przejść dookoła, potrafi stanąć w miejscu nielegalnym, i rozumiem też, że powinien dostać za to mandat, więc mandat można wystawić i ten kierowca może być oczywiście (Dzwonek) tym mandatem obarczony, ale ta blokada sprawia, że on tam stoi w tym nielegalnym miejscu godzinę, 2 godziny, dłużej. Może po prostu zrezygnujmy z tego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska, z kolejnym pytaniem. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W województwie łódzkim jest kilka dróg krajowych, które wymagają pilnej interwencji w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsza droga to droga nr 48 od Tomaszowa Mazowieckiego przez Spałę, Inowłódz, gminę Poświętne. Tutaj od lat mieszkańcy domagają się interwencji w kwestii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naprawdę tragiczne zdarzenia mają miejsce zarówno na słynnym odcinku w gminie Poświętne, na wysokości Anielina, jak i w Spale, którą wszyscy w Polsce dobrze znają. Pytanie: Co ministerstwo w tej kwestii zamierza zrobić w najbliższym roku?

Dobrze by było, gdyby zaplanowano pieniądze na obwodnicę, natomiast domagają się także innych kwestii poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. I jeszcze droga nr 72, odcinek od Rawy Mazowieckiej przez Złotą. Czy także w tym miejscu doczekają się ludzie chociażby chodników? Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo! Bezpieczeństwo drogowe to nie tylko stan infrastruktury drogowej i przepisy prawa, ale także to, jak zachowują się służby państwowe i jak podchodzą do przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym. Dlatego konkretne pytanie, panie ministrze: Ile było w 2019 r. wypadków ruchu drogowego z udziałem służb państwowych, Służby Ochrony Państwa, Policji i innych służb? Wielokrotnie mieliśmy informacje, że do takich wypadków dochodziło z udziałem właśnie kierowców SOP-u. Dokładnie też pamiętamy, jak kolumna - wtedy ówczesnego BOR-u - stratowała seicento w Małopolsce, kolumna z panią premier. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja.

Raport nie zawiera takich danych, które by do tego uprawniały.

Dlaczego ją robicie? Drugie pytanie: Dlaczego ten raport zestawia dane dotyczące liczby wypadków z Polski z danymi z innych krajów, bez odniesienia do danych porównujących gęstość dróg o klasie autostrady czy drogi ekspresowej?

Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Cezary Grabarczyk, Koalicja Obywatelska, zada kolejne pytanie. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przejazdy drogowo-kolejowe to miejsca szczególnie niebezpieczne. Dochodzi tam do kolizji, które najczęściej mają poważne skutki, jeśli chodzi o ofiary. Co trzeci, co czwarty wypadek na przejeździe kończy się śmiercią. I wprawdzie w 2019 r. było mniej wypadków na przejazdach, ale za to - więcej wypadków ze skutkami śmiertelnymi. Rozwiązanie problemu przejazdów kolejowych to domena ministra infrastruktury, bo ani PLK, ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad samodzielnie nie rozwiążą tych problemów.

To jest idealne rozwiązanie, tam trzeba większych środków budżetowych (Dzwonek), ale to się opłaci, nie tylko dlatego że będzie mniej ofiar, ale także dlatego że nie będzie konieczności zwalniania przed przejazdami kolejowymi dla pojazdów szynowych. Zwiększy się przepustowość. Wszyscy na tym zyskają. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę o zadania pytania, pani poseł. Wysoka Izbo! Przy okazji naszej debaty o bezpieczeństwie ruchu drogowego chciałabym dopytać o kwestię powszechnej dostępność do szkolenia i egzaminu na kartę rowerową dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Wiemy, że rower staje się coraz popularniejszym, codziennym środkiem transportu. To dotyczy i dorosłych, i dzieci. Wiem, że w dokumencie było napisane, że w 2019 r. miała być zrobiona analiza dostępności szkolenia oraz egzaminu na kartę rowerową, ale z powodu braku danych ta analiza nie została przeprowadzona i już samo to sugeruje, że obecny system związany z kartą rowerową nie działa. Dlatego chciałam zadać pytania: Czy mimo braku tej analizy ministerstwo planuje reformę dotyczącą karty rowerowej?

Bardzo proszę, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W dużych miastach bardzo często mamy ulice dwupasmowe i przy przejściach dla pieszych bywa tak, że jeden z samochodów ustąpi pieszemu pierwszeństwa, a drugi nadjeżdża z ogromną prędkością.

Bardzo częste są np. w Warszawie przypadki wyprzedzania i omijania samochodów w rejonie przejścia dla pieszych. Za brak biletu w komunikacji miejskiej kara wynosi 260 zł.

Chciałabym państwa zapytać, czy przewidują państwo jakikolwiek fundusz na poprawę bezpieczeństwa przejść dla pieszych dla samorządów, bo Warszawa robi taki audyt od 5 lat i wydała na poprawę bezpieczeństwa drogowego pieszych ponad 100 mln zł. Dziękuję, pani poseł. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na postawione przez panie i panów posłów pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Rafał Weber. Zapraszam, panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo.

To dobrze, w taki sposób ta debata powinna wyglądać.

Wszyscy wpływamy na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Szanowni Państwo!

W tej chwili ten program to wartość 165 mld zł. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększyliśmy finansowanie na ten program o prawie 60 mld zł właśnie po to, żeby zrobić to szybciej, żeby zrobić więcej. Wszystkie te inwestycje, które są poza limitem, są przygotowywane.

Środki finansowe były potrzebne, żeby je projektować i budować.

Obwodnice. Program budowy 100 obwodnic” - 28 mld zł.

Tak że uruchomimy kolejne narzędzie wspierające tego typu inwestycje.

Tak że w sytuacji, kiedy Rada Ministrów przyjmie specjalną uchwałę, na mocy której powoła ten program, a stanie się to na początku przyszłego roku, będziemy go realizować.

Tysiące zadań na drogach gminnych i powiatowych jest już w realizacji.

Szanowni Państwo! Myślę, że on sam w sobie został - na początku to powiedziałem - przygotowany w sposób rzetelny, merytoryczny. Statystyka odzwierciedla wszystko to, co działo się na polskich drogach w roku 2019. Rok 2020 siłą rzeczy przez epidemię, przez zmniejszenie ruchu był zdecydowanie lepszy. Mam nadzieję, że wprowadzone przepisy prawa i inwestycje, które są realizowane i będą realizowane w przyszłości, przyczynią się do tego, że w kolejnych latach będziemy mieli do czynienia ze spadkiem liczby wypadków, liczby ofiar i rannych, a polskie drogi będą bezpieczniejsze. Dziękuję bardzo, panie ministrze.

Ale w wystąpieniu ministra nie było. Panie Ministrze! Chodziło mi o porównanie.

Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Dariusz Klimczak w trybie sprostowania, choć nie był wymieniany przez pana ministra.

Pan minister zasugerował, że niebawem ruszy dofinansowanie w ramach tego instrumentu. Czy pan już wie, że takie dofinansowanie będzie prowadzone w trybie naboru ciągłego, czy będzie ogłoszony konkurs i czy w przyszłym roku takie miejscowości, które liczą na obwodnice w ciągu drogi wojewódzkiej, będą mogły liczyć na konkurs lub nabór ciągły, jeśli chodzi o dofinansowanie. Bardzo proszę, panie ministrze.

W ramach zmian poszerzamy wartość funduszu o 3 mld zł, a także dopuszczamy nowych beneficjentów do tego funduszu. To są m.in. zarządcy infrastruktury wojewódzkiej, czyli dróg wojewódzkich, którzy będą mogli ubiegać się o środki na budowę obwodnic tychże dróg. Nabór będzie prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury. Na ten cel mamy przeznaczone 2 mld zł, no i zobaczymy. Jeżeli wniosków będzie mniej i będą środki, które będą do dyspozycji w dalszych latach, to będziemy ten nabór powtarzać. Wszystko będzie uzależnione od liczby wniosków, ale też od jakości wniosków. Wbrew temu, co państwo sugerują, co państwo mówią, jakość wniosku, uzasadnienie danej inwestycji wpływają na uzyskanie dofinansowania. Czekamy na bardzo dobre wnioski zarządców dróg wojewódzkich i wtedy takie wsparcie będzie udzielone. Dziękuję bardzo. Komisja Infrastruktury wnosi o przyjęcie dokumentu z druku nr 585. Sprzeciwu nie słyszę.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Marka Gróbarczyka o przedstawienie informacji. Bardzo proszę, panie ministrze.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawozdanie dotyczące ochrony brzegów morskich zawiera kompleksowy zakres inwestycji w zakresie realizacji ochrony brzegów morskich. Wartość tego projektu wynosi 34 mln zł.

Przede wszystkim dotyczy one naprawy, remontu nabrzeży, wykonania wszelkiego rodzaju umocnień, realizacji zadań w zakresie przede wszystkim przeciwdziałania erozji i podniesienia bezpieczeństwa w tym zakresie. Jest to niezwykle ważne działanie również w kontekście ochrony infrastruktury portowej, dostępowej tak dużych portów, jak i małych portów na całym wybrzeżu. Przyszły program będzie realizowany również w oparciu o środki, czyli ma określone finansowanie, i w ramach inwestycji, które zostały i zostaną zakwalifikowane do tego typu działań. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych programów w zakresie przede wszystkim utrzymania bezpieczeństwa i swobodnego dostępu do plaż, które również ten program określa oprócz infrastruktury, a więc są to: refulacja, odtwarzanie plaż i zabezpieczenie swobodnego dostępu do morza w celach turystycznych.

Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę pana posła Dariusza Wieczorka o przedstawienie stanowiska komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze!

Przedstawiony druk i przedstawione dokumenty wynikają z ustawy z dnia 28 marca o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”

W związku z czym można powiedzieć, że to zadanie zostało zrealizowane. Do tego sprawozdania załączone zostały dwie tabelki - jedna tabelka dotyczy wykonania zadań za rok 2019, druga to planowane zadania na rok 2020. W trakcie dyskusji komisja, posłowie i posłanki zwrócili uwagę, po pierwsze, na to, że jeżeli chodzi o konkretne zadania, to rzeczywiście zdecydowanie potrzeby są większe niż te 34 mln zł. Były konkretne przykłady konkretnych inwestycji i pytania dotyczące działań prowadzonych w ramach tego programu, szczególnie jeżeli chodzi o obszar województwa zachodniopomorskiego.

W związku z czym sugestią ze strony komisji, posłów było to, ażeby być może zastanowić się, czy nie powinno się zwiększyć zakresu zadań, jeżeli chodzi o ochronę brzegów morskich i całej linii brzegowej w Polsce.

Cały program jest szacowany na poziomie 911 mln zł, takie były zapowiedzi.

Natomiast komisja niewątpliwie będzie pana ministra i ministra finansów namawiała do tego, ażeby spróbować zwiększyć nakłady na te zadania. Generalnie konkluzja zawarta w druku nr 538 jest taka, że komisja rekomenduje Wysokiemu Sejmowi przyjęcie informacji z wykonania w 2019 r. programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2020. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy wystąpi pan poseł Artur Szałabawka w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stanowiska dotyczącego informacji na temat realizacji „Programu ochrony brzegów morskich” w roku 2019, zawartej w druku sejmowym nr 319. Rok 2019 był kolejnym, w którym urzędy morskie realizowały „Program ochrony brzegów morskich” Urzędy morskie w Gdyni, w Słupsku i w Szczecinie miały do wykorzystania te 34 mln.

Jest to największe wykonanie „Programu ochrony brzegów morskich” w ostatnich latach. Informacja zawiera wymagane elementy, które minister właściwy do spraw gospodarki morskiej winien przedłożyć Sejmowi RP, a mianowicie informację o realizacji w roku ubiegłym zadań wynikających z programu oraz harmonogram na rok następny. Przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informacja z realizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w sposób spójny pokazuje zakres wykonywanych oraz planowanych prac w związku z ochroną brzegów morskich, zaś zawarte w informacji dane dotyczące wydatkowania środków finansowych na ochronę brzegów morskich nie budzą żadnych zastrzeżeń, my to widzimy.

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2019 r. zaplanowano w ramach programu realizację zadań na 8 km linii brzegowej, a wykonano zabezpieczenia brzegu morskiego na łączną długość prawie 13 km. Powyższe wykonanie wartości miernika osiągnięto w wyniku wprowadzenia nowych zadań do realizacji w trakcie roku budżetowego, co dowodzi sprawnej realizacji programu w 2019 r. Na realizację w 2020 r. w ramach programu zaplanowano 34 mln zł, z przeznaczeniem na wykonanie sztucznego zasilania plaż, przebudowę i budowę umocnień brzegowych oraz monitoring brzegu morskiego. Powyższe świadczy o tym, że ochrona brzegów morskich jest realizowana konsekwentnie i systemowo. W związku z powyższym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę, aby Wysoki Sejm przyjął przedstawiony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dokument dotyczący informacji na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” w 2019 r., wraz z harmonogramem na 2020 r., zawartych w druku nr 319. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Tadeusz Aziewicz przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jak już wspomniano, rozpatrywana informacja jest efektem zapisów ustawy z 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego zatytułowanego „Program ochrony brzegów morskich” Głównym celem tego programu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe brzegów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń, zapewnienie stabilizacji linii brzegowej oraz zapobieganie zanikowi plaż. W budżecie państwa na rok 2019 na jego realizację zabezpieczono wydatki w łącznej kwocie 34 mln zł. Planowane działania obejmowały sztuczne zasilanie plaż, budowę, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu oraz monitoring. Powyższe wydatki zostały zrealizowane prawie w pełnej kwocie. Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą wskaźnikiem realizacji programu w danym roku jest długość linii brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskami erozji i powodzi od strony morza liczona w kilometrach. W 2019 r. zaplanowano realizację zadań w wymiarze 8 km linii brzegowej. Na koniec 2019 r. wykonano zabezpieczenia brzegu morskiego przed zjawiskami erozji i powodzi od strony morza na łącznej długości ponad 12 km. Wyższe wykonanie wartości miernika osiągnięto w wyniku wprowadzenia w trakcie roku budżetowego nowych zadań. Wysoki Sejmie! W trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wysłuchaliśmy szczegółowych informacji poszczególnych urzędów morskich. W dyskusji pojawił się natomiast bardzo ciekawy problem przyspieszonego podnoszenia się poziomu wód i potrzeby przygotowania się państwa na długofalowe zmiany. Odpowiedzi przedstawicieli rządu miały charakter ogólny i na pewno wrócimy do tego tematu w nieodległej perspektywie. Tradycyjnie przy okazji dyskusji o ochronie brzegów morskich chcę zwrócić uwagę na potrzebę zabezpieczenia, zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie Klifu Orłowskiego w Gdyni, gdzie w nieodległej przeszłości miały miejsce niebezpieczne osunięcia. Dotychczas obyło się bez ofiar, ale ochrona życia i zdrowia masowo spacerujących tam obywateli jest ciągle poważnym wyzwaniem. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z Gdyni, zwracając uwagę na zagrożenia, postulują m.in. ułożenie w odległości około 200 m od brzegu kamiennych falochronów podwodnych. Dzięki temu po niezbędnej reflacji, czyli nadsypaniu piasku wydobywanego przy okazji pogłębiania kanałów portowych, plaża jako naturalny wygaszacz fal nie tylko będzie znacznie szersza, ale też będzie mogła się utrzymać. Mam świadomość, że w przypadku klifu krzyżują się kompetencje dwóch ministrów: środowiska oraz infrastruktury, dlatego po jednym z niebezpiecznych osunięć próbowałem zainteresować tym problemem prezesa Rady Ministrów, niestety bez pozytywnego efektu. Premier i przedstawiciele wspomnianych resortów ciągle chowają głowy w piasek. Przeczuwam, że podobnie będzie, jeżeli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek. Na razie zabezpieczenie klifu polega na tym, że stoją tam lub leżą tablice z ostrzeżeniami, a ludzie nadal chodzą po osuwisku. Ponieważ „Program ochrony brzegów morskich” w 2019 r. został wykonany zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym, a plan na 2020 r. nie wzbudził kontrowersji, w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie przedstawionych dokumentów. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Stanowisko klubu Lewica przedstawi. Panie Ministrze! Trzeba dodać, że gestorem środków na ten szczytny cel, na ten program, są urzędy morskie. Urzędy morskie bronią brzegów morskich nierzadko z narażeniem życia, jak to miało miejsce w Dziwnowie, kiedy pod pracującą koparką eksplodowała pamiątka z II wojny światowej. Niestety często można odnieść wrażenie, że bronią oni tych brzegów nie tylko przed żywiołami, ale także przed ludźmi, przed nami, przed mieszkańcami, turystami i inwestorami, panie ministrze. Samorządy, doceniając nakłady pracy poniesione przez urzędy morskie, jednym głosem mówią, że współpraca jest żadna. Jakiekolwiek uzgodnienia z tą instytucją są bezcelowe, jest to zwykła droga przez mękę. Można odnieść wrażenie, że ochrona brzegów morskich to sztuka dla sztuki, a jedynym celem tej pracy jest zaspokojenie ambicji zawodowych urzędników za to odpowiedzialnych. Dochodzi do tego, że nawet naprawa starych, kilkudziesięcioletnich chodników - dojść i zejść na plażę, panie ministrze - jest czymś niewykonalnym przez urząd morski. Nie można się dogadać, nie można dostać pozwoleń, nie można nic zrobić, chociaż samorządy chcą robić to za własne pieniądze. Dochodzi do sytuacji takich, że np. w Rewalu w roku 2019 przez cały sezon było zamknięte jedno z trzech zejść na plażę, bo urząd morski nie pozwalał go naprawić. Zastanawiające jest również, że urzędy morskie same interpretują obowiązujące prawo i wydają decyzje te prawo zmieniające, jak choćby Prawo budowlane, i skracają ustawowy termin posadowienia budynków nietrwale związanych z gruntem z ustawowych Kończąc, panie ministrze: „Program ochrony brzegów morskich” prowadzicie dobrze, dlatego będziemy głosować za jego przyjęciem, jednak więzi społecznych na terenie nie budujecie. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nieco ponad 100 lat temu Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego, a przez ten czas poczyniliśmy wiele starań, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał bałtyckiego Wybrzeża. Wybrzeże to wyzwania, zwłaszcza te związane z bezpieczeństwem mieszkańców pasa nadmorskiego i tamtejszego przemysłu, a co za tym idzie, miejsc pracy, a także z turystyką, tak bardzo ważną i dla mieszkańców tamtego regionu, i dla nas. Ale Wybrzeże to także unikalna na skalę europejską przyroda, liczne cenne siedliska roślin, to miejsca bytowania zwierząt, to ujścia rzek z całym ekosystemem, unikalny krajobraz.

Powinniśmy znaleźć więc takie rozwiązania, które sprawią, że pogodzimy te dwie sprawy, rozwój i budowę infrastruktury, zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie obszarów naturalnych. Z informacji przedstawionej przez pana ministra wynika, że w roku 2019 zrealizowane zostały takie zadania jak sztuczne zasilanie plaż, budowa, remont i utrzymanie trwałych umocnień brzegu oraz monitoring. To kluczowe zadania, dobrze, że jest ten harmonogram, dobrze, że są one realizowane. Ale czy to oznacza, że brzegi morza są w Polsce dostatecznie chronione? Nie. Bo chciałabym podkreślić, że nasze polskie Wybrzeże jest w bardzo trudnej sytuacji. Sięgnijmy do raportu NIK-u z 2019 r. dotyczącego ochrony terenów nadbrzeżnych. W 22 na 45 badanych decyzji wydanych przez dyrektorów urzędów morskich dotyczących wykorzystania pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegów w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochroną środowiska stwierdzono nieprawidłowości, które upoważniały do sformułowania negatywnej oceny realizacji tych zadań, ale decyzje zostały sformułowane pozytywnie. Przykłady: Ustronie Morskie i apartamentowce oddalone 10 m od morza czy obiekt, który w Piaskach na Mierzei Wiślanej powstał na niskim podmokłym brzegu Zalewu Wiślanego, co grozi jego podtopieniami. To tylko dwa przykłady, ale jest ich tak naprawdę dziesiątki. Naruszanie pozwoleń, stawianie czasowych zabudowań w pasie nadmorskim to stała praktyka. Przyczyna - lekkomyślność państwa polskiego, chciwość wielkiego biznesu, niewłaściwy nadzór, poddawanie się presji deweloperskiej, niemyślenie o konsekwencjach i to nie tylko tych dla przyrody, ale przede wszystkim dla ludzi i ich bezpieczeństwa. To nie jest tak, że my możemy sobie zamykać oczy na dewastację środowiska naturalnego, uważając, że nas to w żaden sposób nie dotyka. Dlatego że niszczenie klifów, wydm, krajobrazu morskiego, oprócz tego, że jest dewastacją środowiska naturalnego, prędzej czy później przełoży się na atrakcyjność tych terenów dla turystów. Rabunkowy rozwój kosztem przyrody, kosztem krajobrazu może skutkować tym, że turyści będą po prostu wybierać inne kierunki podróży, a mniej turystów to mniej miejsc pracy, to bezrobocie, brak perspektyw i frustracja. Czy chcemy skończyć jak Bułgaria czy Hiszpania, gdzie zabetonowane są setki kilometrów wybrzeża?

Ważne jest więc to, aby urzędy morskie, aby samorządy dobrze współpracowały, ale również stosowały przepisy prawa, bo mamy narzędzia, dzięki którym możemy zatrzymać tę katastrofę. A najmłodszym Polkom i Polakom będziemy w stanie wtedy dać morze w jego najlepszej odsłonie, a nie zabetonowane, zniszczone i w dodatku grożące ich bezpieczeństwu. Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Debata w sprawie ochrony brzegów morskich nie może się odbyć bez odniesienia się do najważniejszych wyzwań w najbliższych latach. Takim wyzwaniem jest też przekop Mierzei Wiślanej. Tego typu inwestycja zakończy wieloletni spór z Rosją, zwiększy dostępność drogi wodnej na linii Hel - Elbląg i przyczyni się w walnym stopniu do rozwoju transportu morskiego. To trzeba pamiętać. Polsce brakuje niestety długofalowej strategii polityki morskiej i bezpieczeństwa morskiego. Pytanie, co będzie dalej.

W tym miejscu trzeba jednak zwrócić uwagę również na inny problem. Dzisiejsza polityka ochrony brzegów morskich często wyklucza się niestety z racjonalną polityką turystyczno-rekreacyjną, np. gwiazdobloki, które są pod wodą, czy gęste falochrony na plażach, to jest zabójstwo walorów polskich plaż, np. w aspekcie sportów wodnych.

Bo sezon plażowy trwa 2–3 miesiące, a niektóre sporty wodne można uprawiać znacznie dłużej, zacząć już wiosną, skończyć nawet jesienią. Przykładem takiego trochę braku racjonalności jest np. okolica portu w Łebie, gdzie falochrony i gwiazdobloki spowodowały w zasadzie wygaszenie fali, a to wygaszenie fali spowodowało brak turystów, którzy przyjechaliby np. uprawiać windsurfing czy kitesurfing. Dlatego Konfederacja postuluje współpracę i konsultacje - bo to jest naprawdę istotne - z gminami, z rybakami, z wodniakami i właśnie ze środowiskami sportowymi. Chcemy naturalnej ochrony brzegów morskich, ale bez wielopoziomowych konsultacji dotyczących konkretnych odcinków to może oznaczać zaszkodzenie samemu sobie. Program ochrony brzegów morskich” nie jest - całe szczęście - wymierzony w polskie rybołówstwo. Jest to branża - o tym też należy wspomnieć przy okazji - bardzo mocno poszkodowana przez politykę unijną, np. przez Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich”, który finansował w zasadzie trwałe i tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej. Krótko mówiąc, Unia Europejska wprost przekupywała polskich rybaków, aby porzucili pracę w tej branży. Polska przestała odgrywać w sektorze rybołówstwa poważną rolę, a bogactwo naturalne Morza Bałtyckiego przypadło po prostu innym państwom członkowskim - wszystko w imię unijnej solidarności, solidarności, na której po prostu cierpimy. Należy także nadmienić, że z racji zakazu połowów np. dorsza w Bałtyku, w wyniku niskiej populacji, część organizatorów np. połowów turystycznych straciła swoje źródło utrzymania i pomimo odszkodowań i pomimo obietnic od pana, panie ministrze, ci ludzie stracili po prostu źródło swojego utrzymania. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapomniało jakimś cudem o tym, aby wesprzeć także tych ludzi w momencie, w którym dostali zakazy połowowe.

Dziękuję, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Jarosław Rzepa. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W pierwszych słowach chciałbym podziękować, panie ministrze, za to, co się stało w roku 2019, tym wszystkim, którzy realizowali te zadania. Bo muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o plan i wykonanie, został on zrealizowany, tak jak państwo założyliście. Natomiast pewnie moglibyśmy być bardziej ambitni, jeśli chodzi o kwoty wydatkowania, ale to też jest uwarunkowane - jak państwo wiecie - wieloma rzeczami.

Na tym obszarze, panie ministrze, myślę, że trzeba jeszcze wiele poprawić. Samorządy jednak funkcjonują w tym obszarze. Oczywiście mamy wiele różnych interesów, tutaj mamy zabezpieczenie, tutaj mamy turystykę, tutaj mamy rybactwo. Musimy znajdować często złoty środek. Chciałbym, panie ministrze, bardzo serdecznie prosić pana o to, żeby w tych wszystkich inwestycjach, które państwo planujecie, element konsultacji i wsłuchania się w interesy samorządów był mocno, mocno słyszany. Bo to jest bardzo, bardzo istotne.

Mam inne zdanie na ten temat, szanowni państwo, bo chciałbym widzieć ten zwrot, jeżeli chodzi o gospodarkę. Natomiast, panie ministrze, pozwoli pan, że z tego miejsca mimo wszystko jednak nawiążę do jednego tematu, który mnie bardzo boli. Szanowni państwo, za kilka dni będziemy mieli święta, a kilkanaście dni temu, panie ministrze, również pana decyzjami 201 osób dostało wypowiedzenia. Mogliśmy mówić o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, mogliśmy mówić o ochronie tego miejsca, mogliśmy mówić o ochronie tych stoczniowców.

Wydaje mi się, że jest jeszcze czas na to, żeby cofnąć tę złą decyzję, żeby uratować to miejsce, żeby znaleźć środki na to, żeby stocznia remontowa Gryfia w Szczecinie mogła realizować swój bardzo ambitny - słuszny, ale ambitny, panie ministrze - plan, ale nie kosztem tego samego zakładu. To są polscy stoczniowcy. Uważam, że. Zresztą pan, panie ministrze, niejednokrotnie na posiedzeniu komisji gospodarki morskiej mówił o tym, że dzisiaj się nie buduje statków, dzisiaj się remontuje. Jeżeli dzisiaj zamykamy, niszczymy jak gdyby. Nie wiem, czy zespół portów znajdzie sposób na to. Może dzisiaj nie mają tego pomysłu, ale panie ministrze, wydaje mi się, że polską racją stanu jest dzisiaj ratowanie tych miejsc pracy, ratowanie tych stoczniowców, dawanie szansy, a nie odsyłanie ich, powiedzmy sobie, do domu. Od dzisiaj nie świadczą przez 3 miesiące pracy, później dostaną odprawy. To będzie kilka milionów złotych straty, panie ministrze, straty. Wolałbym, panie ministrze, żebyśmy szukali rozwiązań. Zachęcam do tego, bo ci ludzie naprawdę chcą tam pracować, chcą pracować dla Gryfii, w ramach tego zakładu - jeżeli nie ma woli, żeby to rozdzielić - nadal funkcjonować. Jeszcze raz, panie ministrze, z tego miejsca proszę w imieniu tych ludzi.

Panie ministrze, bardzo proszę. A za to, co pan zrobił w tym obszarze, o którym dzisiaj mówimy, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie pośle. Przechodzimy do zadawania pytań. Zamykam listę osób chętnych do zadania pytania. Wyznaczam czas na pytanie - 1 minuta. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2019 r. nie zostawił suchej nitki na tym, jak dyrektorzy urzędów morskich podchodzili do obowiązków w zakresie troski o wykorzystanie nadmorskiego pasa technicznego. Raport NIK zdecydowanie najgorzej ocenił funkcjonowanie Urzędu Morskiego w Słupsku, który w ciągu 12 lat nie korygował granicy tego pasa. W konsekwencji szeregu nieprawidłowości rząd PiS zlikwidował Urząd Morski w Słupsku, a dyrektora odpowiedzialnego za wskazane w raporcie NIK błędy uczynił wicedyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni. Nie chcę jednak poświęcać zbyt wiele czasu polityce kadrowej rządu tzw. dobrej zmiany. Mam jedno konkretne pytanie. Chodzi o stan linii brzegowej na odcinku Ustka - Orzechowo.

Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Oni naprawdę dobrze robią swoją robotę i każdy to mówi, ale jeszcze raz mówię: współpracy z samorządami nie ma żadnej.

Powiedział: nie i koniec. Tam sobie ludzie nogi łamią. Nie możemy zrobić zejścia na plażę dla ludzi niepełnosprawnych czy na ludzi z wózkami. Dziękuję bardzo. Pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Nie ma pana posła. Pan poseł Mirosław Suchoń, również Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Oczywiście to, co widać, jest ważne, bo jeżeli poprawimy część brzegu, na który wszyscy patrzą, to będzie to widoczny efekt jakiejś działalności. Natomiast mamy do czynienia z takim typowym, powiedziałbym, rządowym podejściem do tego, co trzeba zrobić, czyli rozwiązujemy problemy, które widać, natomiast te, których nie widać, ignorujemy. Takim problemem, którego nie widać na pierwszy rzut oka, jest kwestia zanieczyszczeń strefy przybrzeżnej tymi rzeczami, które pozostały po wojnie. Teraz one są o tyle niebezpieczne, że ich nie widać, natomiast upływ czasu powoduje, że stanowią coraz większe zagrożenie i dla środowiska, i dla ludzi. W związku z tym pytanie: Czy ministerstwo w ogóle planuje jakikolwiek program, który miałby dotyczyć (Dzwonek) w jakiś sposób tych zanieczyszczeń pozostałych po wojnie? Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Dziambor, koło Konfederacji. Panie Ministrze! Przeczytam list: Przez kilka lat prowadziłam firmę związaną z połowem. Od 1 stycznia 2020 r. został wprowadzony całkowity zakaz połowów na Morzu Bałtyckim we wschodniej części. Minister Gróbarczyk obiecał nam wielokrotnie pomoc, jednak nic z tego nie wyszło. Obiecywał, że nasze statki będą zezłomowane i dostaniemy odszkodowania, by móc od podstaw zacząć nową działalność. Daliśmy się, brzydko mówiąc, urobić. Nasza sprawa trafiła do kancelarii premiera, który też zadeklarował się nam pomóc. Jednak później otrzymaliśmy pismo, że możemy się starać o to, o co starać mogą się przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej. Jak mamy to zrobić, skoro nasze działalności są zamknięte z dniem, w którym wprowadzono zakaz? Nas w ogóle to nie dotyczy. Od 3 miesięcy nie mamy z czego żyć - to było parę miesięcy temu - zostaliśmy z długami, ratami, statkami, które stoją w portach i niszczeją. Nie spłacamy ich, bo nie mamy z czego. Chciałbym, panie ministrze, zapytać: Co pan zrobił w sprawie takich właśnie armatorów? Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Marek Gróbarczyk. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałbym państwu podziękować za to, że kierowaliście tyle ciepłych słów pod adresem urzędów morskich, które realizują te inwestycje, a z drugiej strony za to, że poprzecie państwo nasze sprawozdanie, bo ono faktycznie jest dobre. Czy można było zrobić więcej? Oczywiście. Przecież wybrzeże wymaga wielu, wielu inwestycji, jeśli chcemy należycie je przywrócić czy też chronić.

Myślę, że na pewno znajdziemy złoty środek, ale apelowałbym o to, aby również samorządy wykazały daleko idącą współpracę i dialog.

Z drugiej strony nie jest też prawdą to, że armatorzy wędkarscy nie otrzymali wsparcia.

Oczywiście kwestia niewybuchów jest rzeczą dla nas niezwykle ważną. Powstał specjalny zespół, ale ten zespół również działa na forum międzynarodowym, w ramach HELCOM, który jest organizacją międzynarodową i którego główną agendą jest właśnie praca nad usunięciem niewybuchów. Chodzi o miliardy dolarów, które trzeba wyłożyć na tę okoliczność, a więc chyba nikt nie znajdzie takiego finansowania w Polsce. Temat jest monitorowany, przede wszystkim w zakresie pozostałych wraków. Nie ma żadnego zagrożenia, nic się z nich negatywnego nie wydobywa, a wszelkie obszary, które mogą stanowić zagrożenie, jeśli chodzi o naruszenie tych wraków, są specjalnie oznaczone i monitorowane, aby nie dochodziło tam do żadnych ingerencji. W Łebie jest tzw. podwodna rafa, która zabezpiecza naturalną refulację brzegów. Tylko wejście do portu jest obłożone gwiazdoblokami, a więc to nie jest prawda, to wybrzeże jest przepiękne i bardzo cenione przez turystów.

A więc nasza ingerencja jest zdecydowanie ograniczona. Czy sprawozdawca komisji. Nie ma go. Wobec tego zamykam dyskusję. Komisja wnosi o przyjęcie Informacji z wykonania w 2019 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2020, zawartych w druku nr 319. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Bartosza Grodeckiego o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie oraz Szanowni Panowie Posłowie! Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi rejestr informatyczny nieruchomości, a także udziałów i akcji nabytych przez cudzoziemców bez zezwolenia, jak też na podstawie wymaganych zezwoleń oraz wydanych decyzji - w postaci komputerowej bazy danych. Umożliwia on monitorowanie tendencji w zakresie nabywania nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców oraz analizę skali zainteresowania poszczególnych grup podmiotów nabywaniem konkretnych rodzajów nieruchomości oraz stopień zainteresowania takimi nieruchomościami w poszczególnych województwach. Prowadzony rejestr to baza danych zawierająca w szczególności informacje dotyczące nieruchomości, w stosunku do których minister wydał decyzję, nieruchomości nabytych przez cudzoziemców oraz dane spółek, w których cudzoziemcy nabyli lub objęli akcje lub udziały. Dane te wynikają przede wszystkim z nadsyłanych aktów notarialnych, postanowień sądowych, a także uzyskiwane są w toku prowadzonych przez organ czynności wyjaśniających oraz prowadzonych postępowań administracyjnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż mimo zakończenia wszystkich okresów przejściowych - to dosyć istotna informacja - w których wymagane było zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji nadal jest organem uprawnionym do monitorowania obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców poprzez właśnie prowadzenie niniejszego rejestru. Wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., ustawy chyba najdłużej obowiązującej w obecnym porządku prawnym, są dostosowane do wymogów prawa europejskiego, a w szczególności do swobody przepływu kapitału przysługującej podmiotom z państw właśnie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej. O ile zatem cudzoziemcy spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej mają obowiązek co do zasady uzyskać zezwolenie na nabycie każdej nieruchomości, o tyle cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej od 1 maja 2016 r. mogą swobodnie, a więc bez zezwolenia, nabywać nieruchomości w naszym kraju. W sytuacji, gdy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia - głównie dotyczy to obywateli Ukrainy czy Białorusi, to jest najczęstsza grupa występująca o wydanie takich zezwoleń - minister spraw wewnętrznych i administracji wydaje stosowną decyzję. W przypadku nieruchomości rolnych konieczna jest w tym wypadku opinia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Porównując dane sprawozdawcze, należy stwierdzić, że zarówno liczba wydanych w 2019 r. zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców, jak i powierzchnia nieruchomości objętych zezwoleniami nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzednich 2 lat. Powyższe wynika m.in. ze zwiększającej się liczby wniosków w zakresie zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wpływających do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szanowni Państwo! Podsumowując, należy stwierdzić, że prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji rejestr umożliwia rzeczywiście monitorowanie pewnych tendencji w zakresie nabywania nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców oraz analizę skali zainteresowania poszczególnych grup podmiotów nabywaniem konkretnych rodzajów nieruchomości oraz stopień zainteresowania takimi nieruchomościami w poszczególnych województwach. Niemniej aby był on prowadzony, konieczne jest - właściwie, w sposób rzetelny - zapewnienie rzetelnego przekazywania przez sądy i notariuszy dokumentów dotyczących nabycia przez cudzoziemców nieruchomości, akcji i udziałów, tak aby ten rejestr zawierał rzeczywiście dane jak najbardziej kompletne. Szanowni Państwo! Kończąc to swoje krótkie wystąpienie, przedstawiając sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2019 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwracam się z uprzejmą prośbą o jego akceptację. Dziękuję Wysokiemu Sejmowi za poświęcony czas i uwagę. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Teraz proszę pana posła Pawła Hreniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2019 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, druk nr 292. Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu skierował w dniu 25 marca 2020 r. powyższe sprawozdanie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Paweł Hreniak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister spraw wewnętrznych i administracji, wypełniając zobowiązanie zawarte w ustawie, przedstawił sprawozdanie, w którym w szczególności znalazły się informacje o wydanych zezwoleniach, ich rodzaju oraz terytorialnym rozmieszczeniu nabytych nieruchomości. Przedłożył również informację na temat transakcji w zakresie nieruchomości dokonanych przez obywateli m.in. państw Unii Europejskiej. Należy przypomnieć, że co do zasady obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ale w sprawozdaniu przedłożonym przez pana ministra, jak już wspomniałem, znalazły się również informacje o transakcjach dotyczących nieruchomości nabytych przez obywateli, którzy nie muszą uzyskać zezwolenia u ministra właściwego. Z przedstawionego dokumentu wynika, że w 2019 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło 767 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach. Jest to poziom wzrostu, który jest stały od kilku ostatnich lat. Spośród wniosków o udzielenie zezwolenia ponad 400 dotyczyło nieruchomości gruntowych, 108 zezwoleń zostało wydanych na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych, a 171 zezwoleń - na nabycie lokali mieszkalnych. We wszystkich tych zestawieniach przeważającą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Widać, że obywatele tego państwa coraz bardziej wiążą się z Polską, m.in. poprzez zakup nieruchomości. Należy nadmienić, że największe zainteresowanie zezwoleniami na zakup nieruchomości gruntowych przez obywateli państw trzecich dotyczyło województw lubelskiego i mazowieckiego, a pod względem kryterium zakupu lokali były to województwa pomorskie i zachodniopomorskie. Podstawowym źródłem informacji, o tym już mówił pan minister, o nabytych przez cudzoziemców nieruchomościach są dla ministerstwa wypisy aktów notarialnych przesyłanych przez notariuszy. Na notariuszy nałożono obowiązek przesyłania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wypisów takich aktów. To tworzy oczywiste problemy. Jak wynika z wyjaśnień, podjęto już za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiednie środki dyscyplinujące w stosunku do notariuszy. Myślę, że ważne jest, żeby zaznaczyć w tym miejscu, że problem został zauważony i jest w trakcie rozwiązywania.

Jak wynika z przedstawionych informacji, w zdecydowanej większości grunty zakupione przez tę grupę osób są przeznaczone na inwestycje, ale też na cele mieszkaniowe. Ten wskaźnik jest podobny, na poziomie ostatnich kilku lat. Zresztą podobnie jest w przypadku zakupu przez osoby prywatne. Niezwykle ważne jest, aby monitorowanie odbywających się transakcji z udziałem cudzoziemców, zarówno tych, którzy muszą posiadać zezwolenie, jak i tych, których zakup jest rejestrowany, odbywało się w sposób rzetelny i na podstawie aktualnych danych. Dlatego też klub Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje pozytywnie wszelkie działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości, które w tym obszarze dyscyplinują notariuszy. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości rekomendujemy przyjęcie sprawozdania. Panu ministrowi chciałbym bardzo podziękować za przedstawienie dokumentu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Kazimierz Plocke, Klub Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Rok 2019 był trzecim pełnym rokiem, w którym cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu oraz Konfederacji Szwajcarskiej, mogli nabywać nieruchomości rolne i leśne na takich samych zasadach jak obywatele Polski, tj. od 1 maja 2016 r. Nabywcy z innych państw nadal muszą uzyskiwać stosowne zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na podstawie sprawozdania MSWiA dotyczącego nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w 2019 r. odnotowano 8690 transakcji nabywania nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców o ogólnej powierzchni 5238 ha.

Z powierzchni nabytych przez cudzoziemców w 2019 r. 1349 ha stanowiły grunty rolne i leśne, w tym 377 ha to grunty leśne, które zostały zakupione w przypadku 1279 transakcji.

Dla porównania w 2018 r. były to 1044 transakcje dotyczące powierzchni 799 ha, w tym 182 ha to grunty leśne.

Panie ministrze, prosiłbym o komentarz, jakie były powody tak istotnego wzrostu i jak nabywcy motywowali swoje wnioski. Cudzoziemcy nabywali także udziały i akcje w spółkach prawa handlowego będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych. W 2019 r. zarejestrowano 670 takich transakcji, które dotyczyły 5879 ha.

Jeżeli chodzi o grunty rolne i leśne, to największa powierzchnia tych gruntów dotyczyła województwa zachodniopomorskiego - 949 ha, pomorskiego - 747 ha i opolskiego - 651 ha. Z analizy sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji za 2019 r. wynika, że wydano 19 decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali oraz akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Cudzoziemców z których państw one dotyczą? Z informacji, którą przedstawił minister spraw wewnętrznych, wynika również, że w 2019 r. przeprowadzono 84 transakcje z naruszeniem prawa.

Wysoki Sejmie! Po analizie przedstawionego Wysokiej Izbie sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dzwonek) w roku 2019 Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska będzie głosować za przyjęciem tego sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2019 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a wiec ustawy ze 100-letnią historią. Przedmiotowy druk nr 292 był rozpatrywany podczas prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 30 września br.

W 2019 r. minister właściwy do spraw wewnętrznych wydał łącznie 19 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali oraz akcji i udziałów.

Cudzoziemcami najczęściej występującymi do ministra o uzyskanie zezwolenia na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych, biorąc pod uwagę liczbę zezwoleń, byli obywatele Ukrainy - 105 lokali, Białorusi - 27 i Rosji - 10 lokali. Niepokojąca jest zapewne liczba aktów przesłanych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych z uchybieniem ustawowego terminu przez notariuszy, bowiem w roku 2019 było ich aż 158, o czym mówił mój przedmówca. W 2019 r. odnotowano również niestety 84 transakcje zawarte z naruszeniem przepisów ustawy. W ramach prac komisji w trakcie odpowiedzi udzielanych przez przedstawicieli Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych potwierdzono, że w ministerstwie do tej pory nie była badana efektywność obywatelstw w ramach procesu nabywania nieruchomości. Całe sprawozdanie jest obszerne - zawiera podstawy prawne i wyjaśnienia dotyczące obowiązujących w tym zakresie regulacji, co zapewne ułatwiło prezentację przedmiotowego sprawozdania za rok 2019. W kolejnych sprawozdaniach dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców wnioski i analizy mogłyby być bardziej szczegółowe. Należy również zwiększyć nadzór nad realizacją niniejszej ustawy. Chciałbym podziękować w imieniu komisji administracji za przesłany nam dodatkowy materiał.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Lewicy będzie głosował za przyjęciem niniejszego sprawozdania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz głos zabierze pani poseł Urszula Nowogórska, Koalicja Polska - PSL. Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicji Polskiej - PSL - Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści przedstawić stanowisko wobec sprawozdania MSWiA z realizacji w 2019 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców zawartej w druku sejmowym nr 292 oraz stanowiska komisji zawartego w druku nr 639. Wysoka Izbo! Reglamentacja obrotu nieruchomościami w Polsce z udziałem cudzoziemców polega na obowiązku uzyskania przez cudzoziemca stosownego zezwolenia, które jest podstawą do nabywania nieruchomości na zasadach obowiązujących polskich obywateli. Kluczowe zatem jest rozstrzygnięcie, kto jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy. Definicja jest bardzo szeroka, gdyż przyznaje status cudzoziemca po pierwsze osobie fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej mającej siedzibę za granicą, nieposiadającej osobowości prawnej spółce osób, o której wspomniałam powyżej, mającej siedzibę za granicą, utworzonej zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. Kolejny przypadek to są osoby prawne i spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione powyżej. Po analizie przedstawionego dokumentu okazało się, że w 2019 r. wpłynęło do ministerstwa, MSWiA, 767 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce, a także o wydanie przyrzeczeń, tzw. promes. W stosunku do 2018 r. odnotowano 19-procentowy wzrost liczby wniosków.

434 były to osoby fizyczne, dwa - osoby prawne, trzy - przedstawicielstwa dyplomatyczne. W 2019 r. wykonano, przepraszam, wydano 140 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych. Wydano 20 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości o powierzchni 136 ha. Powodem odmów był brak uzasadnienia trwałego związku z Polską.

Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska obecnie, a w wcześniej samo Polskie Stronnictwo Ludowe, w 1997 r. doprowadziło do tego, że powstał art. 23 konstytucji, który mówił, co jest istotą ustroju rolnego, i wskazywał na gospodarstwo domowe. Należy również przypomnieć, że w zasadzie minęło 100 lat od chwili uchwalenia ustawy z dnia 24 marca 1920 r. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana i była również powodem tego, co w praktyce sprawiało kontrowersje i problemy interpretacyjne. Pozwoliłam sobie również na analizę wcześniejszych raportów.

W związku z powyższym i w związku z tendencją wzrostową sprzedaży gruntów Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści będzie się bacznie przyglądać prowadzonej polityce sprzedaży, ale również będzie prosiła o zwiększenie nadzoru nad tymi działaniami.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w 2019 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zacznijmy historycznie. Ta ustawa jest rzeczywiście stara, ma ponad 100 lat, została uchwalona w 1920 r., jest z czasów świeżo odzyskanej niepodległości. Wspomnijmy, rewolucja na wschodzie zdążyła już zebrać swoje pierwsze krwawe żniwo, nawała bolszewicka rusza na zachód, Polska wówczas dzięki własnej waleczności i dzięki Bogu nie dała się zdeptać wschodniemu butowi. W takich właśnie okolicznościach powstaje ta ustawa. Co ciekawe, powstała zanim jeszcze ujednolicono obowiązujące po zaborach prawo w szeregu innych bardzo ważnych dziedzin. Jest ona wyrazem ważnej myśli, takiej, że niepodległy naród polski powinien niepodzielnie rządzić się w granicach swojego terytorium i nad tym terytorium całkowicie panować. Chciałem przypomnieć również myśl, korzystając z tej okazji, jaką wyraził w 2002 r. narodowy poseł z tego miejsca, z mównicy sejmowej. Szukając narodowego interesu gospodarczego w obrocie ziemią, przypominał różnicę między dzierżawą i sprzedażą. Przywoływał w tym kontekście przykład sprzedanej przez Rosjan Ameryce Alaski i wydzierżawionego Brytyjczykom przez Chińczyków Hongkongu, który do nich po 100 latach wrócił. Te tezy padały w kontekście ziemi, której, jak wiadomo powszechnie, nie przybywa. Zasób jest stały, państwo powinno tego zasobu strzec. Biorąc pod uwagę m.in. unijne zasady swobodnego przepływu kapitału osób, możliwości osiedlania się, również napływ imigrantów ze Wschodu i Azji, słusznie państwo polskie monitoruje corocznie transakcje, jakie zachodzą w przestrzeni obrotu nieruchomościami. Powinno czynić to nadal i nie dopuścić do masowej migracji, zwłaszcza ze Wschodu, z Azji, Afryki, realnie weryfikując kto się w Polsce osiedla, nabywa nieruchomości. Działania te konieczne są po to, aby polska wspólnota mogła żyć i rozwijać się bezpiecznie, jak również po to, aby skończyć z drenażem polskiego kapitału, ludzkiego na Zachód, by państwo polskie było najatrakcyjniejszą ofertą dla młodych Polaków do życia i rozwoju. Zważywszy na dość niski poziom odmów wskazany w raporcie, jawi się pytanie: Czy dostatecznie dobrze sprawdzane są związki nabywców z Polską? Z tym zagadnieniem wiąże się również problematyka wykupowania ziemi przez tzw. słupy, a także przez spółki, których struktura własnościowa jest na tyle skomplikowana, że na pierwszy rzut oka nie można rozróżnić, kto faktycznie pociąga za sznurki. I tu pojawia się fundamentalne pytanie: Czy polskie służby właściwe w tym zakresie ten problem identyfikują i go należycie monitorują? Szczególnie dotyczy to obszarów o strategicznym znaczeniu: obiektów wojskowych, lotnisk, elektrowni, sieci przesyłowych, ujęć wody pitnej czy obszarów geograficznych istotnych, jak obszary przygraniczne czy Mierzeja Wiślana. Pytanie do pana ministra: Czy ta kontrola jest skrupulatnie sprawowana? Teraz głos ma pan poseł Dobromir Sośnierz, również koło Konfederacji. To przykład czegoś, czego kompletnie nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy tej ustawy, nie potrzebujemy tych raportów, nie potrzebujemy tego gadania o niczym, z którego kompletnie nic dla nikogo nie wynika. Państwo w ministerstwie wykonuje kawał ciężkiej i nikomu niepotrzebnej pracy weryfikowania tego, co kto od kogo kupuje. Jeśli właściciel chce coś komuś sprzedać i traktuje ją poważnie, sprawę własności, to jest to sprawa między nim a sprzedającym. Jeśli działka jest moja, to jest moja, a to oznacza, że minister nie ma prawa decydować o tym, a jeśli ma prawo, tzn. że już nie jest do końca moja, bo jest jakby jeszcze trochę ministra. W związku z tym nie widzę żadnego powodu, żebyśmy pochylali się nad tak nieistotną kwestią, żebyśmy kontrolowali własnych obywateli w tym, co komu chcą sprzedać, żebyśmy wydawali pieniądze na zupełnie niepotrzebne etaty dla osób, które ślęczą nad tymi dokumentami, i żebyśmy po prostu przeszkadzali w obrocie działkami własnym obywatelom. Wkładamy po raz kolejny kij w szprychy własnej gospodarki, a potem dziwimy się, że to wszystko kuleje. Dziękuję. Teraz głos zabierze podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Bartosz Grodecki.

A więc zamykam listę zgłoszonych do pytań. Wyznaczam czas pytania na 1 minutę. Pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czy rząd planuje w związku z tym uwolnić handel ziemią, tak żeby Polacy mogli bez problemu, bez ograniczeń z jednej strony sprzedawać, a z drugiej strony nabywać ziemię i choćby budować swoje nieruchomości, zwiększać rozwój i prowadzić normalne, nieskrępowane życie? Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 3 sierpnia 2019 r. na spotkaniu we wsi Dygowo lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział następujące słowa w kontekście ustawy o ochronie ziemi: zabezpieczyliśmy polską ziemię, polska ziemia musi być dla polskich rolników. Mam prośbę: Czy pan minister mógłby przekazać swojemu liderowi oficjalne dane MSWiA, które mówią, że w 2015 r., czyli kiedy PO i PSL oddawały władzę, obcokrajowcom sprzedano 412 ha ziemi, natomiast w latach następnych, kiedy wy rządziliście, tej ziemi obcokrajowcom sprzedawane było coraz więcej? Czy te dane nie mówią jasno, że beneficjentami polityki rolnej PiS są rolnicy niemieccy, a nie polscy? No i trzeba powiedzieć także jasno, że PiS nie stworzył żadnej ustawy o ochronie polskiej ziemi, PiS 3-krotnie umożliwił sprzedaż jej obcokrajowcom. Dziękuję bardzo. Mam pytanie: Czy rząd Zjednoczonej Prawicy, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma jakiś plan, jeśli chodzi o ilość ziemi, która w ręce cudzoziemców będzie trafiała w kolejnych latach? Mój kolega poseł Dariusz Klimczak przypomniał, jakie były zapowiedzi. Miało zero powierzchni, polskiej ziemi trafiać do obcokrajowców, a tymczasem dane przeczą temu całkowicie. A więc dzisiaj warto sobie zadać pytanie: Jaki jest, panie ministrze, plan na przyszłość? Oglądają nas dzisiaj rolnicy, którzy bardzo dobrze pamiętają te słowa i prezesa Kaczyńskiego, i innych czołowych, prominentnych polityków PiS-u, że ziemia przestanie trafiać w ręce cudzoziemców. Tak jak z dopłatami unijnymi, z wieloma innymi rzeczami, oszukaliście polskich rolników.

Panie Ministrze!

Moje pytanie brzmi: Jak wygląda obrót nieruchomościami w kontekście narodowości w województwie lubelskim, jeśli chodzi o zarówno nieruchomości, jak i nieruchomości rolne, udziały w spółkach, udziały, a także lokale? Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! O tym, że tę ziemię sprzedaje się obcokrajowcom za państwa rządów, już wiemy, statystyki o tym mówią.

Panie ministrze, oni są właścicielami albo współwłaścicielami poprzez spółki. Czy ministerstwo ma informacje, ile na dzień dzisiejszy ziemi na Pomorzu Zachodnim jest z udziałem kapitału zagranicznego i w jaki sposób zamierzacie tę ziemię oddać polskim rolnikom?

Dziękuję, panie marszałku. Panie Ministrze! Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie. 30 kwietnia 2021 r. kończy się 5-letni okres, jeżeli chodzi o zakaz sprzedaży ziemi rolnej innym podmiotom niż rolnicy.

Ile spółek prawa handlowego z większościowym i mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego nabyło ziemię rolną i leśną w roku 2019, jakie to są powierzchnie i z jakich państw te podmioty pochodzą?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa, nad którą dzisiaj procedujemy, daje szanse, żebyśmy porozmawiali o tym, jak wygląda współpraca, koordynacja służb w zakresie cudzoziemców.

Te elementy są ważne z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego. Odpowiedź na to pytanie może też otworzyć nam oczy na to, jak rzeczywiście wygląda dzisiaj próba nielegalnego przekraczania granicy. Prosiłbym pana ministra o rzetelną i prawdziwą odpowiedź, tak żeby w przyszłości, w 2021 r., można było w tej sprawie odbyć realną debatę. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wielokrotnie nowelizowana przetrwała cały wiek pomimo istotnych zmian politycznych, a w praktyce powoduje dziś kontrowersje i problemy interpretacyjne nawet u doświadczonych prawników. Przyjęta obecnie interpretacja przepisów ustawy powoduje, że w profesjonalnym obrocie ograniczenia w nabywaniu nieruchomości wynikające z tej ustawy są nieistotne, a praktyczna doniosłość tej ustawy jest niewielka, gdyż bardziej niż reglamentacją obrotu nieruchomościami zajmuje się ona obrotem udziałami i akcjami, co oznacza, że już sam tytuł jest mylący. A cudzoziemiec spoza europejskiego obszaru gospodarczego, chcąc nabyć nieruchomość w Polsce, po prostu najpierw zakłada spółkę, a potem już samo nabycie nieruchomości przez tę spółkę nie wymaga zezwolenia. Nasuwa się zatem pytanie, czy ta ustawa nadal spełnia swój pierwotny cel i czy nie należałoby jej uchylić, zastępując ją nową regulacją, która w sposób niebudzący sporów interpretacyjnych regulowałaby przedmiotową materię.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 13 listopada 2016 r. prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział: Polska ziemia nie dla spekulantów, polska ziemia nie dla obcych, polska ziemia dla polskich rolników. Dzisiaj widzimy, ile ziemi zostało sprzedane. Może to nie byłoby tak bulwersujące, gdyby nie fakt, że rolnicy w Polsce faktycznie mają problem. Jest odbierana ziemia, którą dzierżawią wiele lat i o którą dbają jak o własną, jest wstrzymywany ruch tą ziemią, bo nie są to właściwi dzierżawcy, muszą przyjść nowi, związani koniecznie ze środowiskiem PiS-u. Niestety taka jest rzeczywistość. A nie zadbaliście o to, by cudzoziemcy nie kupowali tej ziemi, bo dla was najważniejsze są pieniądze, które z tego procederu pozyskujecie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze.

Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni Panowie Posłowie! Szczerze powiedziawszy, trochę nie za bardzo rozumiem te głosy oburzenia ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Wzrost sprzedaży gruntów rolnych obywatelom państw pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wynika z tego, że w 2016 r. przestały po prostu obowiązywać okresy przejściowe, a te okresy przejściowe były wynegocjowane na 12 lat w 2004 r. Kto te okresy negocjował? Chyba państwo jako ci, którzy tworzyli wówczas rząd. Myślę więc, że pytanie nie jest właściwie skierowane do nas, tylko chyba powinniście sobie państwo na nie sami odpowiedzieć.

Jest nim ministerstwo rolnictwa, a nie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czytam swoje wystąpienie dotyczące właśnie tego sprawozdania - sprawozdanie dotyczy prowadzenia rejestrów sprzedaży tych gruntów, czyli tych czynności, które zostały wprowadzone do polskiego obrotu prawnego, zostały zarejestrowane przez notariuszy, przez sądy i zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie bardzo się poczuwam do tego, żeby odnosić się do tego, jak funkcjonuje ustawa o obrocie rolnym, bo nie jesteśmy jej depozytariuszem.

Wynika to z wielu różnych spraw. Sąd może zawsze uchylić taką decyzję i przekazać ją do ponownego zbadania, a odmowy, które wydajemy w procesie prowadzenia swoich postępowań, wynikają głównie z niespełnienia przez wnioskującego przesłanek ustawowych, takich jak chociażby niewykazanie, skąd ma środki na nabycie danej nieruchomości. Odnosząc się jeszcze na sam koniec, jeśli można, do tego, co przedstawił pan poseł Sośnierz, rozumiem, że jest rzeczywiście tak, że jest właściciel gruntu, który ma wolną możliwość sprzedaży swojego gruntu, komu chce, jeżeli nie dotyczy to osoby spoza EOG. Jako urząd jesteśmy zobowiązani do jej przestrzegania i kontynuowania tego procesu wynikającego z zapisów ustawy. To też jest jakby odpowiedź po części na postulaty zgłoszone przez panów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To znaczy, że jeżeli ktoś jest właścicielem gruntu i chce ten grunt sprzedać, to słusznie: co państwu do tego, skoro okresy przejściowe już się zakończyły. Chce sprzedać, to je sprzeda. Natomiast tak jak powiedziałem podczas tego wystąpienia, część pytań rzeczywiście powinna trafić do ministerstwa rolnictwa, które jest właściwe, jeśli chodzi o ustawę o obrotach gruntami rolnymi. Bardzo dziękuję. Czy pan sprawozdawca komisji chce zabrać głos? Pan Paweł? Bardzo proszę, w trybie sprostowania. Pół minuty. Ale mówiłem, że właśnie jest to kompletnie zbędna inicjatywa i szkoda pańskiego cennego czasu, żeby pan pochylał się z wysokości swojego stolca nad takimi drobiazgami, jak to ktoś komuś sprzedaje działkę. Wobec zgłoszonego sprzeciwu do głosowania. Wobec sprzeciwu do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 15 grudnia br. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Jako pierwszy pan poseł Fryderyk Kapinos, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Był synem Eugeniusza i Zofii z Sockich. Okres jego młodości przypadł na czasy II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej.

Od sierpnia 1940 r. do stycznia 1945 r. był harcerzem Szarych Szeregów Armii Krajowej w drużynie im. Jeremiego Wiśniowieckiego, natomiast od stycznia 1945 r. do listopada 1951 r. - w tajnej niepodległościowej drużynie harcerskiej im. Jeremiego Wiśniowieckiego, która występowała też pod nazwą Wolność i Sprawiedliwość.

W listopadzie 1951 r. został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia za działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych. Rok później ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej z tytułem inżyniera. Następnie od czerwca 1957 r. do grudnia 1982 r. pracował w WSK i OBR SK Mielec w służbach konstrukcyjno-badawczych m.in. jako (Dzwonek) kierownik sekcji konstruktorskiej nadwozia samochodu Mikrus. Zmiana sytuacji politycznej w Polsce po roku 1989 r. umożliwiła Jerzemu Dębickiemu reaktywowanie rodzinnej biblioteki, zabranej przez komunistyczne władze jego ojcu Eugeniuszowi Dębickiemu. Został awansowany na stopień kapitana Wojska Polskiego oraz odznaczony m.in. Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pełnił funkcję prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu. Kpt. Jerzy Dębicki bardzo angażował się w działalność o charakterze patriotycznym. Chętnie uczestniczył w spotkaniach z młodzieżą, dla której był przykładem i wzorem do naśladowania. Bardzo dziękuję. Pan poseł Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska.

Bardzo dobrze, co z tego. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 12 grudnia 1860 r., 160 lat temu, w Szymborzu koło Inowrocławia urodził się wielki poeta, dramaturg, krytyk literacki, tłumacz, również rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie - Jan Kasprowicz. Był wybitnym przedstawicielem Młodej Polski, związany z naturalizmem, symbolizmem oraz ekspresjonizmem. Uważany za jednego z najwybitniejszych poetów w dziejach literatury polskiej, stawiany na równi z Adamem Mickiewiczem. Ważne miejsce w jego poezji zajmował zachwyt nad przyrodą rodzimych Kujaw, szczególnie inowrocławskich, oraz Tatr, gdzie spędził koniec swojego życia. Dom Jana Kasprowicza w Szymborzu czy właściwie budynek odbudowany na miejscu dawnej chaty, w której urodził się Jan Kasprowicz, jest to muzeum. Niestety to muzeum jest w tej chwili zapomniane, niedofinansowane. Moje wystąpienie jest apelem, aby przypomnieć o tym wielkim poecie, o tym wielkim artyście, również ministerstwu kultury i społeczeństwo, abyśmy też wspólnie może w tej Izbie w przyszłości zastanowili się, jak godnie uhonorować, ale także dofinansować to miejsce, aby przypomnieć o tym, że Jan Kasprowicz był związany przede wszystkim z Kujawami z racji swojego urodzenia, był tak naprawdę też obywatelem świata, bo studiował w Lipsku, znał doskonale język niemiecki, również języki wschodnie oraz był też związany bardzo mocno z Lwowem. To nie tylko „Harenda” w Zakopanem, gdzie jest jego muzeum, ale to również właśnie muzeum w Szymborzu, rodzinnym Szymborzu koło Inowrocławia. I mój apel z tym związany, aby w przyszłości ministerstwo kultury zastanowiło się nad tym, aby dofinansować remont, ale także bardziej upublicznić to miejsce i wspomóc finansowo powiat inowrocławski, który prowadzi jednostkę kultury i gospodaruje tamtym miejscem, aby godnie upamiętnić miejsce narodzin tego wielkiego artysty. Dziękuję.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy okazji nie mogę sobie nie pozwolić na refleksję, że jak na punkt: oświadczenia, to spotykamy się o dość niezwykłej porze, nawet nienaturalnej, bo zazwyczaj są to późne godziny nocne. Dziś Izba przyjęła uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy Grudnia ’70. Jako gdańszczanin chciałbym za nią bardzo podziękować. Projekt uchwały przedstawiło Prezydium Sejmu, zaś za kanwę posłużył projekt zgłoszony przez klub Koalicji Obywatelskiej. Prezydialny projekt uchwały narodził się - co jak najbardziej naturalne w demokracji - na drodze konsensusu. Z tego też powodu nie znalazł się w nim pewien odnoszący się do teraźniejszości, jak i do przyszłości fragment, pewien rodzaj przesłania. Dlatego też chciałbym pozwolić sobie go przytoczyć: Odwołując się do doświadczenia Grudnia ’70, Sejm Rzeczypospolitej wskazuje, że nie siła i przemoc, a dialog oraz kompromis winny służyć rozwiązywaniu konfliktów między społeczeństwem i władzą. Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje oświadczenie poselskie dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców i budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 30 w kierunku Zgorzelca w miejscowości Chmieleń. Chmieleń to kilkukilometrowa miejscowość, przez którą przebiega stosunkowo wąska droga krajowa nr 30 w kierunku Zgorzelca. W szybkim tempie rośnie ruch samochodowy na tej drodze, w tym ciężkiego transportu w kierunku Niemiec. Bezpieczeństwo mieszkańców jest zagrożone i konieczna jest szybka budowa chodnika, a docelowo obwodnicy. Niestety od lat nic się nie dzieje. Mało tego - w odpowiedzi na moją interpelację minister infrastruktury nie jest w stanie określić przybliżonego terminu budowy. Mieszkańcy proszą o chodnik, składają apele i wnioski, a ostatnio protestują na ulicy. Czy naszego państwa, które, jak słyszymy od rządu, ma finanse publiczne w doskonałym stanie, nie stać na 300 tys. zł rocznie przez 2 lata, aby wybudować ludziom chodnik, żeby czuli się bezpiecznie w drodze do szkoły, sklepu, przychodni zdrowia czy na przystanek? Czy nie jest to podstawowa potrzeba? Jak można tak ignorować mieszkańców i lekceważyć ich bezpieczeństwo? Jako poseł tej ziemi piszę kolejne zapytania i interpelacje do ministra infrastruktury. Odpowiedź identyczna od kilku lat: że priorytety, autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, że kolejność realizacji zgłoszonych zadań inwestycyjnych określa się według kryteriów: liczba zabitych, liczba rannych, średni dobowy ruch na danym odcinku drogi.

Czytając to, mam wrażenie, że chodzi o wielomilionową inwestycję, a nie chodnik za 700 tys. zł.

Pan poseł Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy oburzeni. Tak, mówię w liczbie mnogiej - w imieniu samorządowców, a w szczególności w imieniu mieszkańców Opola. Jesteśmy oburzeni tym, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość rozdzieliło miliony z funduszu inwestycji lokalnych, zarówno w wymiarze krajowym, jak i w szczególności w wymiarze lokalnym. Nic nie znaczą. Obiecaliście pomóc samorządom w trudnym czasie pandemii, tymczasem ta pomoc trafia tylko do wybranych samorządów, zapewne nieprzypadkowo tylko do tych, które wspierają PiS. Dokładnie tak to wygląda w Opolu, którego jestem reprezentantem. Pieniądze z funduszu daliście tylko swoim, ale podatki bierzecie od każdego. Wstyd, zarówno politycznie, jak i tak po ludzku. Zostaliśmy kompletnie pominięci pomimo złożenia ważnych społecznie wniosków dotyczących przedszkola, sali gimnastycznej czy domu pomocy społecznej, niezbędnego do normalnego funkcjonowania polityki senioralnej. Tyle okrągłych słów, że troszczycie się o najmłodszych, a seniorom poprawiacie życie. To puste frazesy i niespełnione obietnice. Tyle w praktyce warte są wasze słowa. Wysoka Izbo! Jako rządzący Zjednoczona Prawica zapewniała, że praktyki dzielenia Polski na Polskę A i Polskę B, na lepszą i gorszą, na bogatszą i biedniejszą to już melodia przeszłości. A co zrobiliście? Jeszcze bardziej dzielicie kraj, tylko teraz linia podziału biegnie inaczej. Jest Polska wasza i Polska nie wasza, Polska PiS, która wam przytakuje, oraz cała reszta, która ma odwagą myśleć i mówić inaczej. Gdzie tu prawo, gdzie tu sprawiedliwość? Nie ma ani prawa, ani tym bardziej sprawiedliwości. Tak, jesteśmy oburzeni. Przypominam, że mówię to w imieniu mieszkańców Opola.

Zapowiadaliście transparentność, przejrzystość. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Wysoka Izbo! To, co zrobił rząd Zjednoczonej Prawicy, jest karygodne także dlatego, że krzywdzicie również swoich wyborców. Myślicie, że seniorzy z Opola nie głosowani w ostatnich wyborach na Andrzeja Dudę? Myślicie, że wcześniej nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych? Pomijacie istotną część swoich wyborców. Wielu na was głosowało, ale po tym, co zrobiliście, już tego nie powtórzą. Bądźcie pewni, że ludzie nie zapominają.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

W 1920 r. wraz rodzicami wrócił do Polski.

Odtąd posługiwał się pseudonimem Jelonek. Po wojnie ukończył Wydział Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie. Pracował z dziećmi, stworzył orkiestrę szkolną. Prowadził 120-osobowy chór w Zielonej Górze. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, dwukrotnie Medalem Wojska oraz wieloma innymi medalami, w tym odznaczeniem „Przyjaciel Dziecka” za pracę z dziećmi i młodzieżą. Do końca życia był aktywnym członkiem Związku Inwalidów Wojennych. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Cześć jego pamięci. Chciałam jeszcze, korzystając z wolnego czasu, złożyć drugie oświadczenie.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Monika Falej, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś rano zadzwoniła do mnie zapłakana kobieta z Iławy, która dowiedziała się, że być może jest w ciąży, w wyniku której urodzi martwy płód. To wielka tragedia dla niej i najbliższych. Dlaczego zadzwoniła do mnie? Bo ta przerażająca, trudna sytuacja ma drugie, polityczne dno, które sprawia, że ta kobieta przeżywa podwójne piekło. Chciała porady ginekologa, ale ten odmówił przyjęcia jej na oddział. Przyznał, że od 22 października on i jego szpital omijają temat szerokim łukiem, że dla własnego bezpieczeństwa zasłaniają się klauzulą sumienia, ale może ją przyjąć prywatnie. Tak jest w Iławie. Podobna sytuacja miała miejsce w szpitalu miejskim w Olsztynie. Tzw. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji uchylający możliwość przerywania ciąży z powodu ciężkich i nieuleczalnych wad płodu został wydany 22 października 2020 r. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powinny być publikowane w Dzienniku Ustaw niezwłocznie, ale rząd nie zrobił tego do dziś. Wiele osób mówi, że dzięki temu orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma mocy prawnej. Pewnie tak jest, ale Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nie publikując orzeczenia, nie próbuje złagodzić chaosu i frustracji milionów Polek i Polaków, chowa głowę w piasek i czeka na rozwój wydarzeń. Kancelaria premiera otwarcie przyznaje, że nie publikuje orzeczenia, ponieważ czeka, aż Sejm posprząta ten bałagan i przyjmie nową ustawę aborcyjną, najlepiej zaproponowaną przez prezydenta. Gdy szukam dla tej kobiety miejsca, gdzie spokojnie może się zgłosić i w pełni praw skorzystać z opieki medycznej, w Internecie widzę: „Szpital Bielański wstrzymuje zabieg aborcji”, „Zabiegi aborcji na Polnej wstrzymane”, „Aborcja w Elblągu nadal legalna” Kolejny tytuł: „W szpitalu w Iławie wszyscy lekarze zgłosili klauzulę sumienia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązuje, skutki już są” Szanowna Pani Przyłębska! Panie Kaczyński! Proszę oddzwonić do tej kobiety, która dziś błaga mnie o pomoc, i powiedzieć jej, że załatwiacie swoje problemy, żeby poczekała, aż państwo się dogadacie. Dziwne, że jeszcze państwo tej kwestii nie poruszyliście przy kawie, bo tyle państwa dramat Polki porusza, że pewnie jest on wart drobnego wątku podczas pogaduch pana Kaczyńskiego i jego towarzyskiego odkrycia ostatnich lat. Dziękuję.

Panie Przewodniczący Komitetu Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ nie mogłam zadać pytania odnośnie do raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrobię to teraz. Rocznie w Polsce dochodzi do ok. 500 zabójstw. To straszne, prawda? Otóż nie, prawdziwym zagrożeniem są kierowcy. Co roku z ich rąk ginie 3 tys. osób, a 35 tys. zostaje rannych. To wszystko są śmierci, kalectwa i nieszczęścia, których w większości można byłoby uniknąć. Panie Ministrze Ziobro! Tu jest miejsce na program: zero tolerancji. Bądźcie bezwzględni nie dla bezbronnych, ale dla tych, którzy przekraczają prędkość, wyprzedzają na podwójnej ciągłej, bo to oni są potencjalnymi mordercami. Kiedy skończymy z przyzwoleniem na łamanie zasad ruchu drogowego, z leczeniem kompleksów poprzez kupowanie drogich i szybkich samochodów, z tym największym chamstwem na drogach Europy? Fotoradary w każdej gminie, wysokość mandatów powiązana z zarobkami i koniec pobłażliwości sądów dla piratów drogowych. Oto moje postulaty.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Już 75 lat minęło od zakończenia II wojny światowej. Niestety do dzisiaj nie przeprowadzono dokładnej inwentaryzacji i badań polskiego dna morskiego. Według szacunków Najwyższej Izby Kontroli na dnie Bałtyku w polskiej strefie odpowiedzialności spoczywa ok. 400 wraków, zaś w samej Zatoce Gdańskiej jest ich ok. 100. Dzisiaj mogliśmy usłyszeć jak rząd Polski dba i chroni brzegi morskie. Najwyższy czas, aby zacząć dbać o dno naszego morza, wszak Bałtyk jest jednym z najmniejszych i najbardziej wrażliwych na zmiany ekologiczne akwenów na świecie. Z tego też względu wspólnie z samorządowcami Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań w celu jak najszybszego wdrożenia programu, który dokona szczegółowej inwentaryzacji zatopienia broni chemicznej i bojowych środków trujących, chociażby takich jak iperyt czy sarin. Apeluję także o opracowanie sposobu wydobycia i neutralizacji broni chemicznej. Wreszcie należy wybudować i wyposażyć wielozadaniowy statek zdolny do wydobywania broni chemicznej i produktów ropopochodnych oraz zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Pani poseł Monika Wielichowska, klub Koalicji Obywatelskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś rozwój wsi i miast, powiatów zależy od centrali w Warszawie i od tego, czy wójt, burmistrz czy starosta popiera PiS, czy nie popiera, czy podpisuje porozumienie Duda 2020, czy też nie podpisuje. Tak zabija się samorządy, samorządność, tak zabija się lokalne wspólnoty, tak tworzy się kolejne niepotrzebne podziały. Premier, informując o funduszu inicjatyw lokalnych, zapowiedział, że nie będzie dzielenia Polski na A, B i C. Mówił też: Przeznaczamy dodatkowe środki dla małych ojczyzn - 12 mld zł. Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą motorem napędowym rozwoju gmin i powiatów, podnosząc jakość życia Polaków. Myślimy o zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju. Ale na pustych słowach się skończyło, bo podzielił Polskę na lepszy i gorszy sort. Sprawdźmy jak wygląda według władzy tzw. sprawiedliwy i zrównoważony podział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w okręgu wałbrzyskim. Ani jedna złotówka nie trafiła do wielu miast, gmin, powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, świdnickiego czy też wałbrzyskiego. Miasto Kłodzko dostało zero, miasto Nowa Ruda - zero, Lądek-Zdrój - zero, Kudowa-Zdrój - zero, Lewin Kłodzki - zero, Szczytna - zero, Polanica-Zdrój - zero, Stronie Śląskie - zero, powiat kłodzki, ten samorząd złożył dziewięć ważnych dla mieszkańców powiatów wniosków, zero, Wałbrzych - zero, Jedlina-Zdrój - zero, Głuszyca - zero, Stare Bogaczowice - zero, Świdnica miasto - zero, Świdnica gmina - zero, Dobromierz - zero, Świebodzice - zero, Żarów - zero, Dzierżoniów miasto - zero, Bielawa - zero, Pieszyce - zero, Ząbkowice Śląskie - zero, Stoszowice - zero. To są miasta, gminy i powiaty, w których mieszkańcy ciężko pracują i płacą podatki. Mimo to władza ich wykluczyła, mimo to władza ich zlekceważyła.

Wygrała uznaniowość i partyjny klucz, przegrała sprawiedliwość i uczciwość, przegrała przyzwoitość. Tej skandalicznej sprawy nie zostawimy. Będziemy domagać się od premiera informacji dotyczących kryteriów, zasad, na podstawie których jednostkom samorządu terytorialnego przyznaje się lub przyznano środki z tegoż funduszu. Chcemy poznać protokoły ocen wniosków, które zostały złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, sformułowanych w ramach działalności Komisji do Spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego. Chcemy poznać listę członków komisji, którą prezes Rady Ministrów powołał w celu udzielenia wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego. Sprawę rozdysponowania funduszu zgłosiliśmy także do Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ rozdysponowanie tego funduszu jest absolutnie skandaliczne. Pan poseł Wojciech Król, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym powiadomić Wysoki Sejm o podejrzeniu zaistnienia korupcji, korupcji politycznej, bo sposób, w jaki rząd rozdzielił środki publiczne w ramach funduszu inwestycji samorządowych zmusza właśnie do takiej refleksji. Ze wstępnej analizy wynika, że aż 70% samorządów, które otrzymały środki finansowe, stanowią samorządy związane z Prawem i Sprawiedliwością. Polska coraz bardziej przypomina PRL. Rządzi nami jakiś jegomość, a cała reszta to jest atrapa. Kto nie z nami, ten przeciwko nam. Te ławy również są puste. Sejm jest niemy. Ale to nie jest najgorsze, że te ławy są puste, najsmutniejsze jest to, że to nie ma żadnego znaczenia, czy te ławy są puste, czy są pełne. Muszę zapytać, czy prawdą jest, że są przypadki handlowania publicznymi pieniędzmi. Pieniądze dla samorządu w zamian za stanowisko dla politycznego nominata z Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę dla konia trojańskiego z logo Prawa i Sprawiedliwości, bo w taki sposób chcecie przejmować samorządy - pieniądze za stanowiska. Jeżeli te informacje się potwierdzą, że rząd kupczy publicznymi pieniędzmi, to będzie to kolejny dowód na to, że dla tej władzy nie istnieją żadne granice. To byłaby korupcja, to byłby szantaż, to byłoby przestępstwo, a tak naprawdę byłby to moralny upadek państwa. Kolejny przykład: koperta z nazwiskiem córki leśniczego. Jestem ze Śląska i my na Śląsku pamiętamy, jak PiS umoczył Kałużę, jak przejął władzę w województwie śląskim. Nie wygraliście wyborów w Sejmiku Województwa Śląskiego, bo nie potraficie rządzić samorządami, więc kupiliście sobie władzę. Kupiliście władzę za publiczne pieniądze, kupiliście sobie władzę za pieniądze mieszkanek i mieszkańców województwa śląskiego. Kupczycie, kupczycie Polską jak na zwykłym targowisku, ale to kiedyś się skończy, bo każda władza kiedyś się kończy. Wysoka Izbo!

Wiecie państwo, kogo zabrakło? Zabrakło strony rządowej, rządu, ministerstwa rolnictwa, które nie interesuje się sytuacją w rolnictwie. Panie Ministrze!

Nie ma go. Gdybyśmy mieli holding, może by do tych sytuacji nie dochodziło. Gdybyśmy mieli ceny minimalne, może by do tego nie dochodziło. Co dzisiaj z tego zostało, szanowni państwo? Napuszczanie rolników na koła łowieckie, a Skarb Państwa, który jest właścicielem zwierzyny, umywa ręce. Po nowym roku będziemy mieli masowe likwidacje kół łowieckich, bo nie ma polowań dewizowych, nie ma pieniędzy. Dlatego apeluję bardzo mocno do pana ministra, do pana premiera, żebyśmy wreszcie zajęli się sytuacją w rolnictwie, bo rolnictwo samo sobie nie poradzi.

Ludzie zainwestowali ogromne miliony, budowali swoje gospodarstwa latami, a dzisiaj nie mają wyjścia. I jeszcze na koniec: Polska - kiedyś jeden z liderów, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków Unii Europejskiej. Czyli na którym? Na ostatnim. Bo kończy się perspektywa, wydaliśmy 55%, a zakontraktowaliśmy 74%. To smutne, że państwo nie jesteście w stanie wydać tego, o co my zadbaliśmy, [[Dzwonek]] a boję się o to, co będzie w przyszłości. Poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.